Ponadto informuję, że w dniu dzisiejszym odbędzie się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Sportu Kobiet - o godz. 10.30. Komunikat.

Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania: - o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawartego między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r., - o poselskich projektach uchwał o solidarności w sprawie ochrony polskich granic oraz w sprawie politycznego oraz humanitarnego kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Sprawozdania to odpowiednio druki nr 1755 i 1774. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, marszałek Sejmu podjęła decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań. Marszałek Sejmu proponuje, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 3 regulaminu Sejmu oraz w dyskusjach nad tymi punktami porządku dziennego wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycje przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 16. porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Przypominam, że postawienie pytania nie może trwać dłużej niż 2 minuty, zaś udzielenie odpowiedzi nie może trwać dłużej niż 6 minut. Prawo do postawienia pytania dodatkowego przysługuje wyłącznie posłowi zadającemu pytanie. Dodatkowe pytanie nie może trwać dłużej niż 1 minutę, a uzupełniająca odpowiedź nie może trwać dłużej niż 3 minuty. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu odpowiedzi na pytanie dodatkowe. Proszę państwa, przechodzimy do pytań.

Posłowie Waldemar Andzel oraz Katarzyna Czochara z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zadadzą pytanie w sprawie elektronicznych rozwiązań dla obywateli. To pytanie będzie skierowane do prezesa Rady Ministrów, ministra cyfryzacji, a odpowie z upoważnienia prezesa Rady Ministrów sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pan minister Janusz Cieszyński. Bardzo proszę pana posła Waldemara Andzela o zadanie pytania. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Polacy dysponują szerokim pakietem elektronicznych rozwiązań dla obywateli. Bardzo proszę o wskazanie kluczowych portali i aplikacji służących do załatwienia spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Proszę również o przedstawienie, ile obecnie osób aktywnie korzysta z profilu zaufanego i innych rozwiązań. Panie ministrze, zapraszam pana uprzejmie i serdecznie do odpowiedzi na to treściwe, aczkolwiek krótkie pytanie. Wysoka Izbo! Panie Pośle! Dzisiaj jest ponad 13 mln obywateli korzystających z tej usługi. To jest usługa, która pozwala na wykorzystanie zdalnej tożsamości, czyli zidentyfikowanie się wobec usług administracji na odległość.

Można zalogować się też do usług Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez platformę usług elektronicznych - PUE ZUS.

Wszystkie usługi możecie państwo znaleźć na portalu RP - portalu gov.pl, który umożliwia ujednolicony sposób prezentacji informacji na wszystkich stronach rządowych.

Tych usług jest, tak jak mówię, bardzo dużo. Zachęcam wszystkich państwa do tego, żeby odwiedzać portal gov.pl i sprawdzać, jakie sprawy możemy załatwić przez Internet. Dziękuję serdecznie, panie ministrze. Pytanie dodatkowe zada pani poseł Katarzyna Czochara. Bardzo proszę, pani poseł. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie ministrze, mam dodatkowe pytanie. Mówił pan przed chwilą o tym, iż ministerstwo, rząd Zjednoczonej Prawicy pragnie rozwijać w dalszym ciągu tę tak ważną aplikację.

Proszę, panie ministrze. Wysoka Izbo! Pani poseł, to jest bardzo dobry przykład tego, jak możemy takie usługi cyfrowe rozwijać. To jest ustawa, którą prowadzi pan minister Paweł Szefernaker.

W związku z tym chcemy zaproponować operatorom telekomunikacyjnym zmianę formuły rozliczania za tę komunikację, tak żeby ona była zależna tylko od liczby abonentów, którzy mają taką możliwość, a nie od tego, ile wiadomości jest wysyłanych. Ta infrastruktura dla SMS-ów to jest bardzo często coś, co już od dawna funkcjonuje, często jest zamortyzowane, a koszty wysyłania kolejnych SMS-ów, ten koszt krańcowy zazwyczaj jest bliski zeru. Dlatego uważamy, że to jest dobry pomysł, dobry kierunek, żeby dążyć w stronę spopularyzowania tych usług, ale tak żeby zmienić model rozliczania, żeby polskie państwo w mniejszym stopniu musiało patrzeć na koszt wysyłki tych wiadomości jako na ograniczenie rozwoju usług. To umożliwi tworzenie takich rozwiązań, o których mówi pani poseł. Od strony technicznej, technologicznej to jest bardzo proste i na pewno do zrobienia w krótkim czasie, a zapotrzebowanie na taką i podobne temu usługi jest duże i będzie w mojej ocenie rosło. Dziękuję serdecznie. Panie ministrze, dziękuję za udział w obradach. Przechodzimy do następnego pytania. Posłowie Jarosław Gonciarz i Barbara Bartuś zadadzą pytanie w sprawie zmian w obowiązujących aktualnie symbolach narodowych. To pytanie jest skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Odpowie sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pan minister Jarosław Sellin, którego serdecznie witam. Bardzo proszę, pan poseł Jarosław Gonciarz, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Obecnie obowiązujące symbole państwowe Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy z 1980 r. Z kolei ostatnia zmiana w sferze symboli państwowych związana była ze zmianą ustroju w 1989 r. i przywróceniem godłu państwowemu korony. Od tego okresu otrzymywano wiele analiz oraz opinii, m.in. od heraldyków czy muzykologów, którzy wskazywali, że należy wprowadzić niezbędne zmiany i korekty. Nie mniej istotny wydaje się również kontekst cyfryzacji, gdyż potrzebne jest wprowadzenie wzorów symboli państwowych zgodnie ze współczesnymi technikami drukarskimi i graficznymi, co w ustawie z 1980 r. nie znajduje pokrycia. Ustawa z tego roku posiada oczywiście załączniki graficzne, jednak nie przystają one do dzisiejszych możliwości technicznych. Mając na względzie przywołaną przeze mnie konieczność wprowadzenia zmian, proszę o przybliżenie przygotowywanego projektu nowelizacji przepisów z zakresu symboli narodowych. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, zapraszam. Zapraszam pana z przyjemnością ze względu na naszą wspólną pracę 6-letnią kiedyś. Dziękuję, panie marszałku. Czuję wsparcie za plecami.

Bardzo dziękuję za to pytanie. Myślę, że jakaś dyskusja w domenie publicznej już się na ten temat toczy i warto rzeczywiście wskazać, jakie są główne cele tego zaproponowanego projektu ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej. To jest projekt opracowany przez nasze ministerstwo, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, i jak wskazuje uzasadnienie do tego projektu, ma na celu uporządkowanie stanu prawnego dotyczącego wykorzystywania przez instytucje państwowe, osoby prawne i fizyczne symboli państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, jak również wprowadzenie wzorów symboli państwowych zgodnych ze współczesnymi technikami drukarskimi i graficznymi. Obowiązująca ustawa ze stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych doczekała się wielu nowelizacji, ale pozostaje regulacją przestarzałą - to już 41 lat. Warto zaznaczyć, że wśród jej przepisów wykonawczych znajdują się nawet pochodzące z 1955 r., a więc sprzed 66 lat. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący użytkowania symboli państwowych przez administrację publiczną. Wskazywał on na pilną potrzebę modernizacji przepisów - 16 lat temu wskazano na pilną potrzebę modernizacji przepisów. Uznaliśmy, że trzeba się tego podjąć. Projekt ustawy porządkuje nazewnictwo symboli państwowych, w tym wprowadza rozróżnienie godła i herbu, bo dzisiaj w ustawodawstwie nie mamy tego rozróżnienia. Wskazuje w jasny sposób, które podmioty są uprawnione do używania flagi państwowej z herbem Rzeczypospolitej Polskiej, przywraca chorągiew Rzeczypospolitej jako symbol państwowy, a także zachęca do wywieszania flagi przez osoby fizyczne i prawne.

My chcemy tego ducha zmienić. Jednocześnie projekt stara się ograniczyć nadużywanie symboli państwowych w celach komercyjnych i na przedmiotach w obrocie handlowym. Podsumowując, można wskazać, że nowa regulacja całościowo zajmuje się kwestią użytkowania symboli państwowych. Dodatkowo przewidziane w ustawie rozporządzenie będzie stanowiło rodzaj kodeksu flagowego zawierającego wytyczne w sprawie postępowania z symbolami państwowymi. Obecna ustawa posiada załączniki graficzne, o tym pan poseł wspomniał, które nie przystają do dzisiejszych możliwości technicznych. Brak jest określonych w obecnych zestandaryzowanych systemach graficznych barw narodowych w zdefiniowanej ustawowo wersji cyfrowej godła oraz wizerunku orła Rzeczypospolitej Polskiej. W praktyce oznacza to, że ochrona symboli państwowych nie jest możliwa. Większość używanych dzisiaj flag i godeł nie odpowiada wymogom nawet obecnej ustawy. Współrzędne barw określone w ustawie zostały wskazane w systemie CIELUV, mało przydatnym dla potrzeb grafiki cyfrowej i nieprzekładalnym w prosty sposób na inne systemy. Utrudniało to także tworzenie jednolitej identyfikacji wizualnej państwa i jego urzędów, na co zwracano wielokrotnie uwagę.

Wszędzie tam starano się przyjmować nowoczesne ustawodawstwo dotyczące symboli państwowych.

W opinii ministerstwa nowa regulacja dostosowuje w pełni symbole państwowe do nowych technologii cyfrowych, umożliwiając przez to ich właściwą ochronę. Przepisy przejściowe ustawy zakładają długi okres wdrożenia projektowanej regulacji w celu obniżenia kosztów ponoszonych przez budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. Łączne koszty w okresie 10 lat oszacowano na 147 mln zł - 10 lat. Nie przewidziano obowiązku wymiany dokumentów, mundurów, druków, uznając, że będą wycofywane po ich zużyciu. Pozwala to w praktyce na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z wdrożeniem tej ustawy. Dziękuję bardzo. Pytanie dodatkowe zada pani poseł Barbara Bartuś. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze!

Ustalenie barw, numerów zgodnie z obowiązującymi możliwościami jest konieczne. Ta nowelizacja jest też bardzo, bardzo szeroko komentowana, m.in. moje lokalne media się o tym rozpisywały. Chciałabym więc zapytać, panie ministrze, jak przedstawiają się konsultacje, bo projekt ten jest w konsultacjach.

Dziękuję bardzo. To ciekawe pytanie, panie ministrze. Niech pan odpowie, dlaczego Bonaparte był wcześniej niż potop szwedzki. Bo ja nie mam. Rozumiem, panie marszałku, że były dwa pytania. Pani poseł, postaram się na oba odpowiedzieć, jeżeli starczy mi czasu. Szanowna Pani Poseł!

Uwagi zgłosiło 95 organizacji i osób fizycznych. Dla potrzeb raportu z konsultacji społecznych zostanie opracowana szczegółowa statystyka z podziałem na rodzaj uczestników i na tematy poruszane w tych uwagach. Uznaliśmy, że uwzględnione zostaną wszystkie uwagi, które dotrą do nas przed 5 listopada br. Uwagi zostały ułożone według tematów, a nie uczestników, co dało łącznie 285 uwag. Chcę bardzo mocno podkreślić, że żadna z uwag, a było ich wiele, jak powiedziałem, nie przeczy potrzebie opracowania nowej ustawy zastępującej obecnie obowiązujące przepisy, których część powstała w 1980 r. lub wcześniej.

Głównym celem tej ustawy było dopasowanie możliwości, można powiedzieć, kodyfikowania naszych symboli narodowych, państwowych zgodnie z najnowocześniejszymi technikami po pojawieniu się Internetu i różnych grafik w przestrzeni wirtualnej, ale oczywiście są też w tej ustawie uwagi czy pomysły, które najbardziej absorbują opinię publiczną.

Jednocześnie chcę jasno zadeklarować, że jeżeli w ramach konsultacji publicznych albo dominującego głosu reprezentacji narodu, jakim jest parlament Rzeczypospolitej, uznamy, że nie ma sensu w tym grzebać, to tak zrobimy.

Ale nie będziemy się przy tym upierać. Dziękuję bardzo, panie ministrze, za to elastyczne podejście do hymnu polskiego. Proszę państwa, przechodzimy do następnego pytania. Posłowie Agnieszka Hanajczyk oraz Adam Szłapka zadadzą pytanie w sprawie wydarzeń o charakterze antysemickim, nawołujących do przemocy i dyskryminacji ze względu na narodowość, wyznanie i orientację seksualną, mających miejsce w Kaliszu 11 listopada 2021 r. To pytanie będzie skierowane do ministra sprawiedliwości, a odpowie na nie zastępca prokuratora generalnego pan Krzysztof Sierak. Bardzo proszę panią poseł Agnieszkę Hanajczyk o zadanie pytania. Panie Marszałku! Panie Prokuratorze! Wysoka Izbo! Wieszanie na szubienicy zdjęć europosłów, sprawa Jacka Międlara, brylujący, mocno dofinansowany ze środków publicznych Robert Bąkiewicz, marsze narodowościowe w 2020 r., w 2019 r., hasła „Śmierć lewackiej...” - tutaj z mównicy nie dokończę - i ostatnie wydarzenia, wydarzenia w Kaliszu, będące kwintesencją ksenofobii, antysemityzmu, faszyzmu. To już nie jest kategoria narracji skandalicznego spektaklu. Wszystkie te wydarzenia łączy. No właśnie, panie prokuratorze, co łączy? Bezradność, niemoc czy przeciwnie, ciche przyzwolenie wymiaru sprawiedliwości na takie zachowania? Czy minister Ziobro, czy ministerstwo nie widzi potrzeby delegalizacji organizacji szerzących faszyzm?

Dlaczego Olszański w sobotę jeszcze raz wystąpił publicznie w Kaliszu i nikt temu nie zapobiegł?

Dziękuję bardzo. Panie prokuratorze, bardzo proszę.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że przestępstwa z nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych i z powodu bezwyznaniowości są ścigane przez prokuraturę z pełną determinacją, a postępowania przygotowawcze prowadzone w tych sprawach pozostają przedmiotem stałego zainteresowania Prokuratury Krajowej. Jeżeli chodzi o działania prokuratury w związku ze zdarzeniem mającym miejsce w dniu 11 listopada w Kaliszu podczas wiecu zorganizowanego przez Wojciecha O., Marcina O., prokuratura działała tutaj bez względnej zwłoki oraz według wszelkich zasad Kodeksu postępowania karnego. Dowody tego działania prokuratury - bardzo szybkiego, bezzwłocznego - to kalendarium, które przedstawię Wysokiej Izbie. W piątek 12 listopada do Prokuratury Rejonowej w Kaliszu wpłynęło pismo Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przesyłające notatkę urzędową wraz z nagraniem audio-wideo oraz protokołem oględzin płyty ze sporządzonym stenogramem z przebiegu wiecu zorganizowanego w dniu 11 listopada w Kaliszu przez Wojciecha O., Marcina O., przy udziale Piotra R., celem zapoznania się oraz podjęcia decyzji co do dalszych czynności w sprawie. Chcę tu zaznaczyć, że Policja nie podjęła z własnej inicjatywy żadnych czynności, o jakich mowa w art. 308 Kodeksu postępowania karnego, które mogła podjąć jeszcze w trakcie trwania wiecu lub bezpośrednio po jego zakończeniu, skoro z bieżących policyjnych obserwacji wynikałoby, że zachowania określonych osób wyczerpywałyby znamiona przestępstw publicznoskargowych. W tym samym dniu, w piątek 12 listopada, do Prokuratury Rejonowej w Kaliszu wpłynęło także zawiadomienie prezydenta miasta Kalisza wskazujące na podejrzenie popełnienia przestępstw z nienawiści skierowanych przeciwko ludności żydowskiej podczas zorganizowanego dzień wcześniej wiecu. W dniu 13 listopada, czyli w sobotę, prokurator Prokuratury Rejonowej w Kaliszu wszczął śledztwo w sprawie publicznego nawoływania w dniu 11 listopada br. w Kaliszu do nienawiści na tle wyznaniowym i różnic narodowościowych oraz znieważenia grupy ludzi z uwagi na ich wyznanie, przynależność narodową, tj. o czyn z art. 256 § 1 Kodeksu karnego i art. 257 Kodeksu karnego, zaś prowadzone śledztwo powierzył w całości Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu. Jeszcze w tym samym dniu, w sobotę 13 listopada, prokurator zapoznał się z zapisami nagrań dostarczonymi przez Policję. Polecił KMP w Kaliszu wykonanie oględzin i sporządzenie stenogramów i innych nagrań zarejestrowanych podczas wiecu i marszu oraz polecił przesłuchanie do dnia następnego, czyli do 14 listopada, ewentualnych świadków. W dniu 14 listopada, w niedzielę, prokurator po zapoznaniu się z uzupełnionym materiałem dowodowym wydał postanowienia o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu do prokuratury Wojciecha O., Marcina O., Piotra R., które to czynności zlecił do wykonania Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu.

W tym samym dniu, w poniedziałek, prokurator ogłosił zarzuty wszystkim trzem zatrzymanym mężczyznom i przesłuchał ich w charakterze podejrzanych. Po wykonaniu czynności procesowych z podejrzanymi w dniu 15 listopada prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Kaliszu wniosek o zastosowanie wobec nich środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, uznając, że zachodzi uzasadniona obawa ucieczki i ukrywania się podejrzanych oraz obawa nakłaniania do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień pozostałych osób, których zachowanie podczas wiecu także wyczerpywało znamiona przestępstwa, a których tożsamości do chwili obecnej jeszcze nie ustalono, a tym samym nie wykonano dotychczas czynności procesowych z ich udziałem. W dniu wczorajszym późnym wieczorem Sąd Rejonowy w Kaliszu uwzględnił wnioski prokuratora i zastosował wobec podejrzanych Wojciecha O., Marcina O. i Piotra R. środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd w pełni podzielił tu argumentację prokuratora co do potrzeby stosowania izolacyjnych środków zapobiegawczych. Odnosząc się do pytania pani poseł w sprawie tych nieprawdziwych publikacji - powtarzam: nieprawdziwych publikacji - o rzekomym blokowaniu przez prokuratora czynności Policji w trakcie zgromadzenia w Kaliszu 11 listopada. chciałbym tutaj, panie pośle, stanowczo, jednoznacznie stwierdzić, że nieprawdziwe są informacje, jakoby prokurator zakazał Policji zatrzymywać uczestników zgromadzenia w Kaliszu 11 listopada br. Prokurator nie wydał Policji takich poleceń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami decyzję o zatrzymaniu osoby w takich sytuacjach, czyli na gorącym uczynku lub bezpośrednio po nim, podejmuje samodzielnie Policja, która dopiero po zatrzymaniu niezwłocznie (Dzwonek) informuje o tym prokuratora.

Dziękuję bardzo. Pytanie dodatkowe zada pan poseł Adam Szłapka. Panie Marszałku! Na początek warto przypomnieć, za każdym razem warto przypominać, że pan Mateusz Morawiecki jest kłamcą skazanym dwukrotnie wyrokiem sądu za kłamstwo. Panie Prokuratorze!

To nie jest przypadek, że oni się czują rozzuchwaleni, tylko to jest wasza przemyślana polityka. Chcę zapytać bardzo konkretnie: Czy w prokuraturze są jakieś wytyczne co do pobłażliwego traktowania kwestii mowy nienawiści, antysemityzmu? Wie pan, co mi odpisała prokuratura? Tak działa prokuratura. Pamiętam, kiedy na stadionie warszawskiej Legii był napis: Nowoczesna, KOD, Lis, Olejnik - dla was będą szubienice. Prokuratura też nie dopatrzyła się w tym żadnego znamiona przestępstwa. Doprowadziliście do tego, że antysemici, ludzie, którzy doprowadzają do przestępstw z nienawiści, są bezkarni, bo czują się bezkarni, bo Piotr R. to jest wasz kolega. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, panie prokuratorze.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zdumiony jestem pytaniami. Nie ma w prokuraturze żadnej ulgowej procedury dla kogokolwiek, tym bardziej dla przestępców, którzy nawołują do nienawiści. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, panie pośle. Oczywiście zapoznam się z tymi materiałami. Na pewno ustosunkuję się do tego pytania.

W prokuraturach okręgowych i regionalnych oraz w Departamencie Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej prowadzony jest pełny monitoring spraw tej kategorii, w następstwie czego większość tych postępowań - powtarzam: większość tych postępowań - jest obejmowana zwierzchnim nadzorem służbowym celem zapewnienia ich prawidłowego przebiegu, w tym uniknięcia przez prokuratorów w rejonach czy w prokuraturze okręgowej odmawiania wszczęcia lub też umarzania z powodu czy to znikomej społecznej szkodliwości czynów, czy to czasami badania tych spraw pod tym kątem, gdy prokurator umarza sprawę ze względu na brak znamion czynu zabronionego.

Dane są analizowane przez prokuratorów, koordynatorów tego problemu i raz czy dwa razy w roku, o ile pamiętam, ukazuje się to sprawozdanie na stronie Prokuratury Krajowej. Prokuratura podchodzi z pełnym zaangażowaniem do wszelkiego rodzaju przestępczości, tym bardziej do tej przestępczości, która budzi takie zainteresowanie społeczeństwa. Dziękuję bardzo.

Bardzo proszę pana marszałka, żeby uniemożliwił i potępiał mowę nienawiści ze strony posłów, którzy tutaj oszukują, kłamią i którzy szkalują premiera Rzeczypospolitej oraz ministrów Rzeczypospolitej. Ci sami ludzie, wtedy, kiedy dziennikarze „Faktu” publikowali informacje, że gotowi są mnie zamordować za milion złotych, milczeli.

Panie pośle. Pozwalam posłom na wypowiedzi, tak jak panu. Chociaż regulamin w tej sprawie zakazywałby takich rzeczy, pozwoliłem zabrać głos. A teraz pozwolę zabrać głos panu posłowi Szłapce, gdyż pan go wywołał.

Pan premier Morawiecki w kampanii wyborczej został dwukrotnie skazany za mówienie nieprawdy. Jest po prostu kłamcą. I jest na to potwierdzenie, wyrok sądu. Przechodzimy, proszę państwa, do następnego pytania.

Pytanie będzie dotyczyło działań podjętych przez Centralne Biuro Śledcze i Prokuraturę Krajową w sprawie udziału lokalnych polityków z Bogatyni i powiatu zgorzeleckiego w zorganizowanym wyłudzaniu środków publicznych oraz udziału tych osób w procederze produkcji i dystrybucji amfetaminy. To pytanie jest skierowane do prezesa Rady Ministrów, a odpowie z upoważnienia prezesa Rady Ministrów zastępca prokuratora generalnego, znany już nam pan prokurator Krzysztof Sierak, który odpowiadał na poprzednie pytanie. Bardzo proszę panią posłankę Katarzynę Kretkowską o zabranie głosu. Wysoka Izbo!

Większość zatrzymanych to prominentni działacze lokalnego PiS. Pytanie, dlaczego dotąd nie ma aktu oskarżenia wobec żadnej z osób zatrzymanych na podstawie śledztwa CBŚ i prokuratury.

Konflikt i odwlekanie ugody z Czechami, jak się okazuje, także mają podłoże w tych samych korupcyjnych układach. Bo domagają się niezależnych ekspertów. A czemu PiS ich nie chce?

Dziękuję serdecznie. Zapraszam panią posłankę Małgorzatę Sekułę-Szmajdzińską. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Dodaję tylko do tego, co przed chwilą powiedziała koleżanka, że jest mi bardzo przykro, że Bogatynia, w tym jej dzielnica Turoszów, stała się w Polsce popularna z powodu kłopotów, jakie dotknęły to miasto i gminę. Ja zresztą rozmawiam z mieszkańcami, pytam ich, czy wiedzą, co się dzieje ze sprawą afery korupcyjno-gangsterskiej, i słyszę jedno: cisza, nic się nie dzieje. My, posłowie, mamy prawo wiedzieć, jakie działania podejmują organy państwa do tego powołane. Ja po prostu naprawdę nie mogę już słuchać tego, że mieszkańcy mówią: a, ludzie sobie chodzą po ulicy, ci, którzy powinni w kryminale siedzieć.

Dziękuję serdecznie. Panie prokuratorze, zapraszam pana bardzo grzecznie. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odpowiadając na pytanie dotyczące działań podjętych przez Policję, Centralne Biuro Śledcze i Prokuraturę Krajową w sprawie udziału lokalnych polityków Bogatyni i powiatu zgorzeleckiego w zorganizowanym wyłudzaniu środków publicznych oraz udziału tych osób w procederze produkcji i dystrybucji amfetaminy, uprzejmie informuję, iż powyższe okoliczności są przedmiotem śledztwa prowadzonego przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

W powyższym śledztwie są dwa zasadnicze wątki.

Drugi z głównych wątków śledztwa skoncentrowany jest na zdarzeniach dotyczących tzw. przestępczości urzędniczej i obejmuje osoby piastujące w powiecie zgorzeleckim, głównie w gminie Bogatynia, funkcje i stanowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia i spółkach komunalnych. Osoby te miały dopuszczać się czynów zabronionych polegających na przyjmowaniu i żądaniu korzyści majątkowych w związku z pełnionymi funkcjami i zajmowanymi stanowiskami, nie dopełniały obowiązków i nie wykonywały swoich uprawnień, poświadczały nieprawdę w dokumentach, w tym także miało dochodzić do wielu nieprawidłowości w zakresie działania Urzędu Miasta i Gminy Bogatyni, związanych m.in. z przeprowadzaniem przetargów.

Rola Daniela F. polegała w szczególności na wykorzystywaniu swoich uprawnień i znajomości do udostępniania członkom zorganizowanej grupy przestępczej pomieszczeń i miejsc, w których miały być wytwarzane substancje psychotropowe. Miał on także ułatwiać i organizować przedsięwzięcia związane z inwestycjami członków zorganizowanej grupy, z uzyskiwaniem środków finansowych. Inny wątek, trzeci, to przestępstwa w zakresie gospodarki odpadami.

Na mocy tej ustawy wprowadzono obowiązek składowania odpadów zastrzeżonej kategorii tylko w regionalnych instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych.

Ustalono, że osoby reprezentujące Urząd Miasta i Gminy Bogatynia oraz Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. dążyły do unikania konieczności ponoszenia opłat za odbieranie, składowanie i przetwarzanie odpadów zastrzeżonej kategorii.

Inny wątek omawianego śledztwa dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa otwartego kąpieliska w Bogatyni”

Szanowni Państwo! To nie jest tak, że śledztwo stoi w miejscu.

Czyny te jednak nie zostały popełnione z udziałem lokalnych polityków z Bogatyni i powiatu zgorzeleckiego. Występuje w niej aktualnie 53 podejrzanych, którym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej z art. 258, popełnienia przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przyjmowania korzyści majątkowych z art. 228 k.k., przekraczania uprawnień, niedopełniania obowiązków z art. 231 k.k., poświadczania nieprawdy - tak jak wcześniej opowiadałem - w dokumentacji z art. 271, przywłaszczania mienia, oszustwa, niegospodarności.

Dziękuję uprzejmie. Pytania dodatkowe. Widzę tu w kolejności: pan poseł Marek Dyduch i pan poseł Robert Obaz.

To jak uważacie. Bardzo proszę. Nie ma problemu z kolejnością. Natomiast jest pytanie do prokuratury. Przecież władza jest pełniona w określonym czasie.

Jak funkcjonuje tu relacja organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości do pełnionej władzy? Dziękuję. Proszę państwa, została sekunda, ale ponieważ przedłużyłem panu prokuratorowi, bo to są sprawy prokuratorskie, więc nie widzę sensu, powiem szczerze, po pytaniach skracać wypowiedzi, bo są różne rodzaje pytań. To jest bardzo konkretne, a pan prokurator też odpowiada konkretnie. Proszę o zadanie pytania. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Prokuratorze! Opowiadał pan o tym dużo, to był rok 2018, kiedy nastąpiły te aresztowania. Tak naprawdę to cała wierchuszka Prawa i Sprawiedliwości, wszystkie te osoby, które fotografowały się z prezesem Jarosławem Kaczyńskim.

W ogóle nie było widać, że ma jakiekolwiek obawy, że zostanie skazany.

Kiedy możemy liczyć na to, że te osoby zostaną skazane? Zapraszam pana prokuratora. Szanowny Panie Marszałku! Jeżeli chodzi o śledztwa z zakresu zorganizowanej przestępczości, szczególnie tak rozbudowane, rozległe, jak sami państwo widzicie, jak to ujmujecie, że cała wierchuszka bądź w zasadzie wszyscy funkcjonujący w Bogatyni to przestępcy, to nie da się takiego śledztwa skończyć w rok, dwa, mając na uwadze konieczność wykonania czynności, a szczególnie, jeżeli jest to powiązane z przestępczością i kryminalną, i ekonomiczną, i wynikającą z założeń korupcyjnych. Trudno mi odpowiedzieć na pytanie odnoszące się do pana Sławomira Z., który jest spokojny o wyrok. Nie wiem, czy będzie tak spokojny, jeżeli sprawa zostanie skończona i zostanie skierowany akt oskarżenia do sądu. Trudno mi powiedzieć, czy wtedy pan Sławomir Z. będzie spokojny. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, również nie mogę się odnieść do tego, kiedy prokuratura dowiedziała się o tych zdarzeniach, gdyż nie znam takich szczegółów. Jeżeli mogę prosić o pytania na piśmie, to na pewno prokurator referent odniesie się do tej kwestii. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie prokuratorze. Przechodzimy do następnego pytania. Pan poseł Zbigniew Ziejewski z Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska zada pytanie w sprawie walki z afrykańskim pomorem świń. To pytanie jest skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, a odpowie w imieniu ministra sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan minister Szymon Giżyński. Panu prokuratorowi bardzo serdecznie dziękuję za odpowiedzi. Miło, że pan nas odwiedził. Bardzo proszę, panie pośle. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Od początku roku potwierdzono już 2422 ogniska ASF-u dzików i 119 ognisk ASF-u świń. Od dawna alarmujemy o podjęcie pilnych działań ochronnych, o pomoc dla producentów trzody chlewnej, o należne rekompensaty. Niestety bez efektu. Sytuacja rolników zajmujących się trzodą chlewną z każdym dniem jest coraz gorsza. Walka z ASF jest dla nowego ministra rolnictwa priorytetem.

Chciałbym poznać wyniki tych rozmów. Pytanie drugie. Producenci rolni prowadzący chów i hodowlę świń na obszarach z ograniczeniami mogą ubiegać się o nieoprocentowane pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań. Pieniądze się skończyły, pożyczek brak. Czy będą nowe i kiedy? Rolnicy, u których wybuchły ogniska, ich sąsiedzi, którym wybito trzodę chlewną, czekają na wznowienie produkcji. Czy za okres postoju mogą liczyć na rekompensaty? Kilka miesięcy nie mają już wstawionych świń, a opłaty są - co z nimi? Czy i kiedy nastąpi zmiana zasad udzielania pomocy na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń? Nowe zasady nie uwzględniają gospodarstw, w których zmieniono profil produkcji. Pytanie piąte, ostatnie. Na posiedzeniu podkomisji dotyczącej ASF-u ustalono, że w siedmiu powiatach w Polsce, w których produkcja przekracza (Dzwonek) 150 tys. sztuk, nastąpi bardzo silna depopualcja dzików, m.in. jest tak w Iławie i Nowym Mieście Lubawskim. Jakie są zalecenia dla łowczych w tych powiatach? Dziękuję. Panie ministrze, zapraszam.

Nie dlatego, że te pytania resort przerażają czy mam tutaj coś do ukrycia albo boimy się tego typu pytań. One są szczegółowe.

Czy program odbudowy gospodarstwa po ASF faktycznie działa i czy rolnicy otrzymują wystarczające wsparcie finansowe?

I myślę, że to musi pana posła zaspokoić przynajmniej w tej mierze, natomiast na całą piątkę tych pytań oczywiście odpowiemy na piśmie, bo to w każdej chwili jest oczywiste i dopuszczalne. A więc odpowiadam na pytanie pierwsze, przesłane zgodnie z procedurą. Ile obecnie wynosi liczba stad trzody chlewnej i o ile zmalała w stosunku rok do roku?

Później liczba stad malała.

To są oczywiście gołe liczby, które każdy z nas tutaj na pewno w bardzo podobny sposób będzie interpretował, ale ta tendencja nie może szokować czy dziwić. Ważne jest to, że liczba świń się utrzymuje, natomiast liczba stad jest uzależniona w tym procesie od postępów i od sytuacji bioasekuracyjnych. Jest najzupełniej oczywiste, że rygory bioasekuracji w jakimś sensie wysuwają do przodu - i tak było we wszystkich państwach, które także to przechodziły przed nami, np. w Hiszpanii - wysuwają na czoło te gospodarstwa, które są w stanie w tej konkurencyjnej walce podołać coraz wyższym wymogom bioasekuracji. Bo takie są realia walki z chorobą, inaczej być nie może.

To jest sytuacja obiektywna.

Ale jednocześnie pozostaje ona rynkowo wielką, ogromną potęgą.

Pytanie drugie: Czy program odbudowy gospodarstw po ASF faktycznie działa i czy rolnicy otrzymują wystarczające wsparcie finansowe?

Rolnicy złożyli w tym czasie 776 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę 385 mln zł. Zakontraktowano prawie 5 tys. wniosków na kwotę 225 mln zł oraz wypłacono 115 mln zł dla 2370 beneficjentów.

Proszę bardzo.

Dziękuję bardzo. Sprawdzamy to w tej chwili. Zaraz będziemy wiedzieli, czy ministerstwo pracuje nad tym czy dopiero będzie pracowało.

Pomoc jest ulokowana w tylu miejscach, że musiałem się upewnić, że udzielę prawidłowej odpowiedzi na pytanie zgodnie z intencjami pana posła. Pomoc dla producentów świń, w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, jest w tej chwili na poziomie, który będziemy systematycznie rozszerzać. Bo jest to pomoc do 50 sztuk w stadzie i oznacza to 36 gr dziennie za sztukę.

Prace idą w tym kierunku. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Przechodzimy do następnego pytania, które będą zadawali posłowie Grzegorz Lorek oraz Krzysztof Janusz Kozik z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Będzie to pytanie w sprawie stanowiska Polski na szczycie klimatycznym. Odpowie podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pan minister Adam Guibourgé-Czetwertyński. Bardzo proszę pana posła Grzegorza Lorka o zadanie pytania pierwszego. Dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Za nami kolejny szczyt klimatyczny. Nasz kraj w minionych dekadach zrobił bardzo wiele w sprawie ograniczenia emisji i jesteśmy w Europie emitentem nawet niecałego 1%. Chciałbym powiedzieć, że Niemcy to ponad 2%, Chiny to jest prawie 35%. Chciałbym się zapytać o stanowisko Polski zaprezentowane na szczycie klimatycznym w Glasgow.

Chciałbym dopytać też o kwestie związane z czystymi technologami, z wychwytem i przetwarzaniem CO2. Bo myślę, że nam wszystkim: zarówno ekologom spod znaku pani Grety Thunberg, jak i mnie, środowisku, które reprezentuję, czyli górników i energetyków, zależy na czystym powietrzu, na ograniczeniu emisji.

Bo jak wiadomo, od tego gazu nie da się uciec. To jest gaz, który nam towarzyszył od samego początku ludzkości, a nawet i wcześniej, więc myślę, że musimy się przyzwyczaić do życia z tym gazem. Możemy też starać się poprzez metody techniczne, jak również naukę, która nam w tym powinna pomagać, ograniczać oddziaływanie CO2 na klimat. Chciałbym zapytać, czy tu również w tym obszarze polski rząd będzie realizował przedsięwzięcia. Dziękuję. Bardzo proszę, panie ministrze. Bezpośrednio po pana odpowiedzi przejdziemy do następnego pytania. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Z naszego punktu widzenia najważniejsze jest pewnie dokończenie zasad katowickich, wdrażania porozumienia paryskiego.

Udało się równocześnie uzgodnić tabelę, formaty raportowania dla wszystkich stron, które zapewnią przejrzystość i porównywalność działań na poziomie globalnym.

Chodzi też o rosnącą świadomość, że polityka klimatyczna musi być prowadzona w taki sposób, który nie wygeneruje dodatkowych obciążeń dla społeczeństwa, w szczególności dla najuboższych gospodarstw domowych, w szczególności dla regionów, dzisiaj najbardziej uzależnionych od wydobycia paliw kopalnych.

Takim źródłem jest np. energetyka atomowa, która zapewnia stabilne dostawy energii przy braku emisji CO2. To się nie może wydarzyć tak od razu.

Nad takimi rozwiązaniami pracujemy w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Przechodzimy do następnego pytania.

To pytanie skierowane jest do prezesa Rady Ministrów, który upoważnił do odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych pana ministra Macieja Małeckiego. Super mi to poszło. Wysoka Izbo! Na początku powiem, że bardzo żałuję, że na to pytanie odpowiadać będzie pan minister reprezentujący Skarb Państwa, a nie pan premier Mateusz Morawiecki, bo w sprawie Turowa, w sprawie tego, co dzieje się w Bogatyni. Tak naprawdę ta sprawa skupia w sobie wszelkie patologie rządu PiS. Mówimy tu o głupocie, nepotyzmie, korupcji, aferach. Chwilę temu pan prokurator, zastępca prokuratora krajowego mówił o tym, że działa tam zorganizowana grupa przestępcza.

Tragedią w tej całej sytuacji jest to, panie ministrze, że za tę niekompetencję, za te afery, za tę zorganizowaną grupę przestępczą, jak mówił zastępca prokuratora krajowego, płacą Polacy. Przecież codziennie płacimy gigantyczne kary za Turów.

Co robi prokuratura w tej sprawie? Czy ktoś poniósł konsekwencje? Czy ktoś został zwolniony? Czy wy jako rząd polski, jako resort, który nadzoruje Skarb Państwa, skierowaliście chociaż jedną sprawę do prokuratury? Wygląda na to, że nie robicie kompletnie nic, że pozwalacie, aby ten problem narastał, że pozwalacie na to, żeby Polacy płacili za waszą niekompetencję. Będą płacić, bo kwestia dotyczy strategicznego obszaru działania państwa. To nie jest pierwsza tego typu sprawa. Kiedy wreszcie zaczniecie wyciągać wnioski? Dziękuję bardzo. Zapraszam, panie ministrze. Pan minister Maciej Małecki. Bardzo proszę. Wysoka Izbo!

W wyniku tego nastąpiło osunięcie znacznych ilości mas ziemnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda kopalnia węgla brunatnego, w tym także kopalnia Turów, prowadzi roboty górnicze na podstawie planu ruchu i dokumentacji technicznej kształtowania zwałowiska. Plan ruchu zakładu górniczego podlega zatwierdzeniu przez dyrektora okręgowego urzędu górniczego. Dokumentacja techniczna kształtowania zwałowiska jest dokumentem wewnętrznym i musi być zgodna z zatwierdzonym planem ruchu. Dokumentacja ta jest kontrolowana przez dyrektora okręgowego urzędu górniczego. Zgodność prowadzenia robót górniczych z zatwierdzonymi dokumentami, czyli planem ruchu i dokumentacją techniczną kształtowania zwałowiska oraz projektami technicznymi, a także cyklicznymi ocenami eksperckimi stanu zwałowiska, jest kontrolowana kilka razy do roku przez Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu i Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach. Przyczyny powstania zdarzenia miały wielowymiarowy charakter i wzajemnie na siebie oddziaływały. W celu zbadania przyczyn i skutków osuwiska w Turowie Polska Grupa Energetyczna powołała komisję, której zadaniem była analiza okoliczności i przyczyn powstania tego zdarzenia geotechnicznego, a prezes Wyższego Urzędu Górniczego powołał zespół doradczo-opiniujący do analizy niektórych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego w Turowie. Natychmiast, jeszcze tego samego dnia, powołany został sztab akcji ratowniczej pod przewodnictwem dyrektora oddziału. Ten sztab prowadził czynności bezpośrednio związane z działaniami ratowniczymi w celu minimalizacji skutków zdarzenia, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego zdrowia i życia ludzi oraz majątku przedsiębiorstwa. Równolegle pracował zespół zagrożeń naturalnych, do którego oprócz służb z kopalni powołano również ekspertów zewnętrznych. Zespół służył jako ciało doradcze sztabu akcji. Po zakończeniu akcji ratowniczej i wygaśnięciu ruchów osuwiskowych 3 października 2016 r. powołana została komisja, której zadaniem było dokonanie analizy okoliczności i przyczyn powstania zdarzenia geotechnicznego na zwałowisku wewnętrznym w kopalni węgla brunatnego w Turowie. Na potrzeby prac komisji sporządzono szereg niezależnych ekspertyz z dziedziny geotechniki i hydrologii, których zadaniem było wskazanie okoliczności i przyczyn powstania osuwiska. Wykonawcami tych ekspertyz były Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Wrocławska, Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze przy AGH. W celu kontroli poprawności zastosowanych rozwiązań technicznych oraz działania służb w kopalni Turów PGE GiEK zlecił AGH wykonanie audytu. AGH w listopadzie 2017 r. wykonała dokumentację pt. ekspertyza w zakresie rozwiązań technicznych stosowanych w zakładzie górniczym Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. Nie stwierdzono zaniedbań, które mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu zakładu górniczego, oraz nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzeń z nimi związanych. Dobór rozwiązań technicznych również został oceniony pozytywnie. Zespół, którego zadaniem było m.in. wyjaśnienie okoliczności i przyczyn powstania katastrofy, zakończył swoje działanie 14 czerwca 2019 r. i ocenił, że pomimo prowadzenia zwałowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i najlepszą wiedzą techniczną Stanowisko zespołu było zbieżne z wynikami szeregu ekspertyz w tym zakresie. Również organy nadzoru górniczego prowadziły działania wyjaśniające. Dyrektor okręgowego urzędu górniczego rozpoczął kontrolę prowadzenia ruchu zakładu oraz sprawował nadzór nad działaniami sztabu akcji ratowniczej w kopalni Turów. Dyrektor okręgowego urzędu górniczego wydał szereg decyzji dotyczących wstrzymania ruchu zakładu w obszarze objętym osuwiskiem oraz działań zabezpieczających ruch zakładu górniczego na obszarze nieobjętym osuwiskiem. Nakazał również wykonanie dodatkowego rozpoznania i analiz z zakresu geologii i geotechniki.

Do zadań zespołu należały weryfikacja zasad prowadzenia robót górniczych na terenie zwałowiska wewnętrznego w Turowie należącego do PGE, przygotowanie opinii w zakresie możliwości bezpiecznego prowadzenia robót w rejonie miejsca zdarzenia. W wyniku prac powstała opinia w sprawie możliwości bezpiecznego prowadzenia robót na terenie zwałowiska wewnętrznego w Turowie w rejonie osuwiska, które miało miejsce we wrześniu 2016 r. Eksperci z Wyższego Urzędu Górniczego wydali także zalecenia w celu zapobieżenia podobnym wypadkom w przyszłości. Zalecenia zespołu Wyższego Urzędu Górniczego były generalnie zbieżne z zaleceniami naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Wrocławskiej, którzy wykonywali dokumentację określającą przyczyny powstania osuwiska oraz dalsze wytyczne do eksploatacji. Podkreślam: wszystkie zalecenia komisji powołanej przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego zostały wypełnione, a ich realizacja była monitorowana przez dyrektora (Dzwonek) Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Orzeczenie zawiera ponadto wnioski zmierzające do zapobieżenia podobnym wypadkom w przyszłości.

Dziękuję bardzo. Pytanie dodatkowe zada pani poseł Zofia Czernow. Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Bardzo szybko i krótko pan minister wyjaśnił sprawę katastrofy w kopalni, ale chciałam dopytać, bo tę katastrofę bardzo skrzętnie ukrywano przed społeczeństwem, a zdarzyło się tam bardzo dużo złego. Czy określono przyczyny katastrofy? Kto zawinił i kto poniósł konsekwencje?

Ta sprawa w moim przekonaniu nie (Dzwonek) została dogłębnie zbadana i powinny się tym zająć prokuratura i Najwyższa Izba Kontroli. serdecznie, pani poseł. Zapraszam pana ministra.

Wysoka Izbo!

W tym okresie Polska Grupa Energetyczna prowadziła bardzo transparentną politykę komunikacyjną, wszystkie komunikaty informacyjne były wysyłane także bezpośrednio na skrzynki mailowe do dziennikarzy, którzy byli zainteresowani tą sprawą. 29 września 2016 r., czyli 2 dni po powstaniu osuwiska, w kopalni Turów została zorganizowana konferencja prasowa z udziałem ówczesnych władz spółki PGE GiEK oraz dyrektora kopalni Turów. Podczas tej konferencji udzielano odpowiedzi na wiele pytań dziennikarzy. Co więcej, informacje o osuwisku były publikowane w raportach giełdowych i w rocznym sprawozdaniu finansowym grupy PGE za rok 2016 oraz w sprawozdaniu zarządu PGE GiEK też za 2016 r. Te dokumenty są powszechnie dostępne.

Sytuacja na rynku cen energii elektrycznej jest wypadkową działań tych radykalnych obostrzeń klimatycznych przyjmowanych przez Komisję Europejską. Realizacja tych planów klimatycznych będzie skutkowała zubożeniem społeczeństwa, utratą miejsc pracy w całej Unii Europejskiej. A przypomnę, że partią dominującą w Parlamencie Europejskim jest Europejska Partia (Dzwonek) Ludowa, na czele której stoi Donald Tusk, a tworzą ją m.in. europosłowie Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Przechodzimy do następnego pytania. Posłowie Mariusz Trepka oraz Andrzej Gawron z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zadadzą pytanie w sprawie projektu Legia Akademicka. Na to pytanie odpowie pan minister Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Bardzo proszę, pan poseł Mariusz Trepka. Panie Marszałku! Panie Ministrze!

Jest to bardzo ciekawy projekt skierowany do studentów zainteresowanych pełnieniem służby zawodowej. Obejmuje on dwie części szkolenia, teoretyczną i praktyczną, na podstawie opracowań przygotowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Ten projekt jest bardzo ciekawy i trzeba go promować, aby studenci mogli skorzystać z tego, bo uważam, że osoba, która przejdzie przeszkolenie wojskowe, nabędzie tę umiejętność, będzie przydatna naszej ojczyźnie. Dlatego, panie ministrze, mam takie pytania: Na czym dokładnie polega ten projekt? Jaka kwota zostanie przeznaczona na realizację obecnej edycji i jak wygląda rekrutacja do piątej edycji Legii Akademickiej? Dziękuję. Zapraszam pana ministra. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Zostało też podpisane porozumienie pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Ministerstwem Edukacji i Nauki, wtedy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w zakresie przeprowadzenia szkoleń teoretycznych na terenie szkół wyższych.

Artykuł ten mówi o tym, że minister właściwy dla szkolnictwa wyższego może finansować projekty szczególnie istotne i ważne, w tym wypadku projekt szkolenia w zakresie teoretycznym.

To szkolenie ma charakter teoretyczny, zatem może być również realizowane przez wykładowców czy też pracowników naukowych poszczególnych uczelni. Przypomnę, że w szkołach wyższych cywilnych realizowane są kierunki pn. bezpieczeństwo, bezpieczeństwo narodowe czy bezpieczeństwo zewnętrzne, a więc tutaj ten wymiar teoretyczny jest spełniony.

Na te 15 godzin składa się 13 godzin szkolenia, a 2 godziny przeznaczone są na egzamin.

Gdzie takie szkolenie może się odbywać?

Są to zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne. Jeśli chodzi o szkoły niepubliczne, postanowiony jest warunek, aby liczba studentów na kierunku stacjonarnym była wyższa od 200. Zatem jest to oferta skierowana tak naprawdę do wszystkich szkół wyższych podlegających Ministerstwu Edukacji i Nauki. Chciałbym też bardzo wyraźnie powiedzieć, że ten program z perspektywy Ministerstwa Obrony Narodowej, a projekt z perspektywy Ministerstwa Edukacji i Nauki - jest takim i programem, i projektem, w którym pojawia się to, co moglibyśmy nazwać zjawiskiem synergii. Otóż przede wszystkim Ministerstwo Obrony Narodowej jest zainteresowane tym, aby pozyskiwać młodych ludzi, którzy zdobywają wykształcenie czy to na poziomie inżynierskim, czy też na poziomie studiów II stopnia, więc magisterskich, osoby o bardzo niekiedy wąskich specjalizacjach, wyjątkowo przydatnych chociażby w późniejszej służbie wojskowej.

A więc Ministerstwo Obrony Narodowej ma szansę pozyskania naprawdę świetnych fachowców, którzy mogą być przydatni czy to na poziomie żołnierza szeregowca, czy podoficera, ale również istnieje możliwość kontynuowania szkolenia na poziomie oficerskim - jest to już realizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Jest to też istotne i ważne z punktu widzenia szkół wyższych, dlatego że czymś istotnym i ważnym jest kształtowanie u młodych osób tego, co możemy określić mianem nie tylko patriotyzmu, ale także patriotyzmu rozumianego jako wypełnianie powinności wobec ojczyzny, wobec narodu, wobec państwa. Tak że ta synergia tutaj występuje.

Dotychczas wydatkowano w tych czterech edycjach 3059 tys. zł. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Dziękuję za te dosyć szczegółowe informacje.

Czy są jakieś dodatkowe środki, żeby kampanię informacyjną na temat tych możliwości przeprowadzać?

Czy musi być ten pierwszy etap, żeby przystąpić do modułu szkolenia oficerskiego? Dziękuję. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo!

Ten program cieszy się dużą popularnością, chciałoby się powiedzieć, z tych względów, o których już mówiłem. Ale jest jeszcze jeden wzgląd bardzo istotny.

Szkoła wyższa te środki finansowe otrzymuje.

Przyjmuje się i założenie tego projektu jest takie - programu, a w konsekwencji projektu - że konieczne, niezbędne jest przejście szkolenia teoretycznego na poziomie podstawowym. Później jest ewentualnie poziom podoficerski, a później jest ewentualnie, już we współpracy bezpośrednio z ministrem obrony narodowej, szkolenie na poziomie wyższym.

To jest istotne i ważne, o tym też wcześniej mówiłem.

Posłanki Joanna Jaśkowiak, Iwona Maria Kozłowska i Iwona Hartwich zadadzą pytanie w sprawie zagrożenia zdrowia i życia Polek będących w ciąży. To pytanie jest skierowane do ministra zdrowia, a odpowie na nie sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia pan minister Waldemar Kraska. Bardzo proszę panią posłankę Joannę Jaśkowiak. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Jej serce też biło - wielokrotnie słyszeliśmy ostatnio te słowa. Na każdy kłamliwy argument dotyczący nietykalności życia poczętego będę jak mantrę powtarzać te cztery słowa: jej serce też biło. Jak pan śmie mówić, że to wina lekarza, błąd w sztuce czy jakieś inne bliżej niezidentyfikowane przyczyny? Już małe dzieci uczy się przewidywania konsekwencji ich czynów. Co więcej, ta osoba może ci oddać. a państwo zepchnęliście Polki do podziemia medycznego i wypchnęliście za granicę. Jedynie tam mogą bezpiecznie i bez konsekwencji prawnych usunąć ciąże, szczególnie ciąże zagrożone. Niestety nie wszystkie Polki mogą z takiej drogi skorzystać, chociażby ze względów finansowych, i nie wszystkie Polki chcą z tej drogi skorzystać. To jest niewyobrażalne, że w kraju należącym do Unii Europejskiej kobieta w szpitalu, do którego zwróciła się po pomoc, umiera tylko dlatego, że lekarze czekają, aż serce jej ciężko uszkodzonego płodu przestanie bić. W tym przypadku przestały bić oba serca, a jedno dziecko, dziecko już narodzone, zostało sierotą. Panie ministrze, czy pan, odpowiedzialny za zdrowie i życie również Polek, podejmie działania, by nie dochodziło więcej do takich tragedii? Bardzo proszę, panie ministrze.

Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! W Polsce każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pod szczególną ochroną prawną znajdują się w Polsce kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, którą zapewnia ustawodawstwo krajowe, jak i ratyfikowane przez Polskę umowy międzynarodowe. Zakres i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, zasady i tryb ich finansowania ze środków publicznych oraz zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia równego dostępu do tych świadczeń zostały określone w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Właśnie w tej ustawie zapewniona jest opieka nad kobietą w ciąży, w okresie porodu i połogu, opieka prenatalna nad płodem, opieka nad noworodkiem, wstępna ocena stanu zdrowia i rozwoju niemowlęcia. Zgodnie z tą ustawą kobieta w ciąży ma prawo do świadczeń zdrowotnych poza kolejnością. Jak najwcześniejsze objęcie opieką zdrowotną kobiety w ciąży jest bardzo ważne dla dalszego przebiegu ciąży i zdrowia dziecka. Głównym celem opieki medycznej nad kobietami w ciąży jest zapewnienie prawidłowego przebiegu ciąży oraz jak najwcześniejsza identyfikacja czynników ryzyka, umożliwiająca objęcie pacjentek opieką odpowiadającą ich potrzebom zdrowotnym.

Standard wyznacza sposób organizacji opieki zdrowotnej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej, tj. przebiegu ciąży, porodu, połogu i opieki nad noworodkiem. Szczególne miejsce zajmują w nim przepisy dotyczące organizacji edukacji przedporodowej, wsparcia karmienia piersią, łagodzenia bólu porodowego, a także zasad pracy personelu w przypadkach szczególnie trudnych dla kobiet i ich rodzin, takich jak poronienie, urodzenie martwego lub ciężko chorego dziecka. Zastosowane w standardach rozwiązania kładą szczególny nacisk na współpracę personelu medycznego z rodzicami dla zapewnienia dziecku jak najlepszej opieki. W tym celu standard wskazuje, że wszystkie zabiegi pielęgnacyjne, niezbędne procedury u noworodka są wykonywane w obecności matki, po przekazaniu jej niezbędnych informacji, także po uzyskaniu jej zgody. Standard przewiduje konieczność zapewnienia monitoringu i ewaluacji realizacji jego przepisów. Ponadto zgodnie ze standardem opiekę nad kobietą w ciąży fizjologicznej może sprawować zarówno lekarz ginekolog, jak i położna. Kobieta ma możliwość zapoznania się ze standardem organizacyjnym opieki okołoporodowej, w tym poznania swoich praw i schematu opieki zdrowotnej w okresie ciąży, porodu i połogu oraz opieki nad noworodkiem. Ciężarnej przysługuje co najmniej dziewięć konsultacji z lekarzem lub położną, w trakcie których jest oceniany stan zdrowia i przebieg ciąży.

Opieka jest realizowana w formie wizyt patronażowych. Kobieta ma prawo do co najmniej czterech takich wizyt. Mając na uwadze potrzebę otoczenia szczególną opieką kobiet w ciąży i ich rodzin, w tym przypadku kobiet w ciąży powikłanej i w sytuacji niepowodzeń położniczych oraz dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, zdecydowano o zapewnieniu im kompleksowego wsparcia i przyjęciu stosowanych w tej mierze rozwiązań o wadze rangi ustawowej. W tym celu została uchwalona 4 listopada 2016 r. ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin, tzw. ustawa za życiem, a następnie na jej podstawie został opracowany „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin 'Za życiem'” przyjęty uchwałą Rady Ministrów 20 grudnia 2016 r. Przyjęte rozwiązania wynikają z konieczności zapewnienia przez państwo polskie rodzinom zasłużonego poczucia bezpieczeństwa, szczególnie gdy może wystąpić sytuacja nieodwracalnego upośledzenia lub nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu dziecka. Opieka państwa obejmuje dostęp do odpowiednich świadczeń zdrowotnych, instrumentów polityki na rzecz rodziny realizowanych w ramach programu szeregu działań zmierzających do osiągnięcia przedmiotowego celu określonego w ramach sześciu priorytetów. Dzieciom, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, oraz dzieciom mającym orzeczenie o niepełnosprawności, w odniesieniu do dzieci do 16. roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności, łącznie ze wszystkimi wskazaniami, przysługuje ustawowo prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu finansowanego ze środków publicznych, korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, korzystania ze świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania (Dzwonek), korzystanie z rehabilitacji bez limitu, wyszczególnionych w odrębnych przepisach. W celu poprawy opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu oraz nad nowo narodzonym dzieckiem został wprowadzony zakres świadczeń, koordynowana opieka nad kobietą w ciąży. Panie Marszałku! Szanowni Panie i Panowie Posłowie! Bardzo proszę. Pani poseł Iwona Maria Kozłowska. Panie marszałku, dziękuję bardzo. Panie ministrze, wysokie standardy, a kobiety umierają. Dziękuję, że pan wspomniał o programie „Za życiem”, bo mijają właśnie 4 lata od rozpoczęcia tego programu. Celem tego programu była pomoc kobietom w powikłanej ciąży oraz rodzinom z dziećmi, u których zdiagnozowano ciężkie nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę, która zagraża ich życiu.

Ile rodzin otrzymało potrzebną pomoc w ramach programu? Ile kobiet skorzystało z opieki psychologicznej w ramach programu „Za życiem” W jakiej formie pomoc była realizowana? W ilu mieszkaniach chronionych zamieszkały rodziny z chorymi dziećmi? Ile z deklarowanych 30 (Dzwonek) powstało ośrodków neonatologiczno-pediatrycznych? Czy we wszystkich województwach kobiety miały możliwość skorzystania z opieki paliatywnej i hospicyjnej? Kiedy do Sejmu trafi obiecany po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 22 października projekt pomocy dla kobiet i dzieci ze zdiagnozowaną poważną wadą, w tym letalną? Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Zapraszam, panie ministrze. Uprzejmie pana informuję, że na część tych pytań może pan również odpowiedzieć pisemnie, bo na pewno nie zdążymy ze wszystkim. Szanowni Państwo! Wszystkie te pytania są skierowane akurat nie do Ministerstwa Zdrowia, tylko do ministerstwa rodziny, więc myślę, że odpowiemy na piśmie razem z ministerstwem rodziny. Aż o taki skrót pana nie prosiłem, ale jest, jak jest. Proszę państwa. Tak, właśnie pan minister to powiedział. Przechodzimy do następnego pytania. Pan poseł Marek Polak oraz pani poseł Anna Kwiecień z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zadadzą pytanie w sprawie przygotowania służby zdrowia do czwartej fali pandemii, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania lecznictwa szpitalnego, w tym szpitali tymczasowych, oraz poziomu wyszczepienia Polaków i przewidywanych działań rządu w związku z rozwojem pandemii koronawirusa.

Dobra, zaczynamy. Pan poseł Marek Polak. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Sięgające kilkunastu tysięcy dzienne liczby zakażeń w ostatnich tygodniach wyraźnie wskazują, że jesteśmy w zaawansowanym punkcie czwartej fali koronawirusa. Wszyscy wiemy, że szczepienia są kluczowym narzędziem w walce z utrzymującą się pandemią. Z uwagi na liczne punkty szczepień i trwającą od dłuższego czasu kampanię informacyjno-promocyjną Polacy mają szerokie możliwości uzbrojenia się w to dobrodziejstwo, jakim jest szczepionka. Chciałbym zapytać, jak kształtuje się poziom wszczepienia wśród Polaków, czy są to tendencje rosnące oraz czy w obliczu dalszego wzrostu liczby zachorowań rozważane jest wprowadzenie lockdownu. Dziękuję bardzo. Pani poseł Anna Kwiecień. Dziękuję bardzo. Panie Ministrze! Chciałabym dopytać o stan przygotowań szpitali do czwartej fali epidemii, ze szczególnym uwzględnieniem szpitali tymczasowych. Czy ich uruchomienie obarczone jest jakimiś turbulencjami? Ile mamy przygotowanych miejsc respiratorowych? I czy na bazie doświadczeń z trzeciej fali i drugiej fali wprowadzamy jakieś korekty w walce z epidemią? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszam pana ministra.

Panie Marszałku! Rzeczywiście w tej chwili wkraczamy, właściwie wkroczyliśmy już w czwartą falę. Codziennie mamy bardzo dużo nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Dzisiaj także padł niestety kolejny rekord.

Dlatego tak bardzo ważną rzeczą jest, abyśmy promowali i zachęcali Polaków do szczepień.

Oczywiście jest to niewystarczające, aby osiągnąć odporność populacyjną, dlatego w tej chwili, jak mówią lekarze, którzy na co dzień zajmują się pacjentami chorymi na COVID-19, do polskich szpitali trafiają osoby niezaszczepione i to właśnie te osoby wymagają tej bardzo wysokospecjalistycznej procedury, jaką jest podłączenie do respiratora czy też aparatów ECMO.

To jest związane nie tylko ze szczepieniem na COVID-19, ale także z innymi szczepieniami.

W tej chwili mamy już sprowadzonych 80 mln.

Mamy w tej chwili przygotowanych także prawie 2 tys. łóżek OIOM-owych, czyli łóżek, które są wyposażone w respiratory. Na dzień dzisiejszy mamy 1300 zajętych respiratorów. Niestety coraz częściej trafiają tam osoby bardzo młode. Jeden szpital w Lubelskiem zgłosił, że średni wiek pacjenta, który jest u nich na respiratorze, wynosi 30 lat.

Ta nowa mutacja, która w tej chwili jest w Polsce, powoduje to, że bardzo często niestety chorują osoby młode. Dużo osób trafia także właśnie na oddziały intensywnej terapii, ponieważ zgłaszają się za późno.

Dzisiaj planujemy uruchomienie dodatkowego szpitala tymczasowego we Wrocławiu, a w przyszłym tygodniu, jeżeli sytuacja epidemiologiczna będzie tego wymagała, a wydaje się, że będzie taka konieczność, uruchomimy szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym.

Pytanie dodatkowe? Panie Ministrze! Chciałabym zadać dodatkowe pytanie o to, jak przebiega współpraca samorządów z Ministerstwem Zdrowia w zakresie walki z pandemią koronawirusa. Czy prawdą jest, że blokowane są przyjęcia pacjentów chorych na COVID-19 do niektórych szpitali samorządowych? Jakie macie państwo narzędzia do tego, żeby walczyć z takimi sytuacjami? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Rzeczywiście, pandemia pokazała, że organy prowadzące szczególnie szpitale nie zawsze chcą współpracować. To znaczy, państwo musi zapewnić wszystkim równy dostęp do opieki zdrowotnej. Wojewodowie, przygotowując plany zabezpieczenia, rozmawiają najczęściej z dyrektorami szpitali, z ich organami prowadzącymi. Myślę że takim przykładem braku współpracy - ja zresztą o tym już wielokrotnie mówiłem - jest miasto stołeczne Warszawa, gdzie niestety ta współpraca nie układa się tak, jak byśmy chcieli.

Akurat, jak mówię, miasto stołeczne nie chce tutaj współpracować tak, jak byśmy chcieli, szczególnie na płaszczyźnie między wojewodą a panem prezydentem.

Tych łóżek tutaj naprawdę zawsze potrzeba.

Zada je pan poseł Grzegorz Adam Woźniak z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Pytanie jest w sprawie stanu zaawansowania prac i terminu ukończenia modernizacji wałów wiślanych w gminie Maciejowice i jest skierowane do ministra infrastruktury. Odpowie podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury pan Grzegorz Witkowski. Bardzo proszę, panie pośle. Panie Marszałku! Panie Ministrze!

Rozmówcy wracają wspomnieniami do ostatnich zagrożeń, jakie miały miejsce w latach 2010 i 2014. W roku 2015 oddano do użytku zmodernizowany wał przeciwpowodziowy na odcinku od Antoniówki Świerżowskiej do Krasek.

Udało się doprowadzić do wznowienia prac na wałach.

Część środków pochodzi z Wód Polskich oraz urzędu marszałkowskiego. Wystąpiłem wtedy z pismem do ministra, do Wód Polskich o rozważenie możliwości przeznaczenia pozostałej zaoszczędzonej kwoty na dalszą modernizację wałów w kierunku Wilgi na terenie gminy Maciejowice.

Dziękuję bardzo.

Bardzo proszę, panie ministrze. Pan minister Grzegorz Witkowski. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo!

Projekt obejmuje wykonanie m.in. robót ziemnych związanych z przebudową korpusu wału i ławy przywałowej, uszczelnienie korpusu wału matą bentonitową, przebudowę przepustu wałowego, wykonanie umocnienia drogi eksploatacyjnej.

Tam rzeczywiście w celu realizacji zadania uzyskano niezbędne decyzje administracyjne dla tego trzeciego etapu, które w przypadku niewykonania zadania stracą ważność. I bardzo dziękuję parlamentarzystom z Garwolina, z Mazowsza, z tamtej części za silny nacisk, lobbing w Ministerstwie Finansów i w Ministerstwie Infrastruktury. Jeśli chodzi o gminę Wilga, to tam również jest o wiele większy zakres inwestycyjny, ale też większe kwoty.

Nie da się zacząć inwestycji w gminie Wilga bez zakończenia inwestycji w gminie Maciejowice. To może pan poseł, panie marszałku, dopowie. Bardzo proszę, panie pośle.

Będziemy wiedzieć, co mieszkańcom przekazać. Bardzo proszę. Tak, rzeka Wilga.

Tam udało się nam wszcząć procedurę przetargową na zabezpieczenie Wisły przed erozją na odcinku 1 km. Będzie tam wykonany narzut kamienny razem z przykryciem brzegu stalową siatką.

Podwyższenie nasypu ziemnego, podwyższenie wału poprzez wykonanie bulwaru.

Generalnie budowa muru oporowego, podwyższenie, wykonanie przejazdów wałowych, nasadzenie wiklin, umocnień brzegowych, budowa drogi eksploatacyjnej.

Mamy takie rozdwojenie jaźni: z jednej strony jest bezpieczeństwo Polski i Polaków, bezpieczeństwo mieszkańców rzek, a z drugiej strony jest troska, czasem nadmierna, o środowisko naturalne.

Proszę państwa, zakończyliśmy punkt dotyczący zadawania pytań opowieścią o powstawaniu wałów i trudnej pracy z tym związanej. Przechodzimy do następnego punktu. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 17. porządku dziennego: Informacja bieżąca. Przypominam, że na obecnym posiedzeniu Sejmu zostanie rozpatrzona informacja w sprawie ubożenia społeczeństwa na skutek skokowego wzrostu cen i braku równoważącego go wzrostu dochodów, w szczególności osób zatrudnionych w sferze budżetowej, o której przedstawienie wnosi Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni. Przypominam również, że przedstawienie uzasadnienia wniosku przez posłów przedstawicieli wnioskodawców, a będzie ich dwoje, nie może trwać dłużej niż 5 minut, a udzielenie odpowiedzi przez przedstawicieli Rady Ministrów, a też będzie ich dwoje - dłużej niż 10 minut. Wystąpienia posłów w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 2 minuty. Na zakończenie dyskusji głos zabierają kolejno przedstawiciel wnioskodawców oraz przedstawiciel Rady Ministrów. Wystąpienie przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a wystąpienie przedstawiciela Rady Ministrów - dłużej niż 10 minut. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie wystąpienia przedstawiciela Rady Ministrów. Czas przeznaczony na rozpatrzenie punktu: Informacja bieżąca nie może być dłuższy niż 90 minut. Zanim oddam głos i poproszę o zabranie głosu pana posła Sławomira Nitrasa, zwrócę się z pytaniem do Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska.

W ten sposób zadacie pytania, a jeżeli będzie pytanie wyjątkowo skomplikowane, to dołożymy kilka sekund, dobrze?

Bardzo proszę pana posła Sławomira Nitrasa o zadanie pytania w pierwszej części, a potem poproszę panią poseł Izabelę Leszczynę. Panie Marszałku! Z tego, co zdążyłem się zorientować, wynika, że odpowiadać będzie nam pan minister Patkowski z Ministerstwa Finansów. Rozmawiamy o sprawie niezmiernie poważnej, w której moim zdaniem powinna nastąpić pewna zgoda w tej Izbie, o wynagrodzeniach w sferze budżetowej, o tym, ile zarabiają polscy urzędnicy, ile zarabiają polscy nauczyciele, o tym, ile zarabiają pracownicy służby zdrowia. Wymieniam te największe grupy. Panie ministrze, chciałbym pana zapytać, jaką dostał pan ostatnio podwyżkę. Ile zarabia pan więcej? Bo według moich informacji w ciągu ostatnich miesięcy dostał pan ponad 4 tys. netto podwyżki. Pana podwyżka, tylko podwyżka, jest wyższa niż wynagrodzenie, które otrzymują urzędnicy, którzy dla Polski pracują, nauczyciele, którzy uczą nasze dzieci. Zadajemy to pytanie z prostego powodu. Słyszymy praktycznie każdego dnia pana premiera Morawieckiego i innych urzędników rządu, którzy mówią: szanowni państwo, wasze pensje rosną szybciej niż inflacja. Co z tego, zdaniem pana Morawieckiego, że inflacja rośnie już w tempie prawie 8-procentowym w skali rok do roku - tak będzie - skoro pensje rosną szybciej? Przeanalizujmy to, szanowni państwo. Myślę, że jest zgoda również polityków PiS-u na to, żeby to spokojnie przeanalizować.

Pomyśleli sobie: pensja minimalna wzrasta, jest szansa, że dostaniemy podwyżki, bo nasze wynagrodzenia są poniżej płacy minimalnej. Przecież to nie zależy od was, a jeżeli zależy, to raczej podnosicie ludziom podatki. Od was, od rządzących w Polsce, poza inflacją, która zależy od was, realnie zależą wynagrodzenia w administracji, w sferze publicznej, w szkołach, w szpitalach. Ale dramatyczna inflacja w tej chwili zżera te zarobki. Co z tego, że podnosicie płacę minimalną ludziom pracującym w szkołach, skoro inflacja rośnie dwukrotnie szybciej?

Największą grupę stanowią komendy powiatowe Policji i komendy powiatowe straży pożarnej.

Z wszystkimi się filmujecie. Sądy i prokuratury przez ostatnie 6 lat zostały tak zreformowane, że kamień na kamieniu nie został. Wiecie, że tu już nie chodzi w tej chwili o minimum egzystencji. Tu już nie chodzi w tym wszystkim o to, czy ludzie mają poczucie, że są w stanie się utrzymać. Tu chodzi o elementarną godność, o to, że ktoś, kto pracuje dla państwa polskiego, kto uczy nasze dzieci, ktoś, kto pracuje w sądzie, ktoś, kto pracuje w prokuraturze, zarabia płacę minimalną. Pan minister Niedzielski miał odwagę powiedzieć ratownikom medycznym, żeby się nie martwili. Ich płace muszą wzrosnąć w przyszłym roku, bo rośnie płaca minimalna i nie mogą pozostać poniżej płacy minimalnej. O tym jest dyskusja. Pytanie jest o to, czy jesteście gotowi usiąść i na poważnie się zastanowić, jak ten problem rozwiązać. Jak tę wielką dysproporcję pomiędzy gospodarką, która się rozwija, a administracją państwową, którą doprowadziliście na skraj ruiny, jeśli chodzi o kadry. Czy jesteście gotowi do poważnej debaty? Jesteśmy. Tu chodzi dzisiaj o to, żeby ratować egzystencję polskiej administracji, polskiej szkoły, żeby ktokolwiek chciał uczyć nasze dzieci, żeby państwowa służba zdrowia, publiczna służba zdrowia była realna, bo dzisiaj staje się fikcją. Ciekawi jesteśmy, czy jesteście gotowi do tej debaty. My jesteśmy do niej gotowi dla tych wszystkich pracowników i ludzi, którzy ze sferą publiczną wiążą swoje nadzieje. Dziękuję, panie pośle.

Człowiek rzuci perłę i po prostu lecą diamenciki z tej sali równiutko. Proszę o udzielenie odpowiedzi sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej panią minister Annę Schmidt. Wszystko się zmienia, panie pośle. 10 sekund trwa 40, jeden minister zmienia się na drugiego ministra. Dobrze, ale nie ma jeszcze pani minister, więc już może mnie nie. Dobrze, ale mogę w tym czasie coś mówić czy nie za bardzo? Wysoka Izbo! Polska, podobnie jak wiele innych krajów na świecie, boryka się z problemem wzrostu cen. Jak poinformowała Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, globalny indeks cen żywności we wrześniu 2021 r. ponownie wzrósł, tym razem do poziomu najwyższego od 10 lat. To, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że nasz kraj boryka się z problemem braku rąk do pracy.

Wśród pięciu najbardziej pożądanych specjalizacji znaleźli się pracownicy obszaru logistyki, operatorzy produkcji i maszyn, pracownicy działu IT, pracownicy administracji i obsługi biura oraz pracownicy bezpośredniej obsługi klienta. Był to jeden z powodów, dla którego pracodawcy mimo pandemii koronawirusa ostrożnie podejmowali decyzje kadrowe i przy wykorzystaniu wsparcia, jakie otrzymali z tarczy antykryzysowej, zachowali miejsca pracy. Dzięki temu nie doszło do drastycznego wzrostu bezrobocia, choć w pierwszych miesiącach po wybuchu pandemii pojawiały się takie zapowiedzi. W bieżącym roku sytuacja na rynku pracy z miesiąca na miesiąc się poprawiała. W czerwcu br. po raz pierwszy od ponad roku poziom rejestrowanego bezrobocia spadł poniżej 1 mln osób. Według wstępnych danych w końcu października 2021 r. w urzędach pracy zostało zarejestrowanych 912 tys. osób bezrobotnych, czyli w porównaniu ze stanem z końca września 2021 r. liczba ta zmniejszyła się o ponad 22 tys. Tempo spadku było pięciokrotnie silniejsze niż w październiku 2020 r. W odniesieniu do października ub.r. poziom bezrobocia zmniejszył się o ponad 106 tys. osób, czyli o ponad 10%.

Polska od kilku miesięcy jest krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej.

Tym samym Polska zajęła ex aequo z Niemcami czwarte miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w Unii Europejskiej. Pokazuje to, że szybko i dobrze zaplanowane działania rządu zawarte w tarczy antykryzysowej pomogły przezwyciężyć trudności finansowe i umożliwiły kontynuację działalności gospodarczej wielu firmom, a pracownikom pozwoliły zachować miejsca pracy.

Dzięki tym zmianom będzie można uzyskać nie tylko wyższe świadczenie pieniężne, ale objąć wsparciem także większą liczbę osób i rodzin. Dotyczy to w szczególności zasiłków stałego, okresowego i celowego. Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wynoszą 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej, to jest wzrost o 11%, i 600 zł dla osoby w rodzinie, wzrost o 14%. Należy podkreślić, że polityka rodzinna jest jednym z najważniejszych obszarów działania polskiego rządu, dlatego ustawicznie podejmowane są nowe inicjatywy zmierzające do zwiększenia wsparcia na rzecz rodzin. Instrumenty polityki rodzinnej są. Panie marszałku, pan poseł mi przeszkadza. Panie pośle, chce pan posłuchać, co mam do powiedzenia? Ale posłuchajcie, posłuchajcie.

Ale posłuchajcie, możemy zakończyć ten etap? Bardzo proszę. Efektem działań rządu w zakresie polityki rodzinnej jest wprowadzenie znaczącej pomocy finansowej rodzinom. Zdaje się, że mówimy o obłożeniu społeczeństwa, więc polityka prorodzinna w mojej ocenie, panie pośle, nie wiem czy w pańskiej, wpisuje się w zakres pytania. Jednym z flagowych programów rządowych jest wprowadzony 1 kwietnia 2016 r. rządowy program 500+, który stanowi fundament wsparcia polskich rodzin. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze ma charakter powszechny i przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia niezależnie od dochodu rodziny.

Odmienił życie wielu rodzin. Stały się one zamożniejsze, pojawiły się lepsze perspektywy ich rozwoju. Wsparcie to przyczynia się do zapewnienia dzieciom solidnego wykształcenia, odpowiedniego odżywiania i leczenia, a także pozwala rodzinom na zwiększenie wydatków, m.in. na edukację i rekreację.

Kolejny program, o którym chcę wspomnieć, to wprowadzony w 2018 r. rządowy program „Dobry start”, który ma na celu wsparcie rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. Jest on kolejnym komponentem prowadzonej przez rząd kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej kierowanej do wszystkich rodzin wychowujących dzieci. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych niezależnie od kapitału kulturowego, społecznego i materialnego rodziny.

Jednocześnie rząd, zmierzając do jeszcze szerszego wsparcia polskich rodzin, przedstawił najnowszą deklarację programową Polski Ład.

Przewiduje także dużo większe nakłady na rozwój sieci instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi. Jednym z rozwiązań przewidzianych w Polskim Ładzie jest wprowadzenie nowego finansowego instrumentu wsparcia, jakim będzie rodzinny kapitał opiekuńczy. Dodatkowo w ramach Polskiego Ładu planowane jest wprowadzenie dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w przypadku dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie świadczeniem wypłacanym rodzicom na pokrycie kosztów opieki nad drugim dzieckiem pomiędzy 12 a 36 miesiącem życia.

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ma wynosić 400 zł miesięcznie i będzie przekazywane bezpośrednio prowadzącemu instytucję opieki. Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym nowelizująca ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 zakłada, że przepisy dotyczące finansowania opłaty za pobyt dziecka wejdą w życie od 1 kwietnia 2022 r. Karta tworzy system zniżek ustawowych i handlowych oferowanych przez podmioty z różnych branż. Obecnie zniżki oferuje 9 tys. partnerów.

Proszę państwa, przechodzimy do zadawania pytań. Pan poseł Wiesław Janczyk, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Zapraszam, panie pośle.

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Z uwagą wysłuchałem wystąpienia pana posła Nitrasa, które było wyjątkowo spokojne.

Proszę państwa, inflacja nie jest domeną tylko tej szerokości geograficznej.

My pytamy o zarobki osób pracujących w sferze budżetowej, tych, które są zależne od państwa, a państwo opowiadają o 500+. My pytamy o inflację, państwo opowiadają o 500+. Całkowicie nie na temat. Nauczyciel stażysta, który ma przyjść do zawodu, który zwykle nie ma jeszcze dzieci, więc nie pobiera 500+, dostaje minimalną pensję w wysokości 2949 zł. To jest pauperyzacja zawodu nauczyciela. Oznacza to, że do tego zawodu trafiają nie najlepsi, tylko ci, którzy nie mają innego wyjścia lub są niesamowitymi pasjonatami. W wyniku tego w bardzo wielu miejscach w Polsce w ogóle nie ma nauczycieli.

64% Polaków powiedziało bardzo jasno: w ciągu ostatniego roku nie dostaliśmy żadnych podwyżek. Dziękuję. Pan poseł Jan Szopiński, klub parlamentarny Lewica.

Faktyczny skokowy wzrost cen i kosztów życia już teraz znacznie przekracza kwotę symbolicznych podwyżek.

W związku z tym, szanowna pani minister, dwa pytania. Kiedy rząd podejmie działania antyinflacyjne, które przywrócą siłę nabywczą pensji pracowników budżetówki?

Pan poseł Jacek Protasiewicz, Klub Parlamentarny Koalicja Polska. Panie Marszałku!

Cieszcie się więc, obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Jak rosną ceny produktów? Masło kosztuje już prawie 10 zł. Olej kujawski - 100% podwyżki.

Dziękuję. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Uprzejmie dziękuję. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Drożyzna to jest to jedno słowo, które opisuje dokonania rządu PiS w ostatnich latach. Pędząca inflacja, rosnące ceny w sklepach, rosnące ceny usług. To efekt rządów pana prezydenta Dudy, premiera Morawieckiego i prezesa Glapińskiego. Złe decyzje, podwyżki podatków, drukowanie pieniędzy, mętna polityka budżetowa i utrata zaufania rynku. Polska 2050 proponuje konkretny program antyinflacyjny: piątka Hołowni. Proponujemy obniżkę VAT do 20% i do 7%, zawieszenie poboru opłaty emisyjnej, przeznaczenie przychodów z handlu emisjami na dopłatę do rachunku za energię, przeznaczenie 6 mld zł z gazowego arbitrażu na redukcję cen za gaz i zawieszenie Polskiego Ładu na co najmniej rok, bo to jest kolejny impuls inflacyjny. Co dla rządu PiS jest ważniejsze: troska o ludzi czy dalsze bezmyślne trwanie u władzy? Czy prawdą jest, że za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, począwszy od 2017 r., poziom cen oscyluje w granicach 2%, a więc jest zgodny ze średniookresowym celem inflacyjnym?

Czy prawdą jest, że wzrost cen w drugiej połowie 2021 r. jest spowodowany czynnikami niezależnymi od rządu i polityki gospodarczej, często pozostającymi poza obrębem naszej gospodarki? Chodzi mi tutaj o czynniki podażowe, o wzrost cen paliw wskutek wzrostu ceny ropy naftowej, a także ograniczania jej podaży.

Podobnie ceny energii elektrycznej, które są - jak państwo powinniście wiedzieć - wymuszane przez politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Pourywane sieci dostaw.

Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo! W zeszłym roku w Polsce zmarło 485 tys. ludzi. Chcę się upomnieć o tych, dla których premier Morawiecki nie ma czasu od września, od momentu, kiedy powstało białe miasteczko.

Kształcenie skończyło 5 tys., a więc o połowę mniej. Cztery pielęgniarki odeszły, a jedna trafiła do publicznej służby zdrowia.

To pokazuje, w jakiej sytuacji jest dzisiaj Polska. Szpitale nie będą funkcjonowały bez pielęgniarek i położnych, a ludzie będą umierali, jeśli nie przedstawicie projektu realnego podwyższenia płac dla pielęgniarek i położnych. Pan poseł Rafał Adamczyk, klub parlamentarny Lewica. Panie Marszałku! Pani Minister! Mówimy o ułożeniu społeczeństwa ze względu na wzrost cen. Nie mówimy głośno o ubóstwie energetycznym Polek i Polaków. Węgiel w przeciągu 1 roku zdrożał o ponad 80%.

Gdzie są wypowiadane w 2019 r. zapewnienia, że cena prądu się nie zmieni?

Pan poseł Dariusz Klimczak, Klub Parlamentarny Koalicja Polska. Wysoka Izbo! Według danych GUS poziom tzw. ubóstwa skrajnego za rok 2020 wynosił w Polsce 5,2%, co oznacza, że poniżej minimum egzystencjalnego w Polce żyło prawie 2 mln osób. To oznacza wzrost o 1% w stosunku do roku 2019, co - przekładając to na liczby bezwzględne - wynosi 377 tys. osób więcej żyjących w skrajnym ubóstwie. Natomiast w tym roku mamy dodatkowy problem, jest nim inflacja, drastyczny wzrost cen, szczególnie na artykuły pierwszej potrzeby. Dotyka to osób najmniej zarabiających. I pytanie do rządu, szczególnie do pani minister, która tu przedstawiała szeroki wachlarz działań, jakie działania osłonowe w związku z tym planuje rząd, planuje ministerstwo, żeby nie doprowadzić do tego, aby ta (Dzwonek) ogromna liczba osób jeszcze się zwiększyła. Dziękuję. Panie i Panowie Posłowie! W skrajnej biedzie żyje w Polsce już 2 mln Polek i Polaków. Powtórzę: 2 mln obywateli żyje w skrajnej biedzie. Najpierw pandemia, teraz drożyzna. Rosnące koszty życia będą w tę grupę wpychać kolejne osoby - pracujące, mniej zarabiające, ale także emerytów, także dzieci. Mówicie, że inflacja jest w całej Europie. Nie taka. Polska ma jedną z najwyższych inflacji i doprowadziliście do tego swoją polityką gospodarczą przez ostatnie lata. To m.in. osłabianie złotego, dodrukowanie na masową skalę pustego pieniądza, ale także wprowadzanie do systemu podatkowego licznych nowych opłat i podatków.

Bo w ustawie budżetowej na przyszły rok, pani minister, nie ma w ogóle odpowiedzi na podstawowe wyzwanie, jakim jest narastająca drożyzna i wzrost ubóstwa w gronie Polek i Polaków. Proszę o zabranie głosu pana posła Tadeusza Cymańskiego. Jakie znaczenie dla osłabiania, dla łagodzenia skutków inflacji, dla szerokich grup społecznych ma Polski Ład? Krótko. 2020 r., rok pandemiczny, spowodował nieoczekiwane skutki. Jeżeli chodzi o grupę najlepiej uposażonych Polaków, odnotowano realny wzrost o ponad 7%. Tymczasem jednocześnie grupy najsłabsze straciły ponad 6%. I reakcją każdego rządu nie tylko od inflacji, ale w ogóle reakcją muszą być działania, których celem jest poprawa sytuacji ogromnych grup społecznych. Rozwarstwienie jest dalej faktem pomimo ogromnych, bardzo skutecznych działań obecnego rządu. Proszę to rozwinąć, bo mi skromny czas nie pozwala. Chciałbym i mógłbym, ale nie mogę w tej chwili, a pan może. Bardzo dziękuję. Pytanie zada pan poseł Arkadiusz Myrcha. Pani Minister! Pracownicy sfery budżetowej, w tym pracownicy prokuratur i sądów, pytają: Skoro jest tak dobrze, to dlaczego musimy walczyć o godność? Skoro jest tak dobrze, to dlaczego ulicami Warszawy przeszedł największy od 30 lat protest pracowników prokuratur i sądów? Skoro jest tak dobrze, to dlaczego mamy czerwone miasteczko i ludzi, którzy od wielu dni siedzą w namiotach na mrozie, kosztem swojej rodziny, kosztem swojej pracy? Skoro jest tak dobrze, to gdzie są te pieniądze? Ministerstwo Sprawiedliwości w 6 lat swój budżet zwiększyło trzykrotnie: z ponad 200 mln do ponad 600 mln.

Proszę pana posła Tadeusza Tomaszewskiego z klubu Lewica. Wysoki Sejmie! Drożyzna wynikająca z inflacji, brak konkretnych działań rządu zżerają każdego dnia w szczególności płace, świadczenia społeczne, renty i emerytury. Dziś bardzo wielu ludzi, zwłaszcza osób samotnych, będących w trudnej sytuacji z powodu złego stanu zdrowia zastanawia się, czy utrzyma swoje mieszkanie, czy utrzymana swój dom, dorobek swojego życia. A rząd w tej sprawie nic nie czyni. W związku z powyższym chciałbym zapytać: Jakie konkretne działania rządu będą w najbliższym czasie przedstawiane parlamentowi, jeśli chodzi o sprawę dotyczącą energii elektrycznej? Czy tylko wybrane gospodarstwa, czy pomoc dla wszystkich gospodarstw? Czy będzie obniżka akcyzy na paliwa?

Bardzo proszę o konkretne odpowiedzi. Bardzo dziękuję. Pytanie zada pan poseł Stefan Krajewski. Szanowny Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo!

Bardzo proszę o pomoc dla ludzi, których nie stać na założenie gazu i nadal palą w piecach węglem. W ogóle nie ma węgla na składach. Babcia ma emerytury 2100 zł, a tona węgla kosztuje już w tej chwili 1800 zł. A gdzie reszta: opłaty, życie, leki? Kopalnie wydają tylko po 5 t i za chwilę będzie problem z dostępnością. Rozumiem wszystko, ale tak żyć się nie da. Jak żyć? Będziemy ganiać z płachtą po chrust do lasu? Oczywiście z przekąsem pisze pani. Tak to wygląda. Bardzo dziękuję panu posłowi. Proszę teraz o zabranie głosu pana posła Michała Gramatykę. W takim razie pan poseł Robert Gontarz. Wysoka Izbo! Ale podstawową kwestią jest to, żebyśmy zrozumieli, z czego wynika inflacja. Inflacja, przynajmniej bazowa, wynika z dwóch podstawowych kwestii: tempa cyrkulacji pieniądza i ilości pieniądza w gospodarce. Rok 2020 był szczególnie trudnym rokiem w naszej gospodarce i dzięki zdecydowanej i natychmiastowej działalności rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego do polskiej gospodarki na ratowanie milionów miejsc pracy do gospodarki zostało wtłoczonych nawet ponad 200 mld zł. W momencie odbicia gospodarczego ten pieniądz zaczął krążyć i to niestety spowodowało wzrost inflacji. Do tego dochodzą ceny surowców energetycznych, a także przerwanie łańcuchów dostaw. Pojawia się pytanie, być może nawet pytanie zasadnicze.

Przecież taki kryzys, który był porównywalny do kryzysu z II wojny światowej, mógłby doprowadzić do utraty miejsc pracy (Dzwonek) nie przez dodatkowy 1 mln, ale nawet przez 2 mln osób. Szanowni państwo, gdybyśmy podjęli tak nieodpowiedzialną decyzję jak wy teraz, moglibyśmy być pod kątem rynku pracy w naprawdę tragicznej sytuacji. Proszę o zabranie głosu panią poseł Barbarę Nowacką. Pani Minister! Nie wiem, co pani właśnie zrobiła. My pytamy o strefę budżetową, o to, dlaczego pracownicy, którzy pracują dla instytucji publicznych, dla dobra Rzeczypospolitej na państwowych posadach, są coraz biedniejsi. Doprowadzacie do pauperyzacji ludzi, którzy ratują instytucje, które wy rozwalacie, którzy działają jako kuratorzy sądowi, nauczyciele, pielęgniarki, często pracownicy biurowi. Bardzo często żyją bardzo biednie, bardzo skromnie, ratując państwo i patrząc na to, w jaki sposób wy niegospodarnie działacie. Jeżeli urzędnicy państwowi zarabiają płacę minimalną albo trochę powyżej, pracownicy budżetówki żyją bardzo często wspólnie ze swoimi rodzinami na granicy ubóstwa, a wy im opowiadacie, że jest świetnie, to to jest po prostu niegodne. Musicie pamiętać, że na was jako rządzących spoczywa specjalna odpowiedzialność dbania o państwo.

To jest bardzo złe dla państwa i przynosi tragiczne konsekwencje. Bardzo dziękuję. Głos zabierze pan poseł Marcin Porzucek. Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! To znamienne, że wniosek Koalicji Obywatelskiej nie był prezentowany przez osoby, które zajmują się finansami publicznymi na co dzień, przez panią minister Leszczynę, przez panią przewodniczącą Skowrońską. Wybraliście państwo do tego pana posła Nitrasa. Dlaczego? Bo państwo chcecie robić polityczną hucpę. Państwo nie macie żadnego pomysłu, jak rozwiązać problem inflacji. Sytuacja jest opanowywana przez nasz rząd. Faktycznie. Inflacja jest od lat najwyższa w Polsce, ale spójrzcie, co się dzieje w Niemczech, gdzie zarządza pani Kanclerz Merkel. Tam jest najwyższa od prawie 30 lat. W 2004 r. Polska weszła do Unii Europejskiej razem z dziewięcioma innymi krajami, głównie z naszego regionu. W żadnym z tych krajów (Dzwonek) ceny paliw nie są niższe niż u nas. Dlaczego? Być może po prostu rząd Mateusza Morawieckiego dobrze zarządza Polską?

Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana marszałka Cezarego Grabarczyka. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Inflacja i drożyzna to rezultat, jak mawiał Stefan Kisielewski - Kisiel, to skutek rządów Prawa i Sprawiedliwości. Drożyzna oszalała, ale chciałem zwrócić uwagę także na sektor rolniczy. Oszalały ceny nawozów sztucznych. Kilka tytułów: „Ceny na rynku nawozów oszalały, podbiją koszt żywności”, „Rolnicy w szoku, ceny nawozów zwariowały”, „Ceny nawozów od stycznia bardzo wzrosły” Jaki będzie tego rezultat? Zdrożeje żywność. Tymczasem mamy grupy zawodowe, które otrzymują minimalne wynagrodzenie.

I jeszcze jedno pytanie: Czy to prawda, że chcecie pozbawić premii motywacyjnej znaczną część pracowników cywilnych Policji? Proszę o zabranie głosu pana posła Adama Gawędę. Wysoka Izbo! Wzrost inflacji nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie rzeczywiście budzi zaniepokojenie wielu ekspertów.

Wzrost cen ma swoją genezę w niespotykanej dotąd skali oddziaływania na gospodarkę, bo pandemia, z którą się zderzyliśmy, instrumenty, które zastosowaliśmy, rzeczywiście uchroniły Polskę przed bardzo poważnymi konsekwencjami. Również nie ukrywam, że bardzo duże znaczenie ma polityka klimatyczna Unii Europejskiej prowadząca do drożyzny cen energii i nośników energii. Kilka faktów. Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej poprawiła deficyt o 17 punktów procentowych. To najlepszy wynik wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Panie marszałku, i kilka zestawień, dosłownie 10 sekund.

Dla średnio zarabiających - 618 l, obecnie - 917 l. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana posła Janusza Cichonia. Wysoka Izbo! Jeszcze dzisiaj głosować będziemy nad podwyżkami dla osób zajmujących się cyberbezpieczeństwem.

to jest ponad 40 tys., bo trzeba walczyć i zapewnić bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo. Na pewno tak. Ale w tym kontekście upominam się o administrację skarbową. Bez nich tak naprawdę nie będzie dochodów budżetu państwa. Od nich one zależą. Brakuje wykwalifikowanych kadr. Najlepsi odchodzą ze względu na wynagrodzenia, przechodzą na ciemną stronę mocy. To jest zagrożenie (Dzwonek) dla bezpieczeństwa finansów państwa.

Głos zabierze pani poseł Katarzyna Czochara. Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam pytanie do pani minister: Czy ministerstwo posiada dane, aktualne dane dotyczące sytuacji rodzin wielodzietnych po wprowadzonych programach, chociażby „Mama 4+”, 500+, 500+ dla niesamodzielnych, skokowy wzrost rent i emerytur, 13., 14. emerytura.

Dzisiaj ponownie słyszałam tutaj wiele słów krytyki. Znamy już. Koalicja Obywatelska, Platforma potrafi tylko jedno: krytykować. Ale też pamiętam dokładnie barszcz i mirabelki. Pewnie też pamiętacie, prawda? Rozwiązanie Donalda Tuska (Dzwonek), rozwiązanie rządu Platformy Obywatelskiej i PSL.

Panie i Panowie z PiS! Jesteście ekspertami w przeliczeniu, ile czego możemy kupić za średnią pensję. To spróbujmy z węglem. Przecież Polska węglem stoi. Wasz prezydent, wasz premier, ministrowie przekonywali, tak? Kopalnie węgla są pod waszym zarządem, pod butem. Czy jest chętny do przeliczania? Proszę podnieść rękę. Nie widzę. A może pani minister podniesie rękę i przeliczy? To zacznijmy z najniższą emeryturą, czy z najniższą emeryturą z ZUS-u, czy z KRUS-u, nie starcza na tonę. Nie przeliczymy na tony. Teraz na worki się kupuje.

Cofamy się do lat 50., 60. Jak tak będziecie rządzić, ludzie będą chodzić na tory. Dziadkowie mi to opowiadali, jak to było. Takie są ceny opału w tej chwili. Nie robicie z tym nic, nie macie zielonego pojęcia, jak tym zarządzać, nie macie pomysłu, jak pomóc ludziom. Żeby nie starczyło na tonę węgla? 33% ludzi w Polsce opala, grzeje się węglem. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wszystko wskazuje na to, że ubocznym skutkiem działań podejmowanych podczas pandemii, których celem było ratowanie przedsiębiorców przed bankructwem i ochrona miejsc pracy, jest dzisiejsza inflacja. Dotyczy to nie tylko Polski, ale także innych wysokorozwiniętych państw o silnej i stabilnej gospodarce, zarówno w Europie, jak i na świecie, zwłaszcza tych, które najlepiej poradziły sobie z wywołanym pandemią kryzysem gospodarczym. Są to np. Czechy, Niemcy, Rumunia, a nawet Stany Zjednoczone. Poziom inflacji w tych państwach jest porównywalny z naszym, a takiego wyniku nie odnotowano tam od kilkudziesięciu lat. Jeszcze go nie znamy, ale chciałbym zapytać, czy zawarte w nim rozwiązania pokrywają się z działaniami prowadzonymi przez rządy innych państw dotkniętych inflacją (Dzwonek) i jakie są najbliższe prognozy. Bardzo dziękuję. Pytanie zada pani poseł Monika Wielichowska. Wysoka Izbo! Chcę dziś upomnieć się o medyków, którzy przy już czwartej fali pandemii są na pierwszej linii frontu walki z COVID. Rząd ich nie słucha. Białe miasteczko działa już 67 dni. Medycy biją na alarm od wielu miesięcy. Publiczna służba zdrowia umiera, wszyscy to widzimy. Z pracy ze względu na niskie pensje i ignorancję rządu odchodzą lekarze i pielęgniarki. Medycy nie chcą już waszych oklasków, chcą godnego wynagrodzenia za swoją ciężką pracę. Gdzie jest premier? Gdzie jest minister zdrowia? Może walczą z COVID-em? Otóż nie.

Na koniec trochę faktów.

Proszę o zabranie głosu pana posła Jana Warzechę. Wysoka Izbo! Ze strony opozycji padają zarzuty, że nic się nie robi w sprawie inflacji. Otóż Narodowy Bank Polski zareagował na skok inflacji, podwyższając kolejno stopy referencyjne. Na początku listopada podwyższył je do 1,25%. Rząd również nie bagatelizuje tego zjawiska i aktualnie intensywnie pracuje nad pakietem antyinflacyjnym. Aktualnie także w USA inflacja jest wysoka i wynosi 6,2%, licząc rok do roku, a w Niemczech sięga 5%. Odnosząc się do troski opozycji, pana posła Nitrasa, o wynagrodzenia w budżetówce, należy przypomnieć, że nie kto inny jak ekipa Donalda Tuska zamroził w 2011 r. na wiele lat pensje w tym sektorze.

Proszę o zabranie głosu pana posła Tomasza Szymańskiego. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Należy pochylić się nad problemem cywilnych pracowników komend powiatowych Policji i komend miejskich Policji nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń. Nie wiem, czy państwo wiecie, że w Polsce jest to grupa blisko 25 tys. pracowników.

To 25 tys. osób, z czego blisko 60% ma najniższe wynagrodzenie. Szanowni Państwo! Nie ma takiej możliwości, żebyśmy pominęli akurat tę część pracowników sfery budżetowej, tę część pracowników sfery mundurowej.

Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Pani Minister! Pracownicy korpusu służby cywilnej, wynagrodzenie - 3427 zł. Kiedy z tej trybuny im dziękujecie, nie myślicie o ich wynagrodzeniach, nie myślicie o Policji, nie myślicie o wojsku, nie myślicie o Straży Granicznej, a teraz - o rolnikach.

Zakupy maszyn. Jak ludzie na wsi, rolnicy mają żyć? Nie ma grup zakupowych, o których mówicie. Nie ma możliwości kupienia tańszego paliwa.

Bardzo dziękuję. Chciałbym poinformować Wysoką Izbę, że pani marszałek Sejmu zwołała na godz. 12.45 posiedzenie Prezydium Sejmu i Konwentu, na które będę musiał pójść, zatem gdzieś ok. godz. 12.40 ogłoszę kilkuminutową przerwę. Postaram się przyjść jak najszybciej. Proszę pana posła Grzegorza Wojciechowskiego. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Słyszę tutaj dramatyczne apele z lewej strony sali.

Nie bardzo rozumiem, skąd te takie dramatyczne apele.

Postaram się jak najszybciej wrócić.

Kontynuujemy rozpatrywanie punktu 17. porządku dziennego: Informacja bieżąca. Bardzo proszę pana posła. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

To jest informacja z wczorajszego dnia. W historii Polski nigdy takich kontraktów nie było, nigdy nie było takich cen, a ponoć mamy energię pochodzącą z polskiego węgla (Dzwonek), taniego polskiego węgla oraz z polskich elektrowni. O gazie już nie wspomnę, bo tam cena poszybowała kwartalnie, z kwartału na kwartał o 140%. Jest podstawowe pytanie: Co rząd robił przez ostatni rok, przez ostatnie miesiące, kiedy mówiliśmy o tym, że trzeba ograniczyć VAT, chronić 2 mln Polaków żyjących w skrajnej biedzie? Mówiła o tym Platforma, mówiła o tym również Komisja Europejska. Brak i bezradność polskiego rządu w chronieniu Polaków. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu panią poseł Annę Dąbrowską-Banaszek. Jeżeli nie ma, to pan poseł Tomasz Kostuś.

Ale ja nie poganiam pana posła. Szanowna Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W strukturach Policji obecnie zatrudnionych jest 25 tys. pracowników cywilnych, z czego 26% otrzymuje wynagrodzenie poniżej najniższej pensji krajowej, wynoszącej - przypominam - 2800 zł.

Brawo, tak, brawo, ja też się do tych braw dołączam, ale proszę nie zapominać, że pracownicy cywilni otrzymali jedynie 167 zł podwyżki. W kontekście galopujących cen i inflacji, która drenuje kieszenie Polaków, jest to niezrozumiałe, jest to nie do przyjęcia, jest to kuriozalne, panie pośle. Proszę o tym pamiętać, jak tak bije pan brawo. Przypominam również, że w październiku br. [[Dzwonek]] Porozumienie Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji wystąpiło w tej sprawie z 14 postulatami. Do dzisiaj nie otrzymali odpowiedzi. Kończąc, panie marszałku, dwie sprawy. Apeluję do pani minister - patrzę, czy jest, jest - by podjęła pilne i kompleksowe działania zmierzające do poprawy sytuacji pracowników cywilnych Policji. To po pierwsze. Po drugie, bardzo proszę, pani minister, o przedstawienie kompleksowej informacji na temat planowanych zmian wynagrodzeń dla pracowników cywilnych. Jak państwo widzicie, nie ograniczam nikomu głosu, ale lista posłów zapisanych do zabrania głosu jest bardzo długa i proszę o streszczanie się. Teraz bardzo proszę o zabranie głosu panią poseł Annę Kwiecień, a następnie głos zabierze pan poseł Czesław Siekierski.

Panie Marszałku! Inne obowiązki mnie wzywają, a chciałem odnieść się do bardzo ważnej sprawy związanej z sytuacją dochodową, jeśli chodzi o rolnictwo. Wzrost kosztów produkcji jest tak ogromny, jeśli chodzi i o sprawy środków produkcji, i o nawozy, i o paliwa, energię, że zagraża to możliwości utrzymania produkcji i jej otworzenia w latach następnych. A więc będzie to miało konsekwencje w obniżeniu poziomu produkcji w roku przyszłym. Oczywiście można trochę tak żartobliwie powiedzieć, że przyczyni się to do realizacji zielonego ładu, ale nie o taki ład nam chodzi, który by zmniejszył produkcję i zagroził bezpieczeństwu żywnościowemu.

Chodzi tu o emerytów, chodzi tu o bezrobotnych. Jakie będą świadczenia, które by przeciwdziałały tej sytuacji, poszerzającemu się ubóstwu i biedzie wśród znacznej części społeczeństwa? Proszę o zabranie głosu pana posła Czesława Mroczka. Panie Marszałku! W wyniku szokująco błędnych decyzji rząd PiS doprowadził do gigantycznych szkód w energetyce. Straty, szkody są wielomiliardowe.

Rząd PiS przez długi czas nie podejmował działań, które zahamowałyby inflację, ponieważ korzystał z tej inflacji. Te pieniądze oczywiście były kierowane na realizację partyjnych celów. Rząd zapominał o sferze budżetowej, na której opiera się sprawne funkcjonowanie państwa. Chcę wspomnieć o nauczycielach, bo sytuacja, kondycja materialna nauczycieli jest tak dramatyczna, że w zawodzie brakuje w tej chwili (Dzwonek) nowych osób, brakuje nauczycieli. Nie ma, proszę państwa, dobrej przyszłości kraju bez dobrego systemu edukacji. W tej sprawie jest potrzebne pilne działanie. Ale rząd nie myśli o państwie, rząd PiS nie myśli o sferze budżetowej. Rząd PiS myśli o własnych interesach wyborczych. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana posła Pawła Rychlika. Jeżeli nie ma, to pani poseł Krystyna Sibińska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Oferty pracy: inspektor w wydziale - 3106 zł, starszy referent zespołu stanowiska kierowania - 2861 zł, wynagrodzenie zasadnicze brutto, starszy księgowy do spraw obsługi świadczeń socjalnych w wydziale finansów i budżetu - 3670 zł, inspektor do spraw kancelaryjnych i archiwum w wydziale do spraw ochrony informacji niejawnych - 3050 zł. To są oferty pracy w Policji dla pracowników cywilnych. Czy to są godne warunki pracy? Czy to są godne warunki płacy? Nie, dlatego że pracownicy cywilni piszą do nas. Piszą o tym, że są grupą najniżej zarabiającą nie tylko w resorcie spraw wewnętrznych, ale również w całej sferze budżetowej. Nie mają tych samych uprawnień ani uposażeń co funkcjonariusze. Obecna sytuacja pracowników Policji jest dramatyczna, dlatego piszą do nas: „Prosimy o pomoc posłów Rzeczypospolitej” Proszę o zabranie głosu pana posła Michała Gramatykę. Wysoki Sejmie! Polsce nie grozi inflacja, krąży nad nami raczej widmo deflacji, tak sobie śmieszkowali pan prezes Narodowego Banku Polskiego i pan premier nieco ponad rok temu. Potem oczywiście prezes NBP zmienił zdanie, bo w lipcu br. zapowiadał już 4% inflacji z tendencją spadkową przez kolejne lata. Jednak rzeczywistość jest bezlitosna - wzrost cen raportowany w październiku tego roku sięga 7%, a miesiąc do miesiąca ceny rosną o 1 punkt procentowy. Z planowaniem w horyzoncie krótkoterminowym pan prezes Glapiński też ma niejakie problemy. Podwyżka stóp procentowych byłaby szkolnym błędem - mówił pan prezes w październiku, czyli niecały miesiąc przedtem, zanim dokonał jednej z największych w ostatnich latach podwyżek stóp procentowych.

Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana posła Andrzeja Kryja. Wysoka Izbo! Wielokrotnie na tej sali mówiono o wzroście cen energii elektrycznej i o wpływie tego zjawiska na inflację. Rzeczywiście, szanowni państwo, ceny energii elektrycznej rosną, a bardzo istotny wpływ na to ma wzrost cen uprawnień do emisji CO2. Te ceny uprawnień zaczęły rosnąć w momencie, kiedy został ogłoszony zielony ład. Skutkowało to tym, że ceny z poziomu dwudziestu kilku euro przekroczyły 50 euro, co miało miejsce w czerwcu 2021 r., a po 2 miesiącach przekroczyły już 60 euro. Mówi się o tym, że one sięgną nawet 100 euro. 15% ceny energii elektrycznej to ceny uprawnień do emisji CO2 Mam pytanie: Czy na poziomie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego prowadzone są prace, które doprowadzą do tego, że te absurdalnie wysokie ceny uprawnień do emisji CO2 zostaną ograniczone, zostaną zatrzymane? Proszę o zabranie głosu pana posła Marka Rząsę. Wysoka Izbo! Według polityków PiS kryzys gospodarczy, galopująca inflacja, drożyzna, wysokie ceny paliwa, drastyczny wzrost opłat za gaz i prąd, łupienie polskich przedsiębiorców, których macie za cwaniaków, to są tylko suche liczby, a w zasadzie to jest coś pozytywnego, bo oto zwiększają się wpływy do polskiego budżetu. Będziecie mieli więcej środków na swoje fundacje, stowarzyszenia, na megalomańskie projekty rodem z PRL-u, na TVP i na jej ohydną propagandę.

Pytam w imieniu swoich koleżanek i kolegów nauczycieli, w imieniu pielęgniarek, a także w imieniu wszystkich pracowników szeroko pojętej sfery budżetowej, bez których funkcjonowanie państwa jest w zasadzie niemożliwe. Ale wbrew temu, co mówił premier Morawiecki, Polacy nie pozwolą na wygaszanie ich aspiracji, a zwłaszcza ci pracujący w sferze budżetowej. Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Padło tu pytanie o ceny węgla i sytuację na rynku węglowym.

O ile w Polsce mamy sytuację czysto spekulacyjną, o tyle na rynkach europejskich i światowych mamy sytuację związaną z po-COVID-em, czyli napędzaniem gospodarki zwiększonym popytem, ale także polityką państwa rosyjskiego i utworzeniem nitki gazowej, co będzie odbijało się czkawką na rynkach energetycznych. Dziękuję bardzo. Czy na sali jest pan poseł Dariusz Rosati? Nie ma. Zatem pani poseł Ewa Szymańska.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Podziwu godna jest troska dzisiejszej opozycji o ludzi zagrożonych ubóstwem, szczególnie w sferze budżetowej. Mam pytanie: A co państwo zrobiliście, żeby w sferze budżetowej były wyższe wynagrodzenia? To za waszych rządów płace były zamrożone. To za waszych rządów dzieci chodziły głodne.

Pytanie zada pani poseł Zofia Czernow. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Chciałam zwrócić uwagę Wysokiej Izby i upomnieć się o pracowników cywilnych Straży Granicznej.

Nie można tak rozwarstwiać wynagrodzenia pracowników, którzy wykonują te same zadania. Do czego tu dojdzie? Bardzo proszę, aby w budżecie uwzględnić te rozbieżności, tę niesprawiedliwość. Bardzo dziękuję, pani poseł. Szanowny Panie Marszałku! Państwo Ministrowie! Poseł Warzecha podsumował dobitnie tragiczne dla Polski rządy Platformy Obywatelskiej i PSL, więc nie będziemy już wracać do tego, co zostało powiedziane. Jednak chciałbym również zwrócić uwagę państwa posłów z opozycji na to, że tendencje wzrostowe w zakresie inflacji obserwowane są na całym świecie, również w większości państw Unii Europejskiej, niezależnie od polityki krajowej prowadzonej tu, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Jesteśmy dziś wszyscy mieszkańcami globalnej wioski.

Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana posła Arkadiusza Marchewkę. Jeżeli nie ma, to pan poseł Tadeusz Woźniak. Też nie ma. Zatem proszę panią poseł Mirosławę Nykiel. Pani Minister! Inflacja to drugie imię PiS-u, a drożyzna - premiera Morawieckiego. To właśnie on w 2013 r. mówił, że ludzie powinni obniżyć swoje oczekiwania i pracować, powiem ładnie, za przysłowiową miskę ryżu. Pytam, panie premierze: Czy to już jest ten moment, aby 25 tys. pracowników służby cywilnej Policji pracowało za przysłowiową miskę ryżu?

Mówicie, że nie macie pieniędzy. Ustalcie zeznania. Bo raz mówicie, że macie niezmierzoną wręcz ilość pieniędzy i cały świat was podziwia i stoi w kolejce, a jak trzeba dać podwyżki sferze budżetowej, to was na to nie stać. A może wystarczy nie kraść? Teraz głos zabierze pani poseł Anna Ewa Cicholska. Dziękuję. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Szanowni Państwo! Państwo parlamentarzyści opozycji! Doskonale państwo wiedzą, że mamy trudną sytuację na granicy polsko-białoruskiej i czwartą falę pandemii. Cały czas wprowadzacie opinię publiczną w błąd, dezorganizujecie życie publiczne. Inflacja dotyczy wszystkich państw Unii Europejskiej, całego świata. Doskonale państwo wiedzą, czym jest spowodowana.

Szanowna Pani Minister! Mam pytanie: Jakie działania podejmują poszczególne ministerstwa (Dzwonek), rząd w celu zminimalizowania skutków inflacji? Bardzo dziękuję. Proszę panią poseł Gabrielę Lenartowicz. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 27 października na konferencji prasowej został ogłoszony plan modernizacyjny, także dla służb mundurowych.

Tabele wynagrodzeń sięgają dużo poniżej najniższej krajowej, więc prawie wszyscy równo otrzymują tę najniższą. Chcę upomnieć się o to w imieniu m.in. pracowników Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, ale nie tylko.

Bardzo dziękuję. Głos zabierze pan poseł Włodzimierz Tomaszewski.

Ale wtedy, kiedy państwo rządziliście, nie słyszałem takich wystąpień. Nie słyszałem.

Szanowni Państwo!

Pokażę państwu, bo to jest bardzo interesujące. Przecież państwo oszaleli.

Szanowny Panie Marszałku! Drogie Posłanki i Posłowie! Czy pani wie może, co to za kraj, w którym młodzi, ambitni ludzie idą na 5-letnie studia, kończą administrację z tytułem magistra, trafiają do pracy w regionalnej izbie obrachunkowej i dostają 2360 zł? Albo trafiają do pracy w Państwowej Inspekcji Handlowej, gdzie 1/4 pracowników zarabia 3240 zł brutto. Ja pani minister powiem, co to za kraj. To kraj, w którym elity złożone z młodych ludzi, którzy chcą być urzędnikami, niestety stają się nędznikami, ponieważ te wynagrodzenia są dramatycznie za niskie, niepozwalające na przyzwoite życie, niepozwalające na samorozwój i de facto podcinające skrzydła tym wszystkim ambitnym osobom. W jaki sposób to państwo ma być efektywnie zarządzane? W jaki sposób ono ma dobrze funkcjonować, jeżeli nie dbacie o własne elity urzędnicze, o własnych pracowników inspekcji handlowej (Dzwonek) czy regionalnych izb obrachunkowych? Zamiast urzędników tworzycie w Polsce nędzników. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana posła Piotra Polaka. Panie Marszałku! Państwo Ministrowie! Polska nie jest czerwoną wyspą na mapie Europy czy świata i nie tylko w Polsce jest inflacja, i nie tylko w Polsce mamy wzrost cen. Wiele czynników na to wpływa i nie będziemy teraz tych czynników analizować. Ale, szanowni państwo, można stać obok tego, ale można też coś z tym tematem robić. Polski rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego nie stoi z założonymi rękoma, tylko pochyla się nad tym problemem.

Chciałbym zapytać pana ministra, jakie jeszcze inne działania osłonowe dla konsumentów (Dzwonek), dla Polaków przewiduje rząd w najbliższym czasie. Pytanie zada pan poseł Czesław Hoc. Pani Minister! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Do wnioskodawców z opozycji: Czy pamiętacie dzieci odbierane od biologicznej rodziny tylko z powodu biedy? Albo głodne dzieci w szkołach? Czy pamiętacie dokonywanie podstawowych zakupów w sklepach na wsiach i w małych miasteczkach na tzw. zeszyt albo na kreskę? Czy pamiętacie dramatyczne momenty, że co trzeci pacjent, głównie spośród seniorów, odchodził od okienka aptecznego, bo nie stać go było na wykupienie leków? Czy pamiętacie skandaliczny wykup polskiej ziemi przez tzw. słupy i kapitał zagraniczny? Szanowna opozycjo, wy macie odwagę i czelność zarzucać obecnemu rządowi politykę zubożenia społeczeństwa? Przecież za waszych rządów była strategia: pieniędzy nie ma i nie będzie. A my sukcesywnie wzmacniamy potencjał rodziny, przywracamy godność pracownika, inwestujemy w dzieci i prowadzimy konkretną politykę senioralną. Pytanie zada pan poseł Jarosław Krajewski.

Wysoka Izbo! Temat inflacji jest dla nas tematem ważnym, nie uciekamy przed taką dyskusją jako parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, ale chcemy rzetelnie rozmawiać w tym miejscu na temat faktów, a fakty są takie, że w ostatnich 5 latach zawsze wzrost wynagrodzeń przewyższał poziom inflacji.

Gdyby wtedy rządziła Platforma i nie było tych świetnych programów polityki rodzinnej, „Rodzina 500+”, wyprawka „Dobry start” czy kwestia podwyższonych świadczeń społecznych, czy kwestia wzrostu płacy minimalnej. Mam pytanie do pani minister i do pana ministra: Chciałbym, żebyście państwo poinformowali, kiedy rząd przedstawi projekt tarczy antyinflacyjnej i czy pani minister ma takie informacje, że w samorządach, np. w najbogatszym samorządzie w Polsce w Warszawie, jest przygotowywany jakikolwiek pakiet antyinflacyjny. Jeżeli mamy Rafała Trzaskowskiego, wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej, to mógłby przedstawić choć jedną państwa propozycję antyinflacyjną w samorządzie warszawskim. O to pytają mnie mieszkańcy Warszawy i to jest dla warszawiaków ważne. Państwo macie z tym problem. Rozumiem, zostawiam państwa z tym problemem. Dziękuję panu, ale mam wrażenie, panie pośle, że dzień bez Rafała Trzaskowskiego to dzień stracony. Na tym lista osób zapisanych do pytań została wyczerpana. Bardzo teraz proszę. Czy pan poseł jeszcze o Rafale Trzaskowskim? Czy pani poseł Leszczyna upoważniła panią Skowrońską do zabierania głosu?

Panie Marszałku! Państwo Ministrowie! Otóż mieliśmy dyskutować o inflacji, czyli drożyźnie, i wynagrodzeniach w sferze budżetowej, o pensjach nauczycieli, pielęgniarek, cywilnych pracowników Policji, urzędników, pracowników sądów, prokuratur, a państwo mówiliście kompletnie od rzeczy i nie na temat. Wystąpienie pani minister i posłów PiS-u rzeczywiście niebezpiecznie korelowało ze słowami premiera Morawieckiego, który powiedział kiedyś, że ludzie powinni pracować za miskę ryżu. Ja pominę milczeniem ten wulgaryzm, którego premier zwykł używać. Otóż słowa Morawieckiego okazały się prorocze. No i pewnie dlatego wystąpienie pani minister było poświęcone zasiłkom, nie wynagrodzeniom. Rzeczywiście jest tak, że w czasie rządów PiS-u [[Oklaski]] urzędnicy, pracownicy administracji publicznej stali się ekonomicznymi pariasami, i rzeczywiście jest tak, że politykę socjalną PiS-u, bo pani minister o niej mówiła, da się połączyć z inflacją, bo wszystkie plusy, które miały uczynić z Polski krainę mlekiem i miodem płynącą, „Mieszkanie+”, 500+, nawet krowa+, skumulowały się w jednym wielkim plusie - to jest drożyzna+. To jest jedyny projekt rządu PiS, który wam się udał. Udał się rządowi, bo będziecie mieli kilkanaście miliardów złotych więcej w budżecie w tym roku, a w przyszłym pewnie kilkadziesiąt miliardów więcej, natomiast niestety to jest porażka dla wszystkich podatników, konsumentów, to jest haracz, jaki ściągacie od kilku lat z Polaków. Powtórzę: od kilku lat. Więc jak państwo pytacie, czy to prawda, że przyczyny inflacji są zewnętrzne, czy to prawda, że to polityka luzowania ilościowego banku centralnego spowodowała inflację, czy to prawda, że to kryzys energetyczny jest winny, to ja wam powiem: nie, winien jest nieodpowiedzialny, awanturniczy rząd PiS-u i winien jest niewiarygodny prezes Narodowego Banku Polskiego, [[Oklaski]] który zrujnował swoją reputację i reputację banku centralnego. I nie macie prawa mówić o tym, że my mroziliśmy wynagrodzenia, co najmniej z trzech powodów. Dlaczego? Po pierwsze, jak mroziliśmy wynagrodzenia w budżetówce, to nie podnosiliśmy wynagrodzeń sobie, [[Oklaski]] a jedyne nagrody przez 8 lat to były nagrody dla czterech ministrów, i to po jednej nagrodzie. Więc nie macie prawa mówić o tym, że mroziliśmy. Po drugie, mniej boli mrożenie pensji, jak mamy do czynienia z bardzo niską inflacją albo wręcz z deflacją, a tak było za naszych czasów. A inaczej boli mrożenie, jak mamy galopującą drożyznę. Ostatnia rzecz: w czasie naszych rządów mieliśmy dwa poważne kryzysy, a bezrobocie, panie pośle, jak u nas było 14%, to w Hiszpanii było 28%. Więc proszę nie opowiadać tu głupot. Natomiast wy mieliście 4 lata świetnej koniunktury. I wy porównujecie wynagrodzenia w sferze budżetowej z tymi z naszych czasów? Wstydźcie się. A więc posłuchajcie uważnie, kto jest winien inflacji w Polsce i szalejącej drożyzny. Dlatego, że doprowadziliście do zapaści w inwestycjach największej od 25 lat, pompowaliście wzrost gospodarczy konsumpcją, a nie inwestycjami, finansowaliście transfery socjalne długiem publicznym, kłamiąc, że to jest uszczelnienie podatków, podnieśliście 40 podatków i danin albo wprowadziliście nowe, bo w czasie pandemii wprowadzacie nowy ład, czyli podnosicie podatki dla producentów, a więc ceny znowu pójdą w górę, wreszcie przez 6 lat nie zrobiliście nic, żeby polepszyć miks energetyczny, wręcz przeciwnie zrobiliście wszystko, żeby miks energetyczny pogorszyć, wreszcie swoim awanturnictwem, kompleksami, chęcią zawłaszczenia sądów, żeby kryć własne przestępstwa, doprowadziliście do takiego konfliktu z Unią Europejską, że nie mamy pieniędzy z KPO i w tym roku nie skorzystają z nich ani pacjenci, ani uczniowie. ani samorządy, ani przedsiębiorcy. I wreszcie, dlaczego prezes Glapiński?

Bardzo dziękuję, pani poseł. Proszę o zabranie głosu podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów pana Piotra Patkowskiego. Panie Marszałku! Opozycja przedstawia obecną inflację, którą - jak tutaj mówili też posłowie Prawa i Sprawiedliwości - dostrzegamy, rozumiemy, o czym będę mówił jeszcze w dalszej części mojej wypowiedzi.

W ciągu tygodnia rząd, premier Morawiecki, przedstawi konkretne postulaty dotyczące tarczy inflacyjnej, pakietu osłonowego dla Polaków.

Dla mnie to jest patriotyzm. Jeżeli dla pana troska o polskie rodziny to jest PRL. Zawsze jak się tworzy pakiety rządowe, korzysta się z doświadczeń historycznych, to normalne. Wie pan jak? Nie mieliście żadnego pakietu osłonowego dla polskich firm w momencie, kiedy wybuchł kryzys finansowy.

Mało tego, szanowni państwo. Tak, to jest państwa odpowiedź na inflację: podwyżka VAT w roku 2011. I jeszcze jedno: państwo ani razu - ani razu - od roku 2009 nie osiągnęliście konsolidacji finansów publicznych. W każdym roku państwa rządów deficyt przekraczał 3% i to za waszych rządów mimo rekordowego bezrobocia, jeśli chodzi o porównanie kryzysów, jeśli chodzi o brak tarcz osłonowych dla przedsiębiorców, mieliście państwo rekordowe bezrobocie i rekordowe deficyty. To jest państwa odpowiedź na inflację.

Przypomnę, że inflacja także była jednym z elementów.

Procentowy wzrost?

Odtworzenie funduszu nagród dla państwowej sfery budżetowej z możliwością wykorzystania także w przyszłym roku - 6%.

Warto także powiedzieć. Państwo bardzo lubicie prognozy Komisji Europejskiej, to je przytoczę.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 18. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Polskiego Romantyzmu (druki nr 1347 i 1578) Proszę panią poseł Joannę Lichocką o przedstawienie sprawozdania komisji.

Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu na temat poselskiego projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Polskiego Romantyzmu.

Pod tą petycją podpisało się 51 profesorów z uniwersytetów z całej Polski oraz Instytutu Badań Literackich. To są reprezentanci takich ośrodków akademickich jak Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Gdański czy Uniwersytet Rzeszowski. Jest to rzeczywiście wielka reprezentacja wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, polskiej humanistyki, którzy zwrócili się do parlamentu o ustanowienie tego roku. Poparcie dla tej inicjatywy wyrazili również - w odrębnych pismach do marszałek Elżbiety Witek - dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie oraz dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Ich twórczość, twórczość romantyków wyrastała organicznie z dziedzictwa pierwszej, wielonarodowej Rzeczypospolitej. Rok 2022 powinien stać się okazją do odczytania na nowo najwybitniejszych utworów tamtej epoki, a przede wszystkim do postawienia pytania o ich aktualność i znaczenie dla nas teraz. Komisja petycji pracowała nad petycją, o której mówiłam, która powstała z inicjatywy prof. Andrzeja Fabianowskiego, i przesłała ten materiał do komisji kultury. Była to jedna z podstaw opracowanego tekstu uchwały. Powiem państwu, że praca nad tym projektem w komisji kultury nie budziła kontrowersji i była właściwie samą przyjemnością. Chciałabym przeczytać tekst tej uchwały ponieważ komisja kultury po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu na posiedzeniu w dniu 17 września 2021 r. wnosi, aby Wysoki Sejm uchwalić raczył ten projekt. W 1822 roku w Wilnie ukazały się 'Ballady i romanse' Adama Mickiewicza, zawarte w tomiku poetyckim, który wyznaczył początek polskiego romantyzmu. Wtedy po raz pierwszy ujrzały światło dzienne 'Romantyczność', 'Powrót taty', 'Świtezianka', 'Pani Twardowska', bez których trudno wyobrazić sobie ostatnich dwieście lat polskiej kultury. To, co nastąpiło potem, było bez precedensu w polskich dziejach. Zrodziła się epoka, w której tworzyli genialni artyści, myśliciele i działacze polityczni, którzy w sytuacji narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności, rozwinęli programy niepodległościowe, a zarazem wynieśli polską literaturę, muzykę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury europejskiej. Romantyzm przyniósł genialne dokonania w literaturze Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego i Cypriana Norwida, w muzyce Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki, w malarstwie Piotra Michałowskiego i Jana Matejki. Twórcy ci byli artystami polskimi, a jednocześnie światowymi, ukazującymi polskie wartości w ich uniwersalnym kontekście. Bez twórczości ich oraz Maurycego Mochnackiego, Aleksandra Fredry, Antoniego Malczewskiego, Seweryna Goszczyńskiego, Wincentego Pola, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Teofila Lenartowicza, Kornela Ujejskiego, Artura Grottgera, Marii Szymanowskiej i Narcyzy Żmichowskiej nie bylibyśmy dziś tym, kim jesteśmy. Literatura i kultura polskiego romantyzmu ukształtowały wymiar i profil duchowy Polaków. Wypracowane i utrwalone zostały najważniejsze cechy pozwalające nam przetrwać nawet najdramatyczniejsze próby zniszczenia narodu. Honor, waleczność, patriotyzm, przywiązanie do tradycji, empatia wobec losu innych i gotowość do ofiar, otwartość na inne kultury oraz przywiązanie do wolności - ten kanon wartości narodowej wspólnoty romantyzm przeniósł z dawnej Rzeczypospolitej i zdefiniował na nowo. Bez Maurycego Mochnackiego i jego pism o wolnych Polakach, bez wieszczów Mickiewicza i Słowackiego, pochowanych w królewskich kryptach, bo Polacy uznali, że królom Polski są równi, nie byłoby Legionów Piłsudskiego czy Powstańców Warszawskich. To z romantyzmu wyrósł nowoczesny mesjanizm Jana Pawła II i unikatowy w dziejach światach ruch 'Solidarność' Pamięć romantyzmu polskiego jest zatem pamięcią najważniejszych znaków określających narodową tożsamość. W roku 2022 przypadają dwusetne urodziny tej epoki i jest to dobry powód do przypomnienia duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - odpowiadając na petycję 51 badaczy romantyzmu reprezentujących Polską Akademię Nauk i wszystkie ośrodki akademickie w kraju oraz spełniając apel środowisk skupionych w Akademickich Klubach Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego - ogłasza rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego” Wydaje mi się, że jest zupełna zgoda wszystkich ugrupowań i ta uchwała może zostać przyjęta jednomyślnie. Bardzo dziękuję. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jako pierwsza głos zabierze ponownie - więc nie jako pierwsza, ale jako pierwsza z katalogu występujących w imieniu klubu - pani poseł Joanna Lichocka. Wysoki Sejmie! W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość oczywiście chciałabym powiedzieć, że popieramy tę uchwałę. Rok romantyzmu jest nam wszystkim bardzo potrzebny po to, żeby przypomnieć sobie te postacie, które stworzyły nasz współczesny, nowoczesny język i nasze współczesne, nowoczesne myślenie o Polsce, o wolności, o rzeczywistości. Maurycy Mochnacki, polityk, publicysta, żołnierz, krytyk literacki, pisał m.in. tak: Nie dosyć na tem, że jesteśmy, potrzeba to jeszcze wiedzieć. Im lepiej to wiemy, tem bardziej rozszerzamy się, umacniamy w jestestwie naszem. Kto jest, a nie ma uznania samego siebie, czyli kto tego, że jest, nie wie, ten jest tak, jakby go wcale nie było. To właśnie ta epoka romantyzmu, ci nasi wielcy, genialni twórcy, artyści, politycy, malarze, filozofowie, politycy ustanowili nas w jestestwie naszym na kolejne dekady i wieki. Warto o nich pamiętać, warto o nich dyskutować, a ponowne przemyślenie naszej tożsamości, kultury, korzeni może być zadaniem Roku Romantyzmu Polskiego, aby uznać się w jestestwie swoim ponownie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę teraz pana posła Krzysztofa Mieszkowskiego o zabranie głosu i przedstawienie stanowiska Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska.

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Klub Koalicji Obywatelskiej oczywiście poprze tę uchwałę, bo ona jest nam bardzo potrzebna do tego, żebyśmy mogli naszą „dzisiejszość” móc weryfikować przez idee romantyków, przez ich kondycję ludzką, przez ich polityczność. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz w sposób bardzo dobitny, jednoznaczny. Nie mam żadnych wątpliwości, że uchodźcy i emigracja polskich artystów, Mickiewicza, Krasińskiego, Szopena, Słowackiego, Norwida weszła w krwiobieg polskiej kultury. To jest w pewnym sensie paradygmat naszego systemu wartości. I dzisiaj trudno sobie wyobrazić, by było inaczej. Warto przypomnieć, że Adam Mickiewicz III część „Dziadów”, a więc popowstańczą refleksję na temat tego, co się wydarzyło w Polsce, napisał w Dreźnie, dzisiaj powiedzielibyśmy, że w Niemczech. Juliusz Słowacki „Kordiana” pisał w Genewie, wydał go w Paryżu, a więc również na uchodźstwie. Można mnożyć przykłady tych wszystkich wielkich dzieł, które dzisiaj kształtują naszą świadomość i naszą wyobraźnię. Przytoczę fragment książki Aliny Witkowskiej „Cześć i skandale” o migracyjnym doświadczeniu Polaków. To jest niezwykle ważna książka, która może jest nieco zapomniana, ale w kontekście dzisiejszych wydarzeń, zwłaszcza w kontekście wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej, może warto przypomnieć fragment tej książki. Witkowska pisze: Otóż droga, którą zmierzało się ku Francji, bo właśnie ona była początkowo docelowym krajem emigrantów, odegrała istotną rolę w ukształtowaniu się świadomości uchodźców i ich wewnętrznego samopoczucia, albowiem znaczna część byłych powstańców odbywała triumfalny pochód przez Niemcy. Wszędzie niemal znajdowali ludność usposobioną entuzjastycznie, nierzadko witały ich bramy triumfalne, a komitety organizacyjne na trasie przemarszu prześcigały się w bankietach ku czci bohaterów, zaopatrzeniu pieniężnym i zapewnieniu wygodnego wypoczynku. Triumfalny przemarsz przez Niemcy miał dalekosiężne i wielorakie skutki dla formowania się polskiej emigracji. W sferze idei politycznych utrwalił przekonanie o solidarności ludów Europy, o rychłości wybuchu rewolucyjnego i gotowości Niemców - z wyłączeniem Prus - do przelania krwi za wolność. W sferze psychiczno-mentalnościowej zaś entuzjazm Niemców skutecznie przeciwdziałał powstaniu kompleksu „nieproszonych gości”, natrętnych tułaczy, którzy nachodzą czyjeś spokojne domy, prosząc o wsparcie. Bardzo dziękuję panu posłowi. Stanowisko klubu parlamentarnego Lewica przedstawi pani poseł Paulina Matysiak. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu parlamentarnego klubu Lewicy mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Polskiego Romantyzmu. Romantyzm jest dla Polski szczególnie istotnym nurtem w dziejach, który nie tylko ukształtował naszą narodową kulturę, ale także wycisnął ogromne piętno na szeroko rozumianej myśli politycznej. Romantyzm przybywa do Polski w wyjątkowym okresie, kiedy formalnie nie istnieje polskie państwo, a polskie ziemie znajdują się pod rządami trzech zaborców. Nurt, który stawia w centrum dominację uczucia nad rozumem, który eksponuje indywidualizm i odmienność jednostki poprzez jej opór wobec zastanej rzeczywistości i ciasnego gorsetu krępujących norm, trafia na bardzo podatny grunt młodej inteligencji zniewolonego narodu. Pasja, uczuciowość, bunt wobec oświeceniowego porządku, mistycyzm i mesjanizm splatają się w nierozerwalną nić, która staje się językiem wyrazu nie tylko osobistych emocji i przeżyć jednostki, romantycznego bohatera, artysty, ale jednocześnie staje się także językiem wyrazu aspiracji i dążeń do wolności narodowej, samostanowienia wspólnoty politycznej, tęsknoty za utraconą ojczyzną i gotowością do poświęcenia siebie w imię większego celu. Romantyzm ukształtował kanon naszej literatury i wywarł ogromny wpływ na myśl narodowowyzwoleńczą. Wystarczy wspomnieć dorobek pisarski Adama Mickiewicza czy Juliusza Słowackiego, malarstwo Jana Matejki czy muzykę Fryderyka Szopena. Romantyzm polski przyniósł także zapowiedź przyszłej walki o wolność i równość kobiet w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym, choćby w osobie Narcyzy Żmichowskiej i Koła Entuzjastek, które zakorzeniły na polskim gruncie myśl feministyczną. Myśl, która w przyszłości zakwita ruchem emancypacyjnym i doprowadza do uzyskania przez kobiety praw politycznych z początkiem XX w. Rok Polskiego Romantyzmu byłby jednak pustym gestem, zaledwie strzałem na wiwat, gdyby ograniczył się tylko do składania peanów na cześć przeszłości, a nie stał się przyczynkiem do dyskusji nad romantyczną spuścizną, która także dzisiaj wybrzmiewa w polskiej kulturze i naszej dzisiejszej myśli politycznej. Chciałabym, żeby rok 2022 był szansą na uczciwe, także krytyczne spojrzenie na minioną epokę wraz z jej dorobkiem, ale nie po to, by żar w piersiach rozpalony przez romantyków wygaszać, ale by zaprząc go do wyzwań XXI w. Zamiast więc ślepo hołubić straceńczy mesjanizm czy altruistyczne samobójstwo, niech romantyczna idea na nowo rozpali polską duszę w dążeniu do świata opartego na miłości, wolności, równości i solidarności międzyludzkiej. Niech ten romantyczny żar roznieci też płomień nadziei na zmianę w tej Izbie. Razem młodzi przyjaciele! W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele” Bardzo dziękuję, pani poseł. Teraz pan poseł Jarosław Rzepa przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska. Wysoka Izbo! Dorobek polskiego romantyzmu jest skarbnicą arcydzieł literatury i kultury narodu polskiego. Tacy poeci jak Adam Mickiewicz, poeta, dramaturg, publicysta, autor „Dziadów”, „Konrada Wallenroda”, „Pana Tadeusza”, czy Juliusz Słowacki, autor „Kordiana”, „Balladyny”, „Beniowskiego” - od lat 60. po koniec XIX w. - uznawani za wieszczów narodowych, twórców natchnionych, genialnych, proroczych, największych artystów narodu polskiego. Ta epoka jest w Polsce powszechnie uznawana za jedną z najciekawszych i najdonioślejszych ze względu na głębokie powiązanie z życiem człowieka.

Najistotniejszym elementem kultury, nad którym zapanował romantyzm, była literatura, jednak nie można twierdzić, iż twórczość romantyków to tylko literatura. Romantyzm został uznany za tak istotny, gdyż jest najściślej związany z życiem, z historią, która ma tak wielkie znaczenie dla Polaków. Epoka „Pana Tadeusza” wytworzyła pewien styl życia, postrzegania piękna, obcowania z elementami metafizycznymi. To także ogromne podkreślenie wartości duszy człowieka, a także konkretnych osobowości, indywidualności posiadających cechy, które rzutowały na całość wizji świata w romantyzmie. Świadczy o tym zdolność panowania nad umysłem, a nie tylko nad poszczególnymi dziedzinami kultury. Ten fakt podsuwa nam stwierdzenie, iż romantyzm zdołał narzucić określony typ zachowania nie tylko jednostce, ale także całemu społeczeństwu. Przy tak wielkim znaczeniu w zależności od różnych dziedzin życia nie sposób zapomnieć o dziełach epoki.

Wiemy także, że i one były przełomowe w dziejach Polski. Tu należy podkreślić tę spójność literacko-historyczną. Interesujące wydają się także odbiór i interpretacja twórczości romantyków przez późniejszych pisarzy i myślicieli. W czasie rozwoju kapitalizmu nie było miejsca dla miłosnych i duchowych uniesień, patriotyzmu, a pojęcia takie jak „mesjanizm” czy „prometeizm” zostały zapomniane. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - PSL, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści Marka Biernackiego chciałbym poinformować państwa, że oczywiście nasz klub będzie głosował za tą uchwałą. Bardzo dziękuję panu posłowi. Proszę teraz pana posła Artura Dziambora o przedstawienie stanowiska koła Konfederacja. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Można sobie przemyśleć czasy, w których romantyzm był omawiany w szkole, i przypomnieć sobie tamte dzieła i to, jak je wtedy rozważaliśmy, co o nich myśleliśmy, jak zmieniło się nasze postrzeganie tego przez okres dorosłości, ponieważ pamiętając tamte czasy, jesteśmy w stanie dzisiaj wystawić tym uczuciom, które nam towarzyszyły, pewną laurkę. Czyli jak miłość, to na śmierć, jak nienawiść, to również na śmierć. Te uczucia były stawiane ponad rozum niestety bardzo często. To były wzorce pokazywane wtedy, żeby nas uczyć, żeby nam pokazywać, że uczucia powinny być jak najsilniejsze. Walka o swoje, oczywiste, to, co teraz w jakiś sposób w pewnym sensie powinno towarzyszyć zawsze. Piękna rola poezji, złożoność postaci, postaci dramatyczne, które były zarazem dobre, jak i złe, które robiły rzeczy dobre, jak i złe, które za każdym razem pokazywały nam, że nie ma bohaterów zawsze krystalicznych, że mimo wszystko zawsze gdzieś znajdzie się jakiś błąd. Rzeczywiście przywiązanie romantyzmu do tej uczuciowej sfery, do snów, do mistycyzmu, do fantastyki, było czymś, co nas poruszało.

Z szacunku zagłosujemy oczywiście (Dzwonek) za, natomiast opinię pozostawiam państwu. Taka dygresja, że jednak kult jednostki towarzyszył chyba bardziej innym epokom niż romantyzmowi. Proszę bardzo pana posła Michała Gramatykę o przedstawienie stanowiska Koła Parlamentarnego Polska 2050. Wysoki Sejmie! O tym, jak wielka siła jest w dorobku polskiego romantyzmu, dobitnie przekonałem się w październiku tego roku w sali Filharmonii Narodowej. To był drugi etap przesłuchań XVIII Konkursu Chopinowskiego. Na scenie Bruce Liu, Kanadyjczyk, geniusz fortepianu, prestidigitator i czarodziej tego instrumentu. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że wygra on tę edycję konkursu.

Niemy zachwyt publiczności z całego świata, która pochłania każdy dźwięk, i ta przejmująca duma, że to jest nasze, że to jest polskie, że ci wszyscy ludzie przyjechali z całego świata do Warszawy, żeby usłyszeć dzieła Polaka, którego muzyka stała się wyznacznikiem tego, co idealnie piękne, specimenem elegancji, definicją polotu, synonimem rozmachu. Ta polska doskonała muzyka napisana we Francji, na uchodźstwie, zagrana przez Kanadyjczyka na włoskim fortepianie i refleksja, że w połowie XIX w. na koncercie w sali paryskiego konserwatorium ten sam utwór grany przez autora wywoływał podobny zachwyt, podobną ekscytację, budził polską dumę, poruszał głęboko ukryte struny i nie pozwalał zapomnieć o polskiej sprawie, którą tak skutecznie i tak bezdusznie tłumiła ówczesna polityka.

Koło poselskie Polska 2050 z wielką przyjemnością i z wielką dumą zagłosuje za tą uchwałą. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Przystępujemy do pytań. Jeżeli nie, zamykam listę posłów zapisanych do pytań. Ustalałam czas na zadanie pytania - 1 minuta. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Jan Szopiński, klub parlamentarny Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym wyrazić głębokie zdziwienie zaprezentowaną inicjatywą.

Czy Polacy w roku romantyzmu odzyskają pełną wolność, wolność zgromadzeń, wolność słowa oraz pełnię swobód obywatelskich, których zostali pozbawieni przez rząd Prawa i Sprawiedliwości? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi. Teraz pytanie zada pan poseł Rafał Adamczyk. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo!

W związku z tym, że jest to kolejna uchwała w sprawie objęcia patronatem roku 2022, cieszy fakt, że wszyscy popierają ten projekt. Bardzo dziękuję. Pytanie zada pan poseł Mirosław Suchoń. Uprzejmie dziękuję.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu panią poseł Iwonę Marię Kozłowską. Wysoka Izbo! Dzisiaj jesteśmy w trakcie kryzysu migracyjnego na granicy. Dziesiątki tysięcy niewinnych osób są wykorzystywane w sposób cyniczny przez Aleksandra Łukaszenkę po to, aby mógł on wzmocnić swoją władzę.

Uwielbiacie wspominać przeszłość. Uwielbiacie wracać do czasów świetności państwa polskiego, nie dostrzegając zupełnie przykrych historycznych doświadczeń. Czy humanitaryzm i dobre relacje na arenie międzynarodowej to pojęcia obce przedstawicielom Prawa i Sprawiedliwości?

Dziękuję bardzo. Chyba nie ma na sali pana posła Franciszka Sterczewskiego. Zatem poproszę o zabranie głosu pana posła Tomasza Olichwera. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Uchwały okolicznościowe, takie jak i ta procedowana dzisiaj, nie powinny wśród posłów wzbudzać żadnych negatywnych wątpliwości czy emocji, bo przecież ich intencją jest uczczenie ważnych i istotnych wydarzeń lub postaci znaczących dla naszej polskiej historii czy tradycji. Niestety jest jednak inaczej. Bardzo często przygotowywane przez posłów PiS-u projekty takich uchwał zawierają w treści informacje, mówiąc delikatnie, nie do końca zgodne z prawdą historyczną, czy też poprawnością polityczną. Nie będę wdawał się w szczegóły, państwo, a w szczególności członkowie komisji kultury doskonale wiedzą, o co mi chodzi. Ale chciałbym przy tej okazji wyrazić swój sprzeciw wobec upolityczniania takich uchwał. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Kaczyński! Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

A jednak prawie 200 lat temu, w erze wielkich mocarstw, a nie demokratycznych państw, ktoś im dał schronienie, pozwolił zostać. Nie słyszałam, by któryś z nich tworzył na mrozie w lesie. Gdyby zostali tak potraktowani jak dwa wieki później my traktujemy ludzi ze Wschodu, to czy powstałyby słynne Chopinowskie mazurki, z których jesteśmy dumni na cały świat? Czy Mickiewicz stworzyłby „Pana Tadeusza”, czy jego Konrad mógłby wadzić się z Bogiem? Pamiętajmy, że tam na mrozie przebywają, kto wie, czy nie mniej zdolni poeci z Syrii, Kurdystanu i Iraku. Bardzo dziękuję. Głos zabierze pan poseł Marcin Porzucek.

Wydawało się, że trudno znaleźć projekt, który powinien łączyć bardziej niż ten, o którym właśnie teraz mówimy. A jednak okazało się, że dla dużej części posłów opozycji - Koalicji Obywatelskiej i Lewicy - to jest kolejna pałka, którą możecie państwo okładać polski rząd. To, że takie będzie wystąpienie pani poseł Jachiry, było czymś oczywistym, ale to, co robi pan Szopiński, pani Kozłowska. Jak państwu nie wstyd nawet w takim kontekście atakować polski rząd? w Polsce też tego nie wiedzą, czego świadkami byliśmy chociażby w ostatnich dniach - Fryderyk Chopin nie był uchodźcą. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę. Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Otóż Chopin był na uchodźstwie i tam do końca życia pracował i tworzył. Chcę państwu przypomnieć, że w 2016 r. dyrekcja Teatru Polskiego we Wrocławiu zwróciła się do pana prezydenta Dudy o honorowy patronat nad całością wystawienia „Dziadów” w naszym teatrze. Dzisiaj pan prezydent Duda jest wielkim zwolennikiem i orędownikiem jubileuszu, jeśli można użyć takich słów w stosunku do tej fantastycznej, wielkiej epoki. Warto jednak pamiętać i warto przypomnieć kilka drobnych faktów towarzyszących wielkiej twórczości naszych wybitnych artystów. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Romantyzm był piękną epoką, ale i trudną. Myśl romantyczna, dorobek artystyczny były bardzo ważne nie tylko w XIX w., ale rzutowały na kolejne dziesięciolecia, w kolejnych dziesięcioleciach na sztukę i wydarzenia historyczne w Polsce. Romantyzm w Polsce nie skończył się w XIX w., a postawa mesjanistyczna i też martyrologiczna wciąż obecna jest w społecznej świadomości. Już w latach 90. wspaniała historyczka literatury, prof. Maria Janion pisała o zmierzchu romantycznego paradygmatu.

Dziękuję bardzo. I pan poseł Grzegorz Rusiecki, Koalicja Obywatelska, zada ostatnie pytanie w tej serii. Wysoka Izbo! Dla mieszkańców Wielkopolski z całą pewnością bliższą epoką byłby pozytywizm i idea pracy organicznej, co wynika z pewnego pragmatycznego podejścia do życia, do pracy. Natomiast nie ulega żadnej wątpliwości, że także romantyzm odgrywa ogromną rolę w życiu każdego Polaka, w tym również Wielkopolanina. Nie można sobie wyobrazić życia bez muzyki i poezji, bez kultury, bez sztuki, w związku z tym przypomnienie takich osób jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid, Jan Matejko, Stanisław Moniuszko czy wielu, wielu innych jest niezwykle istotne, ważne i może wpłynąć na nasze ubogacenie wewnętrzne.

Dziękuję bardzo, panie pośle. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Bardzo bym chciał, żeby kolejny rok stał się Rokiem Polskiego Romantyzmu, żebyśmy pamiętali o tym, jak wyglądało wówczas nasze społeczeństwo. Wszyscy byli migrantami. Wyjeżdżali z różnych powodów: politycznych, ekonomicznych. Jedni byliby wygnani z porozbiorowej ojczyzny, inni szukali lepszego miejsca do życia. Trafili do różnych miejsc na świecie: do Francji, do Włoch, także do Stanów Zjednoczonych czy do Imperium Osmańskiego.

Teraz mamy szansę się odwdzięczyć. Dlatego pamiętajmy o tym wszystkim również w trakcie Roku Polskiego Romantyzmu. Szanowni państwo, na koniec poprosiłabym o głos sprawozdawcę komisji panią poseł Joannę Lichocką. Pani poseł, dopuszczam, ale bardzo proszę o krótką wypowiedź, bo mamy 45 minut opóźnienia. Pani Marszałek! Mnie się wydaje, że ta trybuna sejmowa zniesie wszystko, każde głupstwo. Chciałabym poprosić zwłaszcza posłów z tylnych ław, którzy wypowiadali różne głupstwa, żeby poczytali troszeczkę o tej epoce.

Ich praca jest podstawą do tekstu tej uchwały. Odniosę się także do zarzutów o rzekomym upolitycznianiu tej uchwały.

Proszę pani. Pani poseł, no naprawdę.

Spróbujcie nie zepsuć chociaż tego.

Bardzo proszę. Chciałam tylko powiedzieć, pani poseł, że była pani posłem sprawozdawcą. Wszyscy uważali, że to jest uchwała, która powinna być. Wszyscy akceptowali to, tylko pokazywali różne aspekty, co należy podkreślić, kiedy będziemy mówili i przygotowywali. A jedyne słowa, które padły o upolitycznieniu tej uchwały, padły z państwa strony. Zamykam dyskusję. Do głosowania nad projektem uchwały przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 19. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskich projektach uchwał o solidarności w sprawie ochrony polskich granic oraz w sprawie politycznego oraz humanitarnego kryzysu na granicy polsko-białoruskiej (druki nr 1758, 1759 i 1774) Uprzejmie proszę pana posła Jarosława Zielińskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Bardzo proszę, panie pośle. Wysoki Sejmie! Wczoraj Komisja Kultury i Środków Przekazu - posiedzenie komisji zakończyło się późno w nocy - rozpatrzyła projekt uchwały o solidarności w sprawie ochrony polskich granic, druk nr 1758, oraz poselski projekt uchwały w sprawie politycznego oraz humanitarnego kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, druk nr 1759.

Po przyjęciu tego rozstrzygnięcia niestety - co chcę powiedzieć z ubolewaniem - posłowie opozycji z klubów Koalicja Obywatelska i Lewica, opuścili salę posiedzenia komisji i nie brali udziału w dalszych obradach. Pozostali posłowie pracowali nad dokumentem i zgłoszono szereg poprawek i propozycji nowego brzmienia niektórych fragmentów projektu uchwały.

Reżim Aleksandra Łukaszenki zaatakował Polskę wykorzystując sprowadzone przez siebie tysiące migrantów do szturmu na granice Rzeczypospolitej Polskiej. Od wielu lat nasze państwo nie stało przed tak dużym zagrożeniem swego bezpieczeństwa i integralności granic. W chwili próby Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża w tej sprawie solidarność z polskim rządem wraz ze wszystkimi instytucjami państwa polskiego i osobami zaangażowanymi w obronę Polski i Polaków. Pokolenia naszych przodków walczyły o wolną i niepodległą Polskę. Pamiętając o ich poświęceniu dziś naszym obowiązkiem jest stanąć ramię w ramię z funkcjonariuszami Straży Granicznej i Policji, żołnierzami Wojska Polskiego, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej, i przedstawicielami innych służb dumnie noszącymi polski mundur i strzegącymi granic państwa oraz suwerenności naszej Ojczyzny. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża również wdzięczność lokalnej społeczności i wszystkim, którzy udzielają wsparcia naszym służbom na polskiej granicy oraz niosą pomoc humanitarną ofiarom kryzysu, za który pełną odpowiedzialność ponosi rząd Białorusi. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stanowczo potępia akcje dezinformacyjne i inne działania prowadzące do destabilizacji Polski.

Podstawowym zadaniem spoczywającym na wszystkich obywatelach Rzeczypospolitej, a w szczególności na reprezentantach polskiego narodu - niezależnie od poglądów politycznych - jest wspieranie instytucji państwa i jego służb. Rzeczpospolita Polska jest państwem silnym siłą swoich instytucji i swoich obywateli.

O tę solidarność Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się dziś do wszystkich Polaków” Jako poseł reprezentujący grupę posłów, którzy zgłosili ten projekt uchwały, oraz sprawozdawca komisji zwracam się do Wysokiego Sejmu o jak najszersze poparcie tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo, panie pośle. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Otwieram dyskusję. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość głos zabierze pan poseł Jarosław Zieliński. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Chciałbym, teraz występując w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, powiedzieć, że naszym zdaniem to wielka szkoda, że w polskim Sejmie, nawet w sytuacji tak poważnego zagrożenia bezpieczeństwa naszego państwa, ataku na polską granicę, nie ma solidarności ani zgody, tak bardzo pożądanych dla wzmocnienia naszej siły i odporności na podejmowane przez reżim białoruski, wspierany przez odradzający się imperializm rosyjski, próby siłowego forsowania granicy Rzeczypospolitej, w sytuacji podejmowanych prób dezintegracji polskiej granicy i polskiego terytorium.

One są odnotowywane z radością w Mińsku i na Kremlu, ale na pewno nie służą dobrze Polsce. Szanowni Państwo! Formułowane przez posłów Prawa i Sprawiedliwości apele o to, aby opozycja zaczęła myśleć wreszcie po polsku, nie przyniosły podczas tych posiedzeń żadnego rezultatu. Zamiast pracować. Szanowni Państwo! Można i pewnie trzeba mówić dużo ostrzej, ale oszczędzę państwu tego.

Kończąc to wystąpienie, chciałbym zgłosić wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały o solidarności w sprawie ochrony polskich granic, druki sejmowe nr 1758, 1759 i 1774. W imieniu Koalicji Obywatelskiej głos zabierze pan poseł Rafał Grupiński.

Bardzo proszę, panie pośle. Wysoki Sejmie!

Dlatego przedstawię naszą skróconą nieco ze względu na czas propozycję uchwały w sprawie politycznego i humanitarnego kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Unia Europejska w odpowiedzi na sfałszowanie wyborów, brutalne stłumienie pokojowych demonstracji, uwięzienie i prześladowanie tysięcy Białorusinów - nałożyła sankcje na reżim Aleksandra Łukaszenki. W odwecie Łukaszenka postanowił wywołać kryzys na granicy z Unią Europejską, w tym jej polskim odcinku, próbując zarazem naruszyć naszą suwerenność. W sposób szczególnie cyniczny i wyrachowany użył w tym celu ludzi wielu narodowości, uciekających przed prześladowaniami bądź brakiem perspektyw życiowych. Tysiące oszukanych przez reżim Łukaszenki ludzi koczuje po stronie białoruskiej w warunkach zagrażających ich życiu i zdrowiu. Blokując migrantom i uchodźcom możliwość powrotu do kraju, z którego przybyli, Aleksander Łukaszenka doprowadził do kryzysu humanitarnego, za który ponosi pełną odpowiedzialność. Sejm wyraża solidarność z funkcjonariuszami Straży Granicznej, Policji oraz żołnierzami Wojska Polskiego ochraniającymi granice Polski i Unii, którzy pełniąc odpowiedzialną służbę, winni jednocześnie respektować prawa człowieka i w swoich działaniach kierować się humanitaryzmem i zasadami konwencji do spraw statusu uchodźców. Sejm wyraża również solidarność z oddolnymi inicjatywami niesienia pomocy humanitarnej ofiarom działań reżimu Łukaszenki przez lokalnych mieszkańców oraz organizacje społeczne. Jednocześnie Sejm wzywa rząd do: umożliwienia niezależnym mediom relacjonowania wydarzeń na granicy w sposób bezpośredni i nieskrępowany, zapewnienia pomocy humanitarnej, w tym medycznej, wszystkim tym migrantom, a zwłaszcza kobietom i dzieciom, których zatrzymano na terytorium Polski, którzy takiej pomocy potrzebują, pilnego przedstawienia Komisji Europejskiej pakietu konkretnych propozycji zaostrzających sankcje wobec reżimu Łukaszenki. Ponadto Sejm Rzeczypospolitej uważa za wskazane podjęcie przez rząd oraz prezydenta RP stałej i efektywnej współpracy z odpowiednimi organami Unii Europejskiej odpowiedzialnymi za ochronę granic i migracje. Sejm Rzeczypospolitej wyraża przekonanie, że działając wspólnie i solidarnie z członkami Unii Europejskiej oraz NATO, kryzys wywołany przez Łukaszenkę zostanie opanowany i zażegnany.

Wydaje wam się, że jak tysiąc razy użyjecie słów: naród, Polska, patriotyzm, to patriotami staniecie się z automatu. Otóż nie. Bo nie słowa, a czyny świadczą o patriotyzmie. Pan poseł Maciej Konieczny w imieniu klubu Lewica. Bardzo proszę, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Na wczorajszym posiedzeniu komisji procedowane były dwie propozycje uchwał o granicy, o kryzysie. Jedna autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, druga Platformy Obywatelskiej. Niestety nie znalazła się wśród nich propozycja zgłoszona przez Lewicę, a szkoda. Do dalszego procedowania została wybrana propozycja PiS-u, w praktyce o bezwarunkowym poparciu dla rządu - tym bardziej szkoda. Skorzystam więc z okazji i przywołam to, co w naszej propozycji było najważniejsze. Dzięki temu być może łatwiej będzie zrozumieć, dlaczego nie możemy poprzeć tego, co proponuje rząd. Uchwała Sejmu powinna przede wszystkim jasno określać, kto w tej sytuacji jest agresorem, a kto ofiarą. Musi być jasne, że za kryzys humanitarny i próbę destabilizacji naszej części Europy odpowiada białoruski dyktator Aleksander Łukaszenka. Musi być jasne, że uchodźcy, imigranci cynicznie oszukani i brutalnie wykorzystani przez Białoruś są tutaj stroną pokrzywdzoną. Nie może być naszej zgody na stawianie znaku równości pomiędzy białoruską dyktaturą a demokratyczną Polską i Europą, dokładnie tak samo, jak nie może być naszej zgody na straszenie Polaków uchodźcami i kreowanie sztucznego zagrożenia z ich strony. W tej drugiej kwestii proponowana przez Prawo i Sprawiedliwość uchwała niestety zawodzi. Podobnie zresztą jak cała polityka obozu rządzącego, nastawiona na podsycanie lęku Polaków i straszenie uchodźcami. Dlatego będziemy głosować przeciw. Nie można mówić o kryzysie na polsko-białoruskiej granicy, nie wspominając o dramatycznej sytuacji humanitarnej ludzi. Nie można pomijać zasług mieszkańców Podlasia, personelu medycznego, aktywistów i aktywistek niosących pomoc potrzebującym. Im po prostu trzeba podziękować. Szacunek i uznanie dla wojskowych, policjantów, Straży Granicznej służących Polsce w tej trudnej sytuacji są ważne. Ważne, aby ten szacunek nie był czczym gadaniem, ale realnym wsparciem i zapewnieniem godnych warunków pracy. Szacunek to dobry sprzęt, który pochodzi od państwa, a nie z publicznych zbiórek. To naprawdę jest żenujące, że po paru tygodniach trwania kryzysu państwo polskie nie jest wstanie wyposażyć swoich ludzi w podstawowy sprzęt i organizuje publiczne zbiórki. Szacunek to wsparcie psychologiczne dla funkcjonariuszy mierzących się z ekstremalnie trudnymi sytuacjami. Szacunek w końcu to niezmuszanie ludzi do wykonywania nieludzkich i sprzecznych z prawem rozkazów. Oklaski nie zastąpią realnego wsparcia. Jeszcze bardziej razi wykorzystywanie służb mundurowych do partyjnych gierek. Rządzącym chodzi o to, żeby móc powiedzieć: albo deklarujecie bezwarunkowe poparcie dla rządu, albo nie szanujcie mundurowych. To naprawdę nie jest ładne zagranie w tej sytuacji. Nie godzi się sięgać po takie małe szantaże i manipulacje w świetle poważnego zagrożenia, naprawdę. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej powinna przede wszystkim jasno pokazywać, że granica między Polską a Białorusią to granica między demokracją i troską o drugiego człowieka a brutalną dyktaturą i pogardą dla bliźniego. Obawiam się tylko, że sama uchwała może tutaj nie wystarczyć. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości w tej kwestii, rząd musi w końcu dopuścić media, lekarzy (Dzwonek) i organizacje pomocy humanitarnej do granicy, otoczyć opieką wszystkie osoby, które znalazły się na terytorium naszego kraju, przestać obchodzić konstytucję i ograniczać prawa Polek i Polaków za pomocą ustawowych protez stanu wyjątkowego. Bardzo proszę o zaprezentowanie stanowiska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Solidarność i odpowiedzialność. Te słowa powinny dzisiaj nam przyświecać niezależnie od barw politycznych, bo chodzi o rzecz najważniejszą. Chodzi o bezpieczeństwo naszego kraju i naszych obywateli. Granica nie ma barw politycznych. Granica jest biało-czerwona, jak powiedział z tej mównicy prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Koalicja Polska i Polskie Stronnictwo Ludowe od początku tego konfliktu, jaki ma miejsce na polskiej granicy, nawołują do współpracy i współdziałania. Nie byliśmy przeciwni rozwiązaniom proponowanym przez partię rządzącą. Nie przeszkadzaliśmy przy wprowadzaniu stanu wyjątkowego, ale apelowaliśmy o dopuszczenie naszych dziennikarzy na granicę, bo media na granicy są po to, abyśmy nie byli pozbawieni informacji, abyśmy mogli wygrać wojnę z dezinformacją białoruską. W tej wojnie mamy szansę zwyciężyć, jeżeli będziemy mieli rzetelną informację od naszych dziennikarzy. Głosowaliśmy za ustawą w obronie polskiej granicy, proponując oczywiście nowe rozwiązania telemetryczne i montaż nowoczesnych urządzeń. Bo racja stanu i dobro państwa są dla nas najważniejsze, bo gdzie chodzi o interes Polski, tam kończy się polityka i należy współpracować. Ale tego współdziałania i chęci współpracy nie widać ze strony rządu, nie widać ze strony partii rządzącej. Dlaczego nie zwołano Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Dlaczego nie chcecie państwo podzielić się wiedzą, usiąść do stołu i wspólnie szukać rozwiązań? Z naszej strony proponujemy świetnych ekspertów: doświadczonego ministra posła Marka Biernackiego, doświadczonego dyplomatę Władysława Teofila Bartoszewskiego. Dlaczego nie chcecie skorzystać z ich wiedzy i doświadczenia? Jak najszerzej należy umiędzynarodowić ten problem, do czego nawołujemy od początku. Wczoraj również jako posłowie odpowiedzialni za bezpieczeństwo naszego kraju i otwarci na współpracę wspólnie pochyliliśmy się nad treścią tej uchwały. Niestety z państwa strony kompromis jest wciąż rzeczą bardzo trudną. Pamiętajmy, że ten kryzys jest kryzysem międzynarodowym i skorzystajmy z pomocy Unii Europejskiej, aby go jak najszybciej zlikwidować. Oczekujemy większej aktywności rządu na scenie dyplomatycznej i politycznej, bo to jest zadanie i odpowiedzialność polskiego rządu. Na granicy Polski z Białorusią, która - podkreślam - jest też granicą Unii Europejskiej, niestrudzenie od kilku miesięcy pracują i strzegą jej (Dzwonek) nasi żołnierze, żołnierze WOT-u, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej i jak zwykle. Pani marszałek, proszę jeszcze o minutkę, dobrze? gotowi do niesienia pomocy druhowie z ochotniczych straży pożarnych, za co im z całego serca dziękujemy. Na granicy od wielu miesięcy pracują. nasi obywatele, którym los drugiego człowieka nie jest obojętny, którzy osobiście codziennie, każdego dnia niosą pomoc tym ludziom. Ja tylko jeszcze chciałam zgłosić wniosek. Jako Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe będziemy głosowali za tą uchwałą.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! PiS to są totaliści, a wtórują im w tym Lewica oraz Koalicja Obywatelska. Trzeba pamiętać o tym, że właśnie wszelkie aktywności godzące w wolność słowa to jest wasza wspólna koalicja.

Jakże antypaństwowym ojkofobem trzeba być, żeby w sytuacji takiego kryzysu inspirowanego z zewnątrz, gdzie państwo polskie jest właśnie ofiarą agresji, a instytucje państwa polskiego są poddawane destabilizacji, bojkotować pracę polskich instytucji, funkcjonariuszy czy nawet polskiego parlamentu. My nie jesteśmy anarchistami czy mentalnymi poddanymi lewackich aktywistów, którzy dzisiaj na granicy też robią swoje teatrzyki. Nie będziemy krzyczeć czy epatować obrazkami. Nie będziemy zgadzać się właśnie na anarchię. Stąd współpracowaliśmy w tej konkretnej kwestii, bo najważniejszy jest dla nas interes państwa polskiego. Pamiętajcie, szanowni państwo, że właśnie tam, na Wschodzie, bardzo się cieszą, kiedy my w polskim Sejmie, tutaj, w tym budynku jesteśmy podzieleni, kiedy ulegamy demagogii i kiedy ulegamy szantażowi emocjonalnemu.

Konfederacja wzięła też udział we wczorajszych pracach komisyjnych i wypracowała jakiś model, jakąś propozycję, która dzisiaj została ogłoszona, bo dla nas są rzeczy ważniejsze niż interesiki partyjne, a jest to interes narodowy i bezpieczeństwo Polaków. W tej jednej kwestii możemy mówić jednym głosem, możemy solidarnie wspierać państwo polskie, nie tylko funkcjonariuszy, ale wszystkie instytucje państwa polskiego, bo Straż Graniczna, wojsko, właśnie Policja czy strażacy działają dzisiaj na granicy, działają tam w imię naszego bezpieczeństwa i polski Sejm musi się z nimi solidaryzować. Polski Sejm musi też jasno powiedzieć, kto jest odpowiedzialny za kryzys humanitarny, który jest tam, na granicy, a jest to państwo białoruskie. Ta uchwała, o której dzisiaj mówimy, to jest tylko gest. Naturalnie za gestem muszą iść konkretne czyny, czyli m.in. mur, którego dalej nie mamy, a także sankcje nałożone na Białoruś w zakresie tranzytu. Pamiętajmy, że za każdym takim gestem jest też konkretna informacja dla świata, że państwo polskie jest zdeterminowane, by chronić swoich obywateli. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Poprzednie posiedzenie Sejmu poświęciliśmy wyważonej dyskusji o sytuacji na granicy, wyjątkowo. Chcieliśmy zakończyć tę dyskusję wspólną uchwałą Sejmu wyrażającą solidarność z mundurowymi strzegącymi dziś integralności Rzeczypospolitej, nie zapominając o podziękowaniach dla tych, którzy niosą bezinteresowną pomoc osobom znajdującym się dziś w kryzysie humanitarnym. Poprawkę w tym duchu zanieśliśmy wczoraj do komisji kultury, szukając najmniejszego wspólnego mianownika, pod którym bylibyśmy się w stanie dziś podpisać bez względu na podziały polityczne, bo uważamy, że dziś, w godzinie próby taki wspólny głos jest bardzo potrzebny, by pokazać wsparcie strażnikom, żołnierzom, policjantom, mieszkańcom, wolontariuszom, medykom, wszystkim, którzy dziś bezpośrednio angażują się w obronę polskich granic i niosą pomoc bliźniemu. Choć z uznaniem znajdujemy dodanie do uchwały akapitu doceniającego niosących pomoc humanitarną, to niestety nie możemy zgodzić się z zapisem, który wśród bohaterów polskiej granicy w jednym szeregu umieszcza polski rząd. Rząd ma już swoje media i dość chwały na konferencjach i mógłby taktownie wycofać swoją obecność z treści tej uchwały, tak byśmy mogli podjąć jako Sejm wspólne stanowisko. Koło Parlamentarne Polska 2050 z prawdziwym żalem nie poprze uchwały w tym kształcie, jednak mamy nadzieję, że w przyszłości nie zmarnujemy podobnej szansy, a co do działań, które robimy na granicy, już teraz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wolontariuszom i wszystkim aktywistom Ruchu Polska 2050, który w całej Polsce prowadzi w tej chwili zbiórki, kupuje pakiety ratunkowe. Tych pakietów na granicę dowieźliśmy 300. Każdy z nich zawiera konieczne do ratowania życia i zdrowia akcesoria. Dziękuję też wszystkim organizacjom, wszystkim wolontariuszom i wszystkim mundurowym, którzy w tej chwili strzegą naszych granic i którzy wykazują ludzkie odruchy. Przechodzimy do pytań. Wyznaczam czas na zadanie pytania - 1 minuta. Bardzo proszę. Jak zawsze, panie pośle. Bardzo dziękuję. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałem zadać pytanie panu posłowi, który jest przedstawicielem wysokiej komisji. Panie pośle, to jednak jest zaskakujące, że państwo chcą solidaryzować się z rządem, który nie potrafi zapewnić żołnierzom, funkcjonariuszom odpowiedniego wyekwipowania na granicy. Docierają do nas informacje, że wśród mieszkańców są organizowane zbiórki różnego rodzaju wyposażenia, zbiórki żywności. Oczywiście dobrze, że mieszkańcy wspomagają funkcjonariuszy i żołnierzy, ale takie rzeczy powinien zapewnić rząd. Tymczasem pan chce się solidaryzować, państwo, komisja chce się solidaryzować z rządem, który wysłał żołnierzy na granicę i ich tam po prostu zostawił. Podobnie, jeżeli chodzi o kwestie posiłków.

Szanowni państwo, mamy duże opóźnienie i 20 osób zapisanych do pytań, w związku z czym bardzo proszę o trzymanie się czasu. Wysoka Izbo! Na granicy z Białorusią mamy konflikt o charakterze nie tylko europejskim, ale także światowym. W związku z tym jest takie pytanie: Dlaczego do teraz rząd nie załatwił żadnego realnego wsparcia ze strony krajów Unii Europejskiej? Dlaczego rząd boi się wpuszczenia dziennikarzy do strefy przygranicznej? Dlaczego rząd chowa głowę przed opinią publiczną poprzez brak wpuszczenia dziennikarzy? Czy pan premier Morawiecki poddał się prezydentowi Łukaszence w wojnie propagandowej, który nie bał się wpuszczenia CNN i innych dziennikarzy zagranicznych? Dlaczego w końcu pan prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej nie zechce porozmawiać ze wszystkimi w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Pan poseł Franciszek Sterczewski, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Jeżeli mamy do czynienia z tak poważnym kryzysem, to dlaczego nie zwołaliśmy Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Dlaczego przy każdej z debat na ten temat, na temat stanu wyjątkowego, na temat muru itd., nie było na tej sali pana prezydenta Andrzeja Dudy? Dlaczego w tym samym czasie pan prezydent może pójść na mecz Polska - Węgry? Czy to świadczy o tym, że wam zależy na tym, żeby zakończyć ten kryzys? Nie sądzę. W interesie tego państwa jest bronić zarówno granic, jak i człowieczeństwa, a zatem te rzeczy się zupełnie nie wykluczają. Powinniśmy robić wszyscy, od prawa do lewa, wszystko, żeby ten kryzys humanitarny zakończyć jak najszybciej. Miarą patriotyzmu nie są czcze słowa, które słyszymy w treści tej uchwały, ale czyny. Jeżeli jesteście patriotami, to powinniście wezwać Frontex do pomocy, organizacje pomocowe, dopuścić dziennikarzy do granicy. Pani poseł Małgorzata Pępek, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Za waszych rządów już dawno straciliśmy podmiotowość w polityce międzynarodowej, a kryzys na granicy polsko-białoruskiej, który jest dyplomatyczną i wizerunkową katastrofą naszego kraju, tylko to potwierdza. Doprowadziliście do tego, że o Polsce rozmawia się bez udziału Polski. Tylko dzięki Unii tureckie linie lotnicze już nie będą przyjmować na pokłady samolotów do Mińska obywateli Iraku, Syrii i Jemenu. Trzeba było rozmowy szefowej Komisji Europejskiej i prezydenta USA, żeby zapadła decyzja o sankcjach przeciwko Białorusi, bo wy nie umieliście nawet zacząć debaty na ten temat.

Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Metoda push-back-ów, czyli metoda wypychania uchodźców z polskiego terytorium z powrotem za granicę, jest metodą nieskuteczną, niehumanitarną i niezgodną z międzynarodowym prawem. To jest zgoda na znęcanie się nad ludźmi i zgoda na systemową śmierć. Niestety, ci ludzie po kilku razach, po kilkunastu razach mają coraz mniejsze szanse na przeżycie. Winą za to obarczam rząd i obarczam również parlamentarzystów, którzy za tą ustawą głosowali. Moje pytanie jest takie: Kiedy wycofacie się z tej haniebnej ustawy? Musimy zatrzymać to szaleństwo. Pytanie jest również takie: Ile tych push-back-ów było? Pan poseł Krystian Kamiński, koło Konfederacja.

Wysoka Izbo! To, że część osób na tej sali, która uważa, że bezpieczna granica to bezpieczna Polska, poprze dzisiaj ten projekt uchwały, jest dobrym znakiem. Ale tak naprawdę ludzie, którzy są na granicy, wojsko, Straż Graniczna, Policja potrzebują widocznego znaku, czyli muru, płotu, zapory czy jakkolwiek byśmy to nazwali. To jest zdecydowanie za późno. Oni potrzebują naszego dobrego słowa, ale przede wszystkim muszą czuć się bezpiecznie. Bez szybszego wybudowania tego płotu, tej zapory, to się nie wydarzy. Dlatego apeluję, żeby przyspieszyć to i żebyśmy jak najszybciej zapewnili bezpieczeństwo naszym służbom granicznym. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Z tego miejsca chciałbym po raz kolejny, pomimo że w uchwale dziękujemy, podziękować ludności, mieszkańcom tamtych terenów za to, co robią każdego dnia, jak wspierają tych wszystkich, którzy mimo wszystko przedostają się przez granicę. Jednocześnie mam dwa konkretne apele do rządzących. Niestety tamtejsi przedsiębiorcy cały czas mówią o tym, że wsparcia, rekompensat, które były obiecane. Jakoś trudno przychodzą te rekompensaty, dlatego proszę o przyspieszenie tego tematu, ponieważ oni realnie każdego dnia tracą i tracą. Druga sprawa.

Pani poseł Małgorzata Tracz, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W czasach, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo narodowe, obowiązkiem rządzących jest szukanie i budowanie jedności narodowej. To oznacza też szukanie poparcia opozycji i jej wyborców. Takie działania wymagają wykonywania przynajmniej symbolicznych gestów, a wy takiego gestu nie wykonaliście. Postanowiliście stosować dobrze wszystkim znany sejmowy walec, by przeforsować wasz projekt, a odrzucić nasz projekt uchwały. Co wam się nie podoba w naszym projekcie uchwały? Nie podoba wam się potępianie Aleksandra Łukaszenki za wywołanie kryzysu politycznego i humanitarnego oraz wykorzystywanie zdesperowanych ludzi? Nie podoba wam się stwierdzenie, że polska i światowa opinia publiczna zasługują na relację medialną płynącą nie tylko ze strony białoruskiej? Nie podoba wam się podkreślenie roli wsparcia i solidarności Unii Europejskiej i NATO w rozwiązaniu tego kryzysu?

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

W tej dyskusji pojawiło się wiele słów, padły słowa o zgodzie, o porozumieniu, o poparciu dla tej uchwały. A potem jak przyszło, co do czego, i trzeba było głosować nad wnioskiem o powołanie podkomisji, która miałaby wypracować wspólny tekst uchwały, to okazało się, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości byli przeciw. Proszę państwa, czyny, nie słowa. Jeżeli przychodzi się i mówi o tym, że ta uchwała powinna zostać poparta przez wszystkich, że wszyscy powinniśmy się na nią zgodzić, to oznacza to też tyle, że powinna zostać wspólnie wypracowana przez przedstawicieli wszystkich klubów.

Tego niestety rząd PiS-u nie potrafił zrobić. Mianowicie w dziele Poliajnosa „Podstępy wojenne” jest opisana setka bitew starożytnych i różnych podstępów wojennych, ale jest jeden charakterystyczny fragment o Filipie Macedońskim. Filip osiągnął nie mniej dzięki rozmowom niż za pomocą oręża i, na Zeusa, bardziej się chlubił tym, co zyskał za sprawą wymowy, niż tym, co zdobył zbrojnie. To była podstawa potęgi, na której potem budował swoje imperium Aleksander Macedoński.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Pan poseł Andrzej Szewiński, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dlaczego przedstawiciele formacji rządzącej w Sejmie mówią o potrzebie współpracy w obliczu kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, a nie podejmują współpracy z opozycją?

A jakie są efekty braku skutecznej polskiej dyplomacji?

Pani Marszałkini. Wysoka Izbo! Na granicy polsko-białoruskiej jest ok. 5 tys. uchodźców.

Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Pan przewodniczący Rafał Grupiński powiedział, że czyny, a nie słowa decydują, kto dobrze życzy Polsce. w istocie. Byliście, szanowni państwo, przeciwko budowie zapory, byliście przeciwko budowie muru, przeciwko ustawie o granicy. Wcześniej byliście przeciwko Wojskom Obrony Terytorialnej, a tym samym - przeciwko wzmocnieniu Wojska Polskiego.

Dziękuję bardzo. Pan poseł Grzegorz Rusiecki, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Rzeczywiście ta solidarność jest niezwykle istotna, ważna.

Relacje polsko-białoruskie są niezwykle istotne. Gdyby nie to, że sfałszowano wybory na Białorusi, dzisiaj pewnie mielibyśmy zupełnie inną sytuację, ale to tym bardziej zmusza nas do tego, aby wspólnie postarać się rozwiązać te problemy. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Tak jak oklaskami nie da się uleczyć ochrony zdrowia, tak hashtagiem: murem za mundurem nie wzmocni się polskich funkcjonariuszy służących przy polskiej granicy. PR-owskie zagrywki nie zastąpią godnego traktowania, sprzętu, opieki psychologicznej, a przede wszystkim wolności od przymusu wykonywania nieludzkich rozkazów, takich jak rozkaz nielegalnej wywózki dzieci do lasu. Dziś polski mundur potrzebuje obrony, ale obrony przed splamieniem rozkazami władzy, po których mundurowym trudno będzie spojrzeć w lustro. Pani poseł Daria Gosek-Popiołek, klub Lewica. Wysoka Izbo! Chciałabym przytoczyć kilka zdań napisanych przez mieszkańców Białowieży, którzy założyli Białowieską Akcję Humanitarną: Jesteśmy ludźmi o różnych poglądach, ale łączy nas głębokie przekonanie, że udzielanie pomocy humanitarnej ludziom w skrajnie trudnej sytuacji życiowej jest naszym prawem i obowiązkiem obywatelskim. Mieszkając w strefie stanu wyjątkowego, nie możemy liczyć na pomoc z zewnątrz. Nie mamy wsparcia medycznego ani medialnego. Zostaliśmy zostawieni sami z sytuacją przerastającą wszelkie nasze wyobrażenia. Mimo wszystko chcemy nieść pomoc potrzebującym. Jesteśmy otwarci na współpracę z władzami samorządowymi, służbami mundurowymi, zakładami pracy, organizacjami i osobami prywatnymi. Udzielenie pomocy humanitarnej rozumianej jako zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych w żaden sposób nie narusza zasad obowiązujących w strefie stanu wyjątkowego.

Proszę państwa, nie jest tajemnicą, że wiele i wielu z nas ocenia negatywnie politykę rządu wobec kryzysu na granicy. Podtykanie nam uchwały Sejmu, która wyraża bezwarunkową solidarność z tą polityką, siłowe jej narzucanie i przepychanie w komisji i nazywanie tego współpracą uważam za wyjątkową hipokryzję.

Zamiast tego na tym samym oddechu, na którym wzywacie nas do tej współpracy, obrażacie już nawet nie tylko nas, ale przede wszystkim tych, którzy na granicy niosą pomoc. Nie tylko omijacie ich w tym projekcie uchwały, nie tylko omijacie ich w waszej komunikacji, ale też obrażacie ich wprost, powielając kłamstwa. To jest skandaliczne. Bardzo proszę, panie pośle. Wysoka Izbo! To naprawdę niebywałe, że część opozycji tak mocno działa przeciwko interesom Polski. Chciałbym zapytać, dlaczego państwo głosowaliście przeciwko wprowadzeniu stanu wyjątkowego w Polsce, dlaczego głosowaliście przeciwko przedłużeniu tego stanu. Dlaczego głosowaliście przeciwko ustawie o budowie muru na granicy? Dlaczego wczoraj zgłosiliście wniosek o odrzucenie ustawy o obronie granicy państwowej? Dlaczego - jeszcze raz pytam - działacie przeciwko interesom Polski? Dzisiaj tak ważny jest szacunek dla polskiego munduru. Wczoraj 12 funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej zostało rannych, i jeden żołnierz Wojska Polskiego. Panie pośle, miał pan swój czas na mównicy. Bardzo proszę. Panie pośle. Wysoka Izbo! Założeniem tej uchwały miało być wsparcie nas wszystkich, parlamentarzystów, dla obrony polskich granic, dla ludzi, którzy tych granic bronią. A państwo chcieli zrobić z tego laurkę na cześć rządu. Rząd, który musi chwytać się takich działań, rząd, który za wszystkie swoje niepowodzenia oskarża opozycję, jest rządem słabym. Bo to wy macie odpowiedzialność i wy macie narzędzia do tego, żeby bronić polskich granic. A doprowadzacie do tego, że nie mówicie prawdy, że kłamstwo funkcjonuje w domenie publicznej. Wczoraj na posiedzeniu komisji słyszeliśmy kłamstwa, brak szacunku dla nas, największe obelgi, jakie mogli usłyszeć posłowie. Odbieraliście nam prawo do patriotyzmu, godności i do podejmowania decyzji. Jeżeli tak ma wyglądać współpraca, jeżeli tak mamy razem działać, to będziecie bardzo osamotnieni.

Wysoka Izbo!

Ale na granicy jest również mocny kryzys humanitarny. Myślę, że powinniśmy być wdzięczni i służbom medycznym, i szczególnie wolontariuszom indywidualnym, zorganizowanym, również organizacjom pomocowym, także zorganizowanym, indywidualnym, ludziom wielkiego serca, licznym mieszkańcom terenów przygranicznych, którzy poświęcają własne pieniądze, czas i próbują właśnie w tym ujęciu humanitarnym pomagać nieszczęsnym ludziom na granicy.

Uprzejmie proszę pana posła o udzielenie odpowiedzi na postawione pytania. Szanowni Państwo! Projekt uchwały złożony przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość dotyczył - chciałbym to przypomnieć - wyrażenia solidarności w sprawie ochrony polskiej granicy.

Rzeczywiście się różnimy, i to bardzo, w ocenie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i jej źródeł. Można by dużo mówić, przywoływać wypowiedzi wielu z państwa.

Państwo w różnych wypowiedziach, może w mniej wyrazisty sposób, też to sugerujecie. Zapytał, czy brakuje nam ziemniaków, chleba, soli itd., żeby wszystkich tych nielegalnych imigrantów zaprosić do Polski. Pan poseł Mieszkowski świetnie to wyraził. Jeżeli uważacie, że trzeba do Polski wpuścić wszystkich tych, którzy w sposób brutalny, nielegalny forsują, za sprawą reżimu Aleksandra Łukaszenki, polskie granice, prowadzą do tego, że ranni zostają polscy funkcjonariusze, policjanci, żołnierze, funkcjonariusze Straży Granicznej, to gratuluję.

I bardzo wam przeszkadza, kiedy w jednej z fraz tej uchwały pojawia się również sformułowanie dotyczące polskiego rządu. Tak, właśnie polski rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj - nawet nie napisaliśmy, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale to jest oczywiste - chroni polskie granice.

Mówiliście wtedy, łącznie z waszą panią premier, że Polska przyjmie te wszystkie kwoty i nie powinna się przed tym bronić. Proszę państwa, jak daleko idące jest to nieporozumienie? Ja też do tego się odnosiłem, mówiąc, że tak, kompromis to jest wartość, ale to nie jest wartość ponad wszystko, to nie jest wartość za wszelką cenę. Bo jeżeli kompromis miałby polegać na tym, że odstępujemy od solidarności w Polsce w odniesieniu do ochrony, obrony polskiej granicy, że wpuszczamy imigrantów i narażamy się na wszystkie te problemy i procesy, które to ze sobą niesie, to po prostu tutaj nie może być kompromisu. My też chcielibyśmy, żeby byli, tylko widzieliście państwo, co się działo na początku tego kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Większość dziennikarzy jest odpowiedzialna, większość polityków też jest odpowiedzialna, ale widzieliśmy te zachowania, te spektakle na granicach. Widzimy, co się teraz dzieje pod naporem tych wielkich grup, które są wypychane przez reżim Łukaszenki i jego służby na polską granicę i do Polski. Na pewno nie zapewnią też tego bezpieczeństwa dziennikarze biegający po granicy przed funkcjonariuszami, przepytujący ich na każdym kroku, co robią. Nie wiem, czy to jest tak, że ma tutaj miejsce brak elementarnej wiedzy i realizmu, czy jest coś znacznie gorszego, czego nie chcę się domyślać, w tej waszej postawie. Tak i właśnie to rząd robi wraz ze służbami państwa polskiego. Ale jak się pojawia sformułowanie, że rząd polski w ramach tej solidarności też ma tę swoją rolę, to mówicie: nie, wymieniajcie instytucje, ale bez rządu. Proszę siebie słuchać po prostu, bo to jest coś dramatycznie fałszywego, co wy wyprawiacie w tej dyskusji.

My rozmawiamy o uchwale o solidarności, a wy szukacie wszystkich możliwych i niemożliwych argumentów, żeby właśnie tej solidarności nie było. To jest wasza postawa. Ta postawa, szanowni państwo, ma swoje odniesienia historyczne. Nie będę o tym mówił, bo będziecie zaraz tutaj robić wielki hałas, ale sami wiecie, jakie to są odniesienia, nie trzeba tego nawet przywoływać.

Szanowni Państwo! Teraz tak.

Zapytajcie mieszkańców, oni wam powiedzą.

Nie zyskacie go w ten sposób, to jest błędna droga. Można powiedzieć, że politycznie to jest wasza sprawa, to jest wasz problem, tak? Ale to jest polski problem. żeby obronić się przed zagrożeniem bezpieczeństwa zewnętrznego. Nie róbcie z nich, szanowni państwo, takich ludzi, nad którymi trzeba się pochylać z wielką troską, nad każdym z nich, bo oni przecież forsują siłowo i nielegalnie polskie granice. Na Białorusi się nie da. Chcieliśmy wysłać pomoc humanitarną, ale nie przyjęto, Białoruś jej nie przyjęła. Żeby pomóc w Polsce, trzeba ich wpuścić, czyli trzeba zaakceptować nielegalną masową migrację. To jest wasza filozofia, do tego nas namawiacie. Nie, nie pójdziemy tą drogą.

Przypomnę symboliczną sprawę. Dzisiaj wszystkie placówki Straży Granicznej są bardzo potrzebne i pełnią niezwykle istotne funkcje na granicy polsko-białoruskiej. Wy te placówki chcieliście likwidować. Placówka Straży Granicznej w Krynkach, jedna z placówek na granicy polsko-białoruskiej, miała być przez was zlikwidowana. Broniliśmy, sam broniłem, wtedy jako poseł opozycji, samorządowcy bronili tej placówki. My w ramach programu modernizacji, jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, zbudowaliśmy tam nowe obiekty, zbudowaliśmy wieże obserwacyjne. A gdybyście to zlikwidowali, nie byłoby tego. A chcieliście likwidować także. Bo przeszkodziliśmy wam w tym.

Szanowni Państwo!

Mają.

Myślę, że to jest wyraz wdzięczności mieszkańców tego terenu.

To jest wyraz wdzięczności.

To są bardzo szlachetnie akcje, bardzo cenne, bardzo potrzebne. Oni służą nam wszystkim, wszystkim Polakom. W pierwszej kolejności służą Polakom, którzy mieszkają najbliżej granicy, bo ich bezpieczeństwo jest najbardziej zagrożone. Proszę państwa, gdybyśmy was słuchali, nie byłoby stanu wyjątkowego, nie byłoby placówek Straży Granicznej, nie byłoby programu modernizacji służb mundurowych. Byłoby mniej funkcjonariuszy. Straż Graniczna nie miałaby broni długiej. My im ją przywróciliśmy. Można mówić dalej. Szanowni Państwo! Wasza polityka to było nieszczęście, a dzisiaj macie odwagę, macie czelność atakować rząd za to, co jest robione. Dzięki działaniom polskiego rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości, dzięki instytucjom państwowym, dzięki służbom mundurowym, dzięki wojsku Polska skutecznie chroni się przed tym zagrożeniem. Chronimy polskie granice.

Chcieliśmy dać wam szansę. Wystąpmy razem. Na pewno historycznie byłoby to dobrze ocenione.

W takich sprawach powinniśmy być razem.

Okazuje się, że ani jedno, ani drugie. Szkoda. Polacy was ocenią, historia was oceni.

Mam nadzieję, że dzisiaj przegłosujemy także ustawę o zmianie ustawy o ochronie granic.

Chcemy to uregulować, uporządkować i dopuścić dziennikarzy według reguł, które są zapisane w projekcie ustawy, zaprosić ich w te miejsca, żeby, mamy nadzieję, obiektywnie relacjonowali zdarzenia.

Dziękuję bardzo, panie pośle. W dyskusji zgłoszono poprawkę oraz wniosek o nieodsyłanie projektu ustawy do komisji w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 20. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawartego między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r. (druki nr 1706 i 1755) Uprzejmie proszę pana posła Michała Jacha o przedstawienie sprawozdania komisji. Bardzo proszę.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie połączonych Komisji: Obrony Narodowej oraz Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawartego między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r., druk nr 1706. Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu, skierowała w dniu 28 października 2021 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych do pierwszego czytania. Wysoka Izbo!

Jednym z takich elementów w zamierzeniu był Eurokorpus, który został utworzony przez francusko-niemiecką Radę ds. Obrony i Bezpieczeństwa w dniu 22 maja 1992 r. W kolejnych latach dołączyły do niego Belgia, Holandia i Luksemburg, a korpus osiągnął pełną gotowość operacyjną w 1995 r.

Na posiedzeniu ministrów obrony narodowej państw Trójkąta Weimarskiego w 2006 r. przez Polskę została przedstawiona inicjatywa uzyskania statusu państwa ramowego, tzn. pełnego członkostwa w Eurokorpusie. Inicjatywa ta uzyskała aprobatę ministrów obrony narodowej Niemiec i Francji i w 2008 r. rozpoczęto negocjacje z wszystkimi państwami ramowymi. W 2016 r. działania te zostały wstrzymane wobec niedookreślonych, niejasnych zadań Eurokorpusu w strukturach NATO, a minister obrony narodowej podjął decyzję o stopniowym wycofywaniu się z Eurokorpusu. Obecnie w sytuacji, gdy rola i cele Eurokorpusu w strukturach NATO rosną, jego znaczenie jest bardzo istotne jako korpusu szybkiego reagowania, strona polska powróciła do planów uzyskania statusu państwa ramowego. To bardzo ważne, że będziemy członkiem liczącego się nie tylko w strukturach NATO elementu decydującego o stabilności i bezpieczeństwie nie tylko naszego regionu. Polska skutecznie aspiruje do odgrywania istotnej roli we wszelkich strukturach bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Połączone Komisje: Obrony Narodowej oraz Spraw Zagranicznych po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2021 r. wnoszą, aby Wysoki Sejm uchwalić raczył projekt ustawy z druku nr 1706 bez poprawek. I jeszcze taka refleksja, proszę państwa. Komisja przyjęła tę opinię jednogłośnie. Proszę państwa, w sytuacji kiedy ostatnio tak wiele dzieje się w zakresie bezpieczeństwa, podejmujemy bardzo wiele decyzji, ta zgoda była dla mnie wielce istotna, bo, proszę państwa, liczę na to i apeluję, że w kolejnych przedsięwzięciach, które będziemy podejmować w zakresie bezpieczeństwa, w tym oczywiście w likwidacji największego problemu, największego zagrożenia, jakim jest sytuacja na wschodniej granicy, wreszcie dojdzie do wspólnego głosu całej tej Izby.

Proszę państwa, ci ludzie, którzy pełnią niezwykle ciężką służbę, o której w poprzednim wystąpieniu była mowa, apelują o to, żebyśmy w tej kwestii nie podgrzewali atmosfery, żebyśmy poparli naszych pograniczników, policjantów, strażaków i żołnierzy.

Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jednocześnie uprzedzam, że będę bardzo ściśle trzymać się wyznaczonego czasu na wystąpienia, ponieważ mamy godzinne już w tej chwili opóźnienie. W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość głos zabierze pan poseł Paweł Hreniak. Bardzo proszę. Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić opinię klubu Prawa i Sprawiedliwości odnośnie do projektu ustawy o ratyfikacji traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego dowództwa. Eurokorpus zgodnie z zamysłem ma wzmocnić zdolność Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej do prowadzenia operacji militarnych, w tym misji humanitarnych i ratowniczych, misji przywracania i utrzymania pokoju oraz możliwej realizacji zadań w ramach kolektywnej obrony NATO. Negocjacje z państwami ramowymi Eurokorpusu były prowadzone przez dłuższy czas i zostały wstrzymane przez stronę polską w roku 2016. Ta decyzja była wynikiem zapowiadanych zmian charakteru aktywności Eurokorpusu, polegających na skupieniu się na udziale w szkoleniowo-doradczych misjach reagowania kryzysowego Unii Europejskiej kosztem obrony w ramach NATO, czyli tej części, która jest dla nas częścią najistotniejszą i najbardziej przez nas pożądaną. Obecnie korpus przekierował się w dużo większym stopniu na Sojusz Północnoatlantycki. Dokonano zmian w jego funkcjonowaniu i zwiększono jego rolę w strukturze sił NATO, stąd też decyzja Polski o powrocie do działań, których celem jest pełne uczestnictwo w Eurokorpusie. Status pełnoprawnego członka Polski w Eurokorpusie zapewni nam wpływ na decydowanie o zadaniach, strukturze i rozwoju tej jednostki.

W obecnej sytuacji, po zmianach w Eurokorpusie Polska będzie mogła skutecznie oddziaływać na kierunki i zaangażowanie, licząc na to, że zwiększy się jego rola w polityce odstraszania i obrony wschodniej flanki NATO i Unii Europejskiej. W związku z płynącymi korzyściami wynikającymi z ratyfikacji traktatu Klub Prawa i Sprawiedliwości popiera przyjęcie projektu ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. W imieniu Koalicji Obywatelskiej głos zabierze pan poseł Andrzej Szewiński.

Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu wobec projektu ustawy ujętej w druku nr 1706 oraz w druku nr 1755, dotyczącej ratyfikacji traktatu w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Eurokorpusu. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Już w lutym 2008 r. premier Donald Tusk zaakceptował propozycję osiągnięcia przez Polskę statusu państwa ramowego Eurokorpusu i w konsekwencji rząd podjął działania dotyczące przystąpienia Polski do traktatu. Niestety w 2016 r. ówczesny minister obrony narodowej rządu Prawa i Sprawiedliwości podjął decyzję o nieprzystąpieniu Polski do Eurokorpusu. Patrząc na to z perspektywy czasu, była to zła decyzja. Po 2008 r. Federacja Rosyjska pośrednio była zaangażowana w konflikt w Gruzji, Osetii Południowej, konflikt w Górskim Karabachu, eskalację sytuacji kryzysowej w Bośni i Hercegowinie, Naddniestrzu czy też w konflikt na Ukrainie. Mając na uwadze radykalną zmianę środowiska bezpieczeństwa w Polsce, w krajach nadbałtyckich, na wschodniej flance NATO, dobrze, że obecny rząd powrócił do koncepcji z 2008 r. Tutaj patrzę na pana wiceministra Skurkiewicza. Ratyfikacja przedmiotowego traktatu spowoduje przystąpienie Polski do Eurokorpusu na prawach państwa ramowego. Status państwa ramowego umożliwi współdecydowanie w sprawie kierunków zaangażowania Eurokorpusu, również w ramach kolektywnej obrony NATO. Przedmiotowa ratyfikacja wpisuje się w podniesienie poziomu obronnego Unii Europejskiej, w tym wpłynie na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz wzmocnienie europejskiego wkładu w Sojuszu Północnoatlantyckim. Zwiększenie zaangażowania i odpowiedzialności Unii Europejskiej w obszarze obronności przyczynia się do wzmocnienia zdolności Eurokorpusu, który stanowi mocny komponent wspólnej polityki obronnej nie tylko państw europejskich, ale również państw Sojuszu, NATO. Jest jedną z odpowiedzi na wyzwania i kryzysy, takie jak działania by proxy, działania hybrydowe, jakie np. Federacja Rosyjska przez aktora zastępczego Białoruś może realizować (Dzwonek), testując solidarność państw Zachodu. Nie, mówiłam, że się będę trzymać tego. Bardzo proszę, panie pośle, pan poseł Andrzej Szejna. Przepraszam, mamy godzinne opóźnienie. Panie pośle, pan uniemożliwia w tej chwili dalsze prowadzenie obrad. Proszę wybaczyć. Zapraszam, panie pośle. Wysoka Izbo! Ratyfikacja traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego dowództwa z dnia 22 listopada 2004 r. ma duże znaczenie w rozpoczęciu również europejskiej debaty nad dalszą procedurą zacieśnienia więzi pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej i stronami Paktu Północnoatlantyckiego, w tym przypadku w obszarze bezpieczeństwa i sił zbrojnych. Bardzo dobrze, panie ministrze, naprawiliście błąd ministra Macierewicza, który chciał się z tego w ogóle wycofać, a koncepcję państwa ramowego Polski w ramach Eurokorpusu porzucił. Państwo ramowe wydziela natomiast swój personel dowództwa Eurokorpusu wraz ze zdolnościami bojowymi. Stowarzyszone - nie. Wiodącą ideą, która towarzyszyła utworzeniu Eurokorpusu, było wzmocnienie zdolności Unii Europejskiej oraz organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego do prowadzenia operacji militarnych, w tym misji humanitarnych i ratowniczych, misji przywracania i utrzymywania pokoju oraz możliwej realizacji zadań w ramach kolektywnej obrony NATO. Jest on zatem fundamentem, na którym w przyszłości mogą powstać siły zbrojne Unii Europejskiej.

W efekcie przyjęcie statusu państwa ramowego umożliwi Rzeczypospolitej Polskiej skuteczniejsze oddziaływanie na kierunki zaangażowania Eurokorpusu, w tym w ramach kolektywnej obrony NATO, oraz na utrwalenie zaangażowania jego dowództwa w łańcuch dowodzenia NATO z możliwością udziału w realizacji polityki odstraszania i obrony na flance wschodniej, co dziś dla nas jest niebagatelne. Polskie siły zbrojne są praktycznie pozbawione skutecznej obrony cyberprzestrzeni, czego nie można powiedzieć o innych państwach europejskich. Lewica za każdym razem podkreśla, że szansą na prawidłowy rozwój Rzeczypospolitej Polskiej jest dalsze pogłębienie integracji europejskiej, która jest najwłaściwszą odpowiedzią na obecne uwarunkowania gospodarcze i polityczne, oraz umiędzynarodowianie takich konfliktów i kryzysów jak na wschodniej granicy Polski z Białorusią. Dotychczas rząd prowadził politykę zgoła inną. Przystąpienie do tego traktatu jest niewątpliwie polską racją stanu, ale nie przykryje napiętych stosunków z Unią Europejską.

Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Krystian Kamiński, koło Konfederacja. Bardzo proszę.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mamy przystąpić do formuły kooperacji wojskowej ograniczonej do Unii Europejskiej zdominowanej przez państwa starej Unii, wobec których rząd PiS do tej pory się dystansował, uzasadniając to niezrozumieniem przez Francję czy Niemcy naszych uwarunkowań geopolitycznych oraz ich niechęcią do zaangażowania. Aczkolwiek w przypadku ostatnich rozmów Francji i Niemiec bezpośrednio z Rosją nad naszymi głowami, ale jednak o nas, mam wrażenie, że to zaangażowanie jest nazbyt. Na płaszczyźnie współpracy w dziedzinie obrony doszło jednak z tymi państwami do różnych zgrzytów. Przypominam chociażby zerwanie negocjacji w sprawie zakupu francuskich śmigłowców. Nie oceniam tu samej decyzji, ale forma jej podjęcia, realizacja ogłoszenia była jednak, nazwijmy to, nie najlepsza. W tym kontekście na najważniejszej płaszczyźnie bezpieczeństwa zachowanie rządu wygląda jak zachowanie człowieka, który odbija się od ściany do ściany, który sam właściwie nie wie, czego by chciał. Nasuwa się pytanie: Co zatem się zmieniło, że rząd dokonał tak radykalnej korekty własnej polityki? Jakie konkretne propozycje zaangażowania Eurokorpusu, jeśli chodzi o nasz teatr strategiczny, zostały złożone, że państwo stwierdzili, iż warto w ten projekt wejść? Dziękuję. Dziękuję. Pan poseł Janusz Korwin-Mikke. Wysoka Izbo! Kontynuując myśl kolegi Kamińskiego, chciałbym zwrócić uwagę, że Eurokorpus nie odegra żadnej roli w wojnie ze Stanami Zjednoczonymi, Rosją czy Chinami, natomiast może się bardzo przydać, jeżeli Unia Europejska zechce zrobić porządek np. z rządem Kaczyńskiego, który źle zajmuje się wymiarem sprawiedliwości w Polsce. Do tego Eurokorpus przyda się jak najbardziej.

Proszę państwa, zdajmy sobie sprawę, że jest pewna różnica między stanem Ameryki a krajem Unii Europejskiej. Stany amerykańskie nie są niepodległe, podobnie jak kraje Unii Europejskiej, bośmy stracili niepodległość, podpisując traktat lizboński. Niemniej stany amerykańskie nie mają własnej armii, a rząd federalny ma. W Europie jest odwrotnie. Unia nie ma własnej armii, a poszczególne kraje mają swoje armie. I dopóki tak jest, dopóki jesteśmy uzbrojeni, a Unia nie jest uzbrojona, to możemy się cieszyć dużą dozą autonomii. Z chwilą kiedy będzie odwrotnie i to Unia będzie miała silniejsze wojska, okaże się, że nie będziemy mieli już nic do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Pan poseł Paweł Zalewski w imieniu koła Polska 2050.

Koleżanki! Koledzy! W 2008 r. rozpoczęliśmy negocjacje, a później procedurę legislacyjną, która miała na celu włączenie nas do Eurokorpusu jako państwa ramowego. W 2016 r., tuż po objęciu władzy przez PiS, koleżanki i koledzy, zrezygnowaliście z tego. Dzisiaj do tego wracacie. Wy jej nie rozumiecie. Nie wiecie, czym jest Unia Europejska, nie wiecie, że Unia Europejska stwarza szanse i jest po stronie rozwiązań, a nie tworzy problemy. Niedawno premier Rzeczypospolitej mówił, że Unia Europejska chce wywołać III wojnę światową z Polską.

Dzisiaj ciekawe, z jakiego powodu do tego Eurokorpusu chcecie wrócić.

Dzisiaj słyszałem wywiad wiceministra spraw zagranicznych, który opowiadał, jakie to Polska ma wspaniałe relacje z krajami Unii Europejskiej.

Dzisiaj Unia Europejska jest tym miejscem, które daje Polsce możliwość wywarcia realnej presji na Łukaszenkę. Ale wy z tej presji nie chcecie skorzystać. Nie rozmawiacie z Niemcami, Francuzami czy Komisją Europejską o tym, aby stworzyć realne, bardzo silne sankcje, które mogłyby Łukaszenkę powstrzymać. Cały ciężar obrony polskiej granicy zrzucacie na służby mundurowe, które się na niej znajdują i jej bronią. Otóż dzisiaj widać, jak bardzo nie jesteście kompetentni, jak bardzo waszą polityką europejską przez ostatnie lata zaszkodziliście Polsce. W imieniu koła Polska 2050 deklaruję poparcie dla tej ustawy. Przechodzimy do pytań. Wyznaczam czas - 1 minuta. Pierwsze pytanie tradycyjnie zada pan poseł Jan Szopiński, klub Lewica. Wysoka Izbo! Chciałbym pogratulować rządowi tego, że w okresie toczenia licznych sporów z Unią Europejską zdecydował się na ratyfikację traktatu w sprawie Eurokorpusu. Jest to krok bez wątpienia słuszny i oczekiwany od lat przez Polaków. Chciałbym zapytać: Czy w związku z zapowiedziami pana wicepremiera Kaczyńskiego dotyczącymi tworzenia najliczniejszej i najsilniejszej armii w Unii Europejskiej Polska zamiesza starać się o jakiś specjalny status w ramach tej organizacji? Pan poseł Rafał Adamczyk, klub Lewica. Wysoka Izbo! W uzasadnieniu do ustawy czytamy: Eurokorpus jest przeznaczony do prowadzenia misji i operacji pod auspicjami Unii Europejskiej, NATO i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przystąpienie do Eurokorpusu na prawach państwa ramowego będzie wyrazem znaczenia, jakie Rzeczpospolita Polska przykłada do wzmacniania bezpieczeństwa europejskiego, oraz podkreśleniem woli współpracy wojskowej z państwami Unii Europejskiej. Panie Ministrze! Powstaje tylko pytanie: Czemu tak długo czekaliśmy na to, żeby taki projekt ustawy się pojawił w Sejmie? Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

I trudno nie oprzeć się wrażeniu, że to był minister, który jak mało kto zaszkodził Polsce, zaszkodził polskim interesom. Także jeżeli chodzi o tę decyzję dotyczącą wstrzymania prac w kierunku tego, aby Polska stała się państwem ramowym tej umowy, to widać wyraźnie, że to była zła decyzja, która szkodziła Polsce, i dzisiaj tę decyzję rząd na szczęście zmienia. Natomiast moje pytanie jest takie: Które jednostki mogą być tymi jednostkami, które staną się częścią Eurokorpusu? Dziękuję bardzo. Zapraszam. Wysoka Izbo! Rządowy projekt, o którym jest mowa, to doskonały przykład tego, jak rząd zmienia zdanie i swoje stanowisko, sprawiając przy tym, iż nasz kraj w oczach innych staje się mało wiarygodnym partnerem. W 2017 r. ówczesny szef Ministerstwa Obrony Narodowej Antoni Macierewicz chciał ograniczenia naszego zaangażowania w Eurokorpusie. Z kolei w 2019 r. zaczęto zmieniać narrację, bo struktura ta zaczęła zyskiwać coraz większe znaczenie w łańcuchu dowodzenia NATO.

Wysoka Izbo! Eurokorpus to niezwykle ważny element bezpieczeństwa państw Unii Europejskiej i NATO. On ma jeszcze większe znaczenie dla Polski. Dlatego Polska podjęła decyzję o przystąpieniu do Eurokorpusu na prawach państwa stowarzyszonego w 2002 r., a później w 2008 r. podjęła decyzję, i uzgodniła to z partnerami, że będziemy pełnoprawnym członkiem Eurokorpusu. Znalazły się jednak siły polityczne i ludzie, którzy uderzyli w te wysiłki i starania Polski, którzy podważyli polską rację stanu. Byli to minister Antoni Macierewicz i rząd PiS, którzy postanowili przerwać polskie dążenia do objęcia pełnego członkostwa w Eurokorpusie.

Dziękuję. Pan poseł Michał Krawczyk, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Polska zabiega o pełnoprawne członkostwo w Eurokorpusie, czyli w wojskowych siłach szybkiego reagowania NATO i Unii Europejskiej.

Kiedy wywiążecie się państwo z obietnic składanych od 6 lat fabryce PZL-Świdnik, [[Oklaski]] której obiecujecie, szczególnie przed kolejnymi wyborami, zamówienie śmigłowców bojowych? Państwo obiecujecie zamówienia. Pytam, kiedy się z tego wywiążecie.

Bardzo proszę.

Czy prawdą jest, że w 2016 r. prace nad tą ustawą zablokował pan minister Antoni Macierewicz?

Dziękuję. Pan poseł Andrzej Szejna, Lewica.

Dotyczy to naszego członkostwa w NATO, dotyczy ONZ, Unii Europejskiej, dlatego z dużą przyjemnością przyjęliśmy, jak już podkreśliłem w wystąpieniu klubowym, decyzję o zmianie decyzji pana Antoniego Macierewicza i o ratyfikacji traktatu.

Dziękuję.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przystąpienie Polski do Eurokorpusu jest dla nas szansą na nawiązanie sojuszu współpracy w celu utrzymania pokoju. Nie mamy żadnych sojuszników. A jeżeli ich mamy, to nie chcemy korzystać z ich pomocy. Eurokorpus otwiera nam drzwi do korzystania z doświadczeń innych, silniejszych partnerów w sytuacjach kryzysu. Nasuwa się pytanie, czy rząd PiS będzie chciał korzystać z wiedzy i doświadczeń ekspertów, którzy mają już opanowane strategie. Czy nadal będziecie udawać, że potraficie sprostać problemom, np. napływu uchodźców? Czy będziecie ignorować sygnały proponujące wsparcie? To świadczy o waszej bezsilności i o braku kompetencji. Korzystajcie z wiedzy i doświadczeń innych krajów. Obronność to nie jest walka wprost, to strategia. Niech to się odbywa jak najmniejszym kosztem (Dzwonek) naszych obywateli.

Przepraszam.

Czy naprawdę choć raz nie możecie się zastanowić, zanim zrobicie coś głupiego?

Jeśli oni są zachwyceni tym pomysłem, jeśli oni mówią, że to jest pogłębianie integracji, jeśli ci sami ludzie, którzy zawsze się cieszą, kiedy Unia nam dowali, wyda niesprawiedliwy wyrok albo chce pogłębienia ingerencji w polskie sprawy. Pan poseł Cezary Grabarczyk, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Polska potrzebuje ściślejszej integracji z Unią Europejską. Dobrze więc, że dziś debatujemy nad ustawą ratyfikującą pełne członkostwo Polski w Eurokorpusie.

Bardzo proszę, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pan prezydent Lecz Kaczyński po objęciu urzędu mówił o potrzebie włączenia Polski do Eurokorpusu. Ta sprawa była wielokrotnie podnoszona zarówno przez pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jak i przez pana premiera Jarosława Kaczyńskiego.

Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Proszę państwa, zdecydujmy się.

W 2008 r. oczywiście rząd Platformy Obywatelskiej rozpoczął już formalne negocjacje. W 2016 r., proszę państwa, minister Macierewicz podjął w moim głębokim przekonaniu niezwykle słuszną decyzję, jako że Eurokorpus w tym czasie z jednostki, która miała brać udział w misjach, zapewniać bezpieczeństwo, stał się właściwie korpusem szkoleniowo-misyjnym, i to jedynie we francuskiej Afryce. Zmieniła się sytuacja, zmieniły się zadania Eurokorpusu, Prawo i Sprawiedliwość podjęło słuszną decyzję: będziemy w ważnym korpusie. A nie tak jak kiedyś - mieliśmy być w korpusie szkoleniowym. Bardzo proszę. Dziękuję, pani marszałek.

Gdzie są te statki, czołgi, helikoptery, które tak były zapowiadane? No i kiedy planujemy spełnić warunki, które umożliwią tak naprawdę uzyskanie pełnoprawnego członkostwa? Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Odpowiedzi na zadane pytania udzieli sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej minister Wojciech Skurkiewicz. Zapraszam, panie ministrze.

W pierwszych słowach pragnę podziękować poszczególnym klubom za poparcie inicjatywy ratyfikacji. Dziękuję, bo to jest ważne, to jest bardzo ważny gest i mam nadzieję, że Izba przyjmie to jednomyślnie, tak jak to miało miejsce wczoraj na posiedzeniu połączonych komisji. Wysoka Izbo! Chciałbym zwrócić uwagę na kilka kwestii w kontekście pytań, które padały.

Szanowni Państwo! Mówił już o tym pan przewodniczący Jach - dyskusja na temat zaangażowania Polski w działania Eurokorpusu to rok 2006, później, rok 2008 to rozpoczęcie negocjacji odnośnie do tego, aby Polska została stałym przedstawicielem, państwem ramowym. Tylko pamiętajcie o waszej skuteczności, kiedy rządziła koalicja PO-PSL.

Nie byliście w stanie tego przeprowadzić. Szanowni państwo, bo gdyby to było możliwe, to pewnie minister Siemoniak czy wcześniej minister Klich by to zrealizował i byśmy byli pewnie państwem ramowym już od roku 2014 czy 2015. Proszę pamiętać o jednej bardzo kluczowej kwestii: zmieniło się podejście Eurokorpusu do spraw dotyczących funkcjonowania Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 21. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim (druki nr 1227 i 1685) Uprzejmie proszę pana posła Andrzeja Kosztowniaka o przedstawienie sprawozdania komisji. Bardzo dziękuję. Szanowna Pani Marszałek! Mam przyjemność przedłożyć sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim, druk nr 1227. Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu, skierował w dniu 28 maja 2021 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych do pierwszego czytania. Komisja Finansów Publicznych po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 27 października 2021 r. wnosi: Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Jednocześnie uprzedzam, że będę ściśle przestrzegać czasu wypowiedzi. W pierwszej kolejności stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawi pan poseł Wiesław Janczyk. Bardzo proszę. Dziękuję uprzejmie. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość przedstawić w drugim czytaniu stanowisko klubu w zakresie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim. Pierwsze czytanie już za nami. Komisja Finansów Publicznych pracowała nad tym dokumentem. Przypomnę może tylko, że ustawa dotyczy wykonania przepisów, które uzgodnią obecny stan faktyczny rzeczy z konsytuacją. Nastąpiła taka sytuacja, że po zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim w roku 1997 prezes Narodowego Banku Polskiego nie wydał zarządzenia odnośnie do postępowania po przyjęciu do opinii, do ekspertyzy znaków pieniężnych falsyfikowanych. Dzisiaj właściwie kończymy prace nad nową regulacją, która da możliwość ministrowi sprawiedliwości po konsultacji z ministrem spraw wewnętrznych i administracji oraz prezesem Narodowego Banku Polskiego wydania rozporządzenia w tej sprawie, które określi warunki i tryb postępowania z tak przyjętymi do ekspertyzy, do opinii znakami pieniężnymi co do ich przechowywania, co do ewentualnego zwrotu w sytuacji nieuprawnionego podejrzenia o to, że są to falsyfikaty. Szanowni Państwo! Klub Prawo i Sprawiedliwość w drugim czytaniu składa jeszcze jedną poprawkę. Składam wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim, druki sejmowe nr 1227 i 1685, pani marszałek, bez odsyłania do komisji poprawek i wniosków zgłoszonych do tego projektu ustawy i po doręczeniu ich posłom. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję, panie pośle. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska przedstawi pan poseł Wojciech Saługa. Szkoda, że pan poseł, mówiąc o tej poprawce, nie powiedział, czego ona będzie dotyczyć, bo ustawa jest tak krótka i tak zwięzła, że może by to było dość łatwe, a tak to po prostu nie wiemy. Wysoka Izbo! Projektowana ustawa jest reakcją Komisji do Spraw Petycji naszego Sejmu na petycję skierowaną przez pana Sebastiana Adamowicza, którą komisja uznała za zasadną. Zasadniczym skutkiem prawnym projektowanej ustawy będzie eliminacja przepisu sprzecznego z konstytucją.

Propozycja ustawy nakłada na ministra sprawiedliwości obowiązki wydania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii prezesa Narodowego Banku Polskiego, odpowiedniego rozporządzenia w tej sprawie do 3 miesięcy od czasu jej ogłoszenia. Przynajmniej tak jest w tej chwili. Oczywiście bardzo ważne będzie, jak to rozporządzenie będzie wyglądać. Powinno ono oczywiście precyzyjnie rozgraniczyć kilka etapów procedury. W odniesieniu do pierwszego etapu, gdy dochodzi do zatrzymania podejrzanego znaku pieniężnego, rozporządzenie określi sposób zabezpieczenia tego znaku, tak aby na dalszym etapie nie doszło do jego podmiany, i wydawania potwierdzenia zatrzymania poprzez sporządzenie protokołu.

W odniesieniu do drugiego etapu, gdy zatrzymany znak musi zostać przekazany do ekspertyzy celem potwierdzenia lub wykluczenia fałszerstwa, rozporządzenie określi sposób jego przekazywania, warunki, jakie musi spełnić podmiot dokonujący ekspertyzy, oraz sposób jej dokumentowania. Rozporządzanie określi także dalszy tryb postępowania: albo zwrot zatrzymanego znaku pieniężnego, gdy ekspertyza potwierdzi jego autentyczność, albo zatrzymanie na potrzeby prowadzonego postępowania. Podczas pierwszego czytania głównie dyskusję wzbudzał termin wejścia w życie tej ustawy.

Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska poprze przedmiotową ustawę. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu parlamentarnego Lewicy wobec komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim. Projektowana ustawa jest reakcją Komisji do Spraw Petycji na petycję skierowaną do Sejmu przez pana Sebastiana Adamowicza, którą komisja uznała za zasadną. Celem ustawy jest dostosowanie ustawy o Narodowym Banku Polskim do wymogów wynikających z przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ wskazane w zmienianej ustawie zarządzenie prezesa NBP nie może być źródłem powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z art. 87 ust. 1 oraz art. 93 ust. 2 Konstytucji RP. Omawiany projekt jest bardzo krótki. Są to dwa artykuły, z których pierwszy daje upoważnienie właściwemu ministrowi do wydawania odpowiedniego rozporządzenia określającego zasady i tryb postępowania przy zatrzymaniu znaków pieniężnych podejrzanych co do autentyczności oraz postępowania z fałszywymi znakami pieniężnymi. Projekt przewiduje, że rozporządzenie powinno zostać wydane przez ministra sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz po zasięgnięciu opinii prezesa NBP. Drugi artykuł projektu mówi o vacatio legis.

Jako uzasadnienie komisja wyjaśniła, że tak długie, podkreślam: tak długie, vacatio legis zaproponowano ze względu na konieczność opracowania i wydania rozporządzenia. W kolejnym druku, czyli druku nr 1685, art. 2 zmieniono i zaproponowano 3-miesięczny okres vacatio legis od dnia ogłoszenia. Nasuwa się zatem pierwsze pytanie, które kieruję do ministra sprawiedliwości. Tak jak wspomniałam, ustawa jest krótka. Jednak kluczowe jest to, jak będzie wyglądało rozporządzenie. Zgodnie z opinią Biura Analiz Sejmowych ustawa będzie miała wpływ nie tylko na polską walutę, ale także na inne waluty, w tym euro. Dlatego w trakcie przygotowania rozporządzenia należy uwzględnić szereg aktów prawnych Unii Europejskiej, takich jak np. decyzja Rady w sprawie ochrony euro przed fałszowaniem, rozporządzenie Rady z 2001 r. ustanawiające środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem przez państwa członkowskie, które przyjęły euro jako swoją walutę, ale również rozporządzenie dla tych państw, które nie przyjęły euro jako swojej jedynej waluty, a także dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 2014 r. w sprawie prawnokarnych środków ochrony euro i innych walut przed fałszowaniem. Biuro Analiz Sejmowych wskazuje również na obowiązek konsultacji projektu rozporządzenia z Europejskim Bankiem Centralnym na podstawie Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Konkludując, zwracam się z pytaniami do ministra sprawiedliwości. Czy projekt rozporządzenia, o którym mowa w ustawie, jest już gotowy? A jeżeli nie, to na jakim etapie przygotowania jest? Czy rozporządzenie uwzględnia wszystkie wymienione dokumenty prawa Unii Europejskiej i na jakim etapie konsultacji, jeżeli one się już odbywają, znajduje się projekt rozporządzenia? Czy został on przygotowany w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych? Czy prezes NBP zaopiniował rozporządzenie? Czy zostało ono skonsultowane z Europejskim Bankiem Centralnym? Uprzejmie dziękuję. Zapraszam, panie pośle.

Bardzo dziękuję. Pani Marszałek! Panie Ministrze!

Uważamy go za niezwykle potrzebne rozwiązanie. Wyrażamy wdzięczność zarówno osobie, która zasygnalizowała to komisji, jak i samej Komisji do Spraw Petycji za podjęcie wysiłku przygotowania tego projektu. Ma on walor porządkujący nieścisłości w sprawie wydawania zarządzeń przez prezesa NBP w sprawie zatrzymywania znaków pieniężnych podejrzanych co do autentyczności oraz postępowania z fałszywymi znakami pieniężnymi. Odtąd rozporządzenie w tej sprawie będzie wydawał minister sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii prezesa Narodowego Banku Polskiego. Uważamy, że jak najszybciej to rozwiązanie powinniśmy uchwalić. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.

Wysoki Sejmie! Jako prawnik i kryminalistyk mam pewien problem z tym projektem ustawy, bo w mojej ocenie on po prostu dotyczy sytuacji, które za chwilę odejdą w niebyt. To, co kiedyś było plagą, dzisiaj na szczęście jest tylko marginesem. Fałszowanie znaków pieniężnych, kiedyś i na przestrzeni wieków zagrożone niezwykle surowymi karami, bo będące ogromnym problemem społecznym, dzisiaj odchodzi do legendy. Odchodzi zresztą do legendy razem z gotówką, czyli z samymi znakami pieniężnymi.

A w 2020 r. był to już statystycznie nieco ponad jeden podrobiony nominał. Tego się już po prostu nie robi, dlatego że gotówka przestaje mieć znaczenie w nowoczesnym świecie. Wiem, że pan prezes Narodowego Banku Polskiego kocha gotówkę, że projektuje nowe banknoty i monety. Nawet specjalną ustawę o ochronie gotówki przeforsował przez Sejm, ustawę, co warto dodać, nikomu w obecnym stanie prawnym niepotrzebną. Ale postępu technologii po prostu nie da się zatrzymać. Gotówka jest i będzie marginalizowana, bo taki jest los gotówki w świecie terminali płatniczych, cyberwalut czy mikropłatności. Jego idea jeszcze 50 lat temu byłaby absolutnie słuszna i ze wszech miar uzasadniona, natomiast dziś jest po prostu marginalna - i dalej słuszna, choć archaiczna. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Od 6 lat każde przekazanie kompetencji, w jakiejkolwiek sprawie, obecnemu ministrowi sprawiedliwości w naszym kraju wiązało się, w bliższej lub dalszej przyszłości, z głębokimi kryzysami w koalicji rządzącej, problemami obywateli Rzeczypospolitej oraz osłabieniem pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej. Lista takich przypadków jest niezmiernie długa. Dlatego chciałbym się dowiedzieć, dlaczego sposób postępowania z podrobionymi środkami płatniczymi wymaga uchwały wydawanej przez ministra Ziobrę, a nie może być, tak jak do tej pory, określany przez wewnętrzne przepisy Narodowego Banku Polskiego. Jeśli projektodawca zakłada, że prezes NBP nie jest kompetentny do podejmowania takich decyzji, to z jakiego powodu nie zaproponował rozwiązania tego problemu na poziomie ustawowym? Dziękuję bardzo. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Bardzo dziękuję. Panie Ministrze! Fałszowanie znaków pieniężnych jest oczywiście poważnym problemem, zwłaszcza dla osób, które są ofiarami tego procederu. Dlatego bardzo bym prosił o udzielenie informacji, w formie pisemnej, panie ministrze, ile było takich spraw, w których zachodziło podejrzenie, że ma się do czynienia właśnie z fałszywką - w tym roku, od stycznia do końca października. W ilu przypadkach, w których było takie podejrzenie, to rzeczywiście się potwierdziło?

Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Zastanawiający jest czas tej nowelizacji. Przypadkiem zbiega się to z okresem, kiedy zaczęło się robić ciepło wokół prezesa Glapińskiego - prezesa, który w międzynarodowym rankingu został zaliczony do grona najgorszych prezesów banków centralnych w Europie; prezesa, który jeszcze we wrześniu drwił z pomysłu podnoszenia stóp procentowych, a potem podniósł je dwa razy na przestrzeni miesiąca; wreszcie prezesa, za którego kadencji mamy najwyższą inflację od 20 lat i który swoimi decyzjami powoduje, że jego wiarygodność w oczach Polaków topnieje w ekspresowym tempie. Teraz słyszymy, że pan prezes ma dostać od prezydenta i większości sejmowej w nagrodę drugą kadencję w Narodowym Banku Polskim.

Nie ma pana posła. Pan poseł Krzysztof Grabczuk, Koalicja Obywatelska. O udzielenie odpowiedzi na pytania uprzejmie proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pana ministra Michała Wosia. Bardzo proszę, panie ministrze. To nie uchwała, panie pośle, a rozporządzenie. Zarządzenie nie może być źródłem powszechnie obowiązującego prawa. Mianowicie pan poseł Gramatyka mówił, jak bardzo nieistotna jest ta ustawa, natomiast pan poseł Suchoń mówił, jak bardzo jest ona istotna. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie ministrze. W dyskusji złożono wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy bez odsyłania go do komisji po doręczeniu zgłoszonych poprawek. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 22. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (druk nr 1742) Uprzejmie proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Macieja Wąsika o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przedstawiam państwu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Przepisy projektowanej ustawy stanowić będą odpowiedź na współczesne wyzwania dla cyberbezpieczeństwa związane z postępem technologii informatycznych i powszechnością dostępu do nich. Działalność przestępcza w cyberprzestrzeni w znacznej części nie tyle polega na tworzeniu nowego rodzaju przestępstw, co dostarcza nowych metod i środków lub stanowi nową przestrzeń do ich popełnienia. W związku z tym wymaga specjalistycznego podejścia w kwestii rozpoznania środowiska internetowego, identyfikowania pojawiających się w nich nowych zagrożeń oraz skutecznego na nie reagowania. Pojawiające się wraz z nieustannym rozwojem technologii nowe rozwiązania z dziedziny informatyki stają się coraz częściej zarówno narzędziem wykorzystywanym do popełnienia przestępstw, jak i celem działalności przestępczej i stanowią coraz większe wyzwania w zakresie wykrywania i zwalczania przestępstw. Należy zauważyć także stale i dynamicznie rosnącą skalę przedmiotowego zjawiska. W 2013 r. Policja wszczęła 18 226 postępowań przygotowawczych w sprawach związanych z tego rodzaju przestępczością, w trakcie prowadzenia których stwierdzono łącznie 52 291 przestępstw. Natomiast w 2020 r. liczby te wynosiły odpowiednio 53 687 wszczętych postępowań przygotowawczych oraz 107 518 przestępstw stwierdzonych. Skuteczne reagowanie na tego rodzaju zagrożenia wymaga wprowadzenia gruntownych zmian w strukturach Policji pozwalających na znaczne skrócenie czasu reakcji na zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni, umożliwiających szybsze i efektywniejsze podejmowanie działań. Niezbędne jest zatem ustanowienie jednolitej w skali kraju jednostki organizacyjnej Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, odpowiedzialnej za realizację zadań w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości popełnionej przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej, wykrywanie i ściganie sprawców tej przestępczości oraz wspieranie w tym zakresie pozostałych jednostek organizacyjnych Policji. Dotychczas działania w tym obszarze realizowane były przez biura zwalczania cyberprzestępczości Komendy Głównej Policji i komórki organizacyjne komend wojewódzkich Policji. Struktury te miały zatem charakter rozproszony i nie zapewniały jednolitego podejścia, jak ma to miejsce przykładowo w odniesieniu do przestępczości zorganizowanej przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Panie i Panowie Posłowie! Podniesienie efektywności działania Policji w zakresie zwalczania cyberprzestępczości wymaga wprowadzenia zmian nie tylko w odniesieniu do struktury tej formacji, ale także w kontekście naboru do służby: skutecznego i profesjonalnego, wyszkolenia oraz wzmocnienia motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy. Konieczne jest usprawiedliwienie i dostosowanie do współczesnego świata cyfrowego postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, jak również już pełniących służbę funkcjonariuszy. Celem będzie pozyskanie kandydatów na stanowiska, na których wymagane są specjalistyczne wykształcenie, umiejętności lub kwalifikacje pożądane ze względu na potrzeby kadrowe Policji w zakresie cyberbezpieczeństwa. W przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości na stanowisko związane z bezpośrednim rozpoznawaniem, zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości popełnionej przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej, a także wykrywaniem i ściganiem sprawców tej przestępczości, zrezygnowano z konieczności przeprowadzania części etapów naboru, tj. testów wiedzy oraz testu sprawności fizycznej. Osoba ta nie będzie przechodziła również procesu adaptacji służbowej w oddziale prewencji Policji albo samodzielnym pododdziale prewencji Policji. Natomiast dodano w tym przypadku niezwykle istotny etap w postaci sprawdzenia wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, funkcjonowania systemów informatycznych, systemów teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz znajomości języka obcego obejmującej te dziedziny. Szczególna ścieżka naboru w przypadku funkcjonariusza starającego się o przyjęcie do służby w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości wynika z charakteru zadań stawianych przed tą jednostką organizacyjną Policji, a także ma pomóc w pozyskaniu kandydatów do służby o szczególnych umiejętnościach, które nie wymagają powiązania ich np. ze sprawnością fizyczną czy umiejętnościami typowymi dla służby prewencyjnej. Łącznie przewiduje się otworzenie 1800 nowych etatów przeznaczonych do walki z cyberprzestępczością w CBZC. Wysoka Izbo! Utworzenie nowej jednostki organizacyjnej Policji wymaga także posiadania adekwatnych środków finansowych pozwalających na jej wyposażenie oraz wprowadzenie motywacyjnego systemu uposażeń. Aby móc realizować powyższe zadania, konieczne jest zwiększenie dofinansowania Policji w tym zakresie. Obecne rozwiązania systemowe skutecznie utrudniają pozyskanie do służby w Policji specjalistów w dziedzinie cyberprzestępczości. Dlatego projekt zakłada przyjęcie zmodyfikowanego mechanizmu określenia wysokości uposażeń funkcjonariuszy bezpośrednio zwalczających cyberprzestępczość. Wprowadzone zostanie świadczenie związane z pełnieniem służby w CBZC w miesięcznej wysokości nie niższej niż 70% i nie wyższej niż 130% przeciętnego uposażenia policjantów, którego wysokość będzie uzależniona od oceny wywiązywania się policjanta z obowiązków oraz realizacji powierzonych mu zadań i czynności.

Wysoka Izbo! Funkcjonariuszom nowopowstałego CBZC przysługiwać będzie w pełni możliwość prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz administracyjno-porządkowych wynikających z dotychczas obowiązującej ustawy o Policji na dotychczas przewidywanych zasadach. Proponowana zmiana art. 19 ust. 1 ustawy o Policji poprzez uzupełnienie katalogu przestępstw, w przypadku których możliwe jest zastosowanie kontroli operacyjnej, ma na celu zwiększenie szybkości i efektywności reagowania Policji w zakresie zwalczania i zapobiegania cyberprzestępczości oraz wyposażenia ich w niezbędne narzędzia w tym celu. Dlatego konieczne jest umożliwienie Policji realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych w pełnym zakresie w odniesieniu do takich przestępstw jak nawiązywanie kontaktu z małoletnim poprzez Internet w celach pedofilskich, publiczne propagowanie pedofilii, celowe powiadamianie o nieistniejącym zagrożeniu, tzw. fałszywe alarmy, niszczenie danych informatycznych i zakłócanie ich przetwarzania, zakłócanie funkcjonowania systemów teleinformatycznych, oszustwo komputerowe.

W dalszym ciągu będzie miała ona charakter subsydiarny, tzn. może być stosowana, kiedy inne środki okażą się bezskuteczne albo będą nieprzydatne i sformalizowane. Ściśle określony jest m.in. sposób postępowania z uzyskanymi materiałami. Ponadto na każdym etapie prowadzenia kontroli operacyjnej prokuratura ma zagwarantowany dostęp do całości uzyskanych materiałów, a samo zarządzenie kontroli operacyjnej jest uzależnione od decyzji sądu. Szanowni Państwo! Pragnę jednak podkreślić, że przedstawiony projekt ustawy ma na celu zwiększenie efektywności działania Policji, a co za tym idzie - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców Polski. Skutkiem przyjęcia ustawy będzie zwiększenie zdolności państwa do reagowania na zdarzenia w sferze cyberprzestępczości oraz zapewnienie na terytorium całego państwa jednolitego systemu przygotowania do takich działań. Mając to na uwadze, proszę Wysoką Izbę o poparcie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Uprzejmie dziękuję, panie ministrze. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół.

Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jestem przekonany, że nikomu na tej sali nie trzeba udowadniać, że pojawił się narastający problem związany z cyberprzestępczością i że nie jest to wyłącznie nasz, polski problem, ale jest to coś, co wykracza daleko poza granice naszego państwa.

Świat się zmienia, a my musimy za tymi zmianami nadążyć, również w wymiarze bezpieczeństwa, i dostosować nasze służby do pojawiających się nowych wyzwań.

Kluczem do zwalczania cyberprzestępczości będzie nowoczesna formacja uzbrojona w odpowiednie narzędzia prawne, odpowiednio wyposażona i zmotywowana. Zgodnie z zapisami projektu ustawy proponujemy jako środowisko polityczne powołanie jednolitej w skali kraju jednostki organizacyjnej Policji, nowej służby w jej ramach, odpowiedzialnej za rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości oraz ściganie sprawców tych przestępstw. Tym, co będzie wyróżniało tę formację od wszystkich innych rodzajów służby w Policji, będzie zakres wykonywanych zadań, system rekrutacji i szkolenia funkcjonariuszy, a także wynagrodzenie zwiększające atrakcyjność służby w stosunku do zarobków dostępnych na rynku pracy. Do zadań Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości będzie należeć m.in. zwalczanie przestępstw związanych z oszustwami w sieci, kradzieżą tożsamości czy też walka z pedofilami, którzy często poszukują swoich ofiar w Intrenecie. System rekrutacji do nowej formacji w ramach Policji ma być dostosowany do zadań, jakie przed tą formacją chcemy postawić. W ten sposób racjonalizujemy system naboru.

W ustawie zakłada się, że w ciągu 4 lat formacja uzyska docelową liczbę wysoko wykwalifikowanych funkcjonariuszy. Warto podkreślić, że proponowane zmiany ustawy o Policji są kolejnymi regulacjami prawnymi wpisującymi się w zapisy Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie zwiększenia skuteczności państwa w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości. Panie i Panowie Posłowie! Przestępstwa w sieci są ogromnym wyzwaniem, przed jakim stoi polska Policja, a naszym zadaniem jako władzy ustawodawczej jest dać tej formacji takie regulacje prawne, które pozwolą policji skutecznie zadbać o bezpieczeństwo Polaków w sieci.

Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę.

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Szanowni Państwo!

Ale na początek powiem, że słabe państwo mnoży służby, a można powiedzieć, że państwo autorytarne mnoży służby. Państwo przekonujecie, że kolejna instytucja będzie zwalczać pedofilię w sieci, będziecie państwo przeciwstawiać się wyłudzeniom, kradzieżom, manipulacji różnego rodzaju atakom, cyberzagrożeniom. To nie będzie nowa formacja. W strukturze Komendy Głównej Policji, szanowni państwo, funkcjonuje Biuro do Walki z Cyberprzestępczością, a do zadań tego biura należy: nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie ukierunkowanych na zwalczanie cyberprzestępczości działań prowadzonych przez Policję; prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych pozostających we właściwości biura; inicjowanie i prowadzenie współpracy z organami administracji rządowej, sądami, prokuratorami, instytucjami państwowymi, podmiotami prywatnymi w zakresie zadań pozostających we właściwości biura; prowadzenie współpracy międzynarodowej; prowadzenie całodobowej służby mającej na celu koordynowanie działań Policji itd. Szanowni Państwo! Dziś polska Policja posiada już te narzędzia. Okazuje się, że pan minister Kamiński ani pan minister Wąsik o tym nie wiedzą, że takie narzędzia już państwo macie. Absolutnym hitem, szanowni państwo, jest to, że również wszystkie komendy wojewódzkie mają takie biura. Ilekroć PiS mówi, szanowni państwo, że robi coś dla obywateli, to robi coś faktycznie przeciwko Polakom. Nowa służba ma być po prostu narzędziem do inwigilacji milionów Polaków. W ramach tego będziecie państwo mogli po prostu zaglądać do naszych telefonów, komputerów i będziecie inwigilować Polaków, tak jak robicie to z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Powołanie nowej służby, szanowni państwo, zbiega się w czasie dokładnie z wyciekiem maili ze skrzynki ministra Dworczyka. Czy to jest przypadek? Oczywiście, że nie. Ale czy to jest powód do tego, żeby stworzyć nową instytucję tylko po to, by przykryć błędy w higienicznym zachowaniu państwa przedstawicieli? Nie przestrzegacie podstawowych zasad bezpieczeństwa, więc wpadliście na pomysł, że zrobi to za was nowa służba. Chcecie mnożyć etaty, wydatki, tylko dlatego, że nie potraficie zarządzać tym, co już macie. To wprost zapowiedź nowych problemów. CBA ma dziś tyle wspólnego z antykorupcją, ile IPN z pamięcią i TVP z informacją. Zatem można jasno powiedzieć, że państwa rząd z cyberprzestępczością i jej zwalczaniem ma tyle wspólnego, ile właśnie maile ministra Dworczyka. Szanowni Państwo! Jak będzie ta instytucja wyglądać w rękach Prawa i Sprawiedliwości, można łatwo opisać na przykładzie Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

2020 r. - słynna spowiedź agenta Tomka, tego samego, którego dzisiaj zwalczacie. Agent Tomek mówi: Fundusz operacyjny, który został we mnie wpompowany, był nieograniczony. Luksusowe samochody, droga biżuteria, drogie, markowe ubrania czy zegarki. W styczniu w programie „Superwizjer” na antenie TVN wyemitowano reportaż „Spowiedź agenta Tomka” Agent Tomek oskarżał w nim wówczas byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego oraz byłego wiceszefa Macieja Wąsika o wywieranie na niego nacisków podczas operacji dotyczącej rzekomej willi Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich. Na koniec, szanowni państwo, chciałbym powiedzieć, że państwo proponujecie przeniesienie wszystkich policjantów z biura ds. walki z przestępczością w Policji do nowej służby i poddanie ich weryfikacji, łącznie z wariografem.

Pan mówi, że to pozwoli na lepszą koordynację, ale są inne instytucje i służby (Dzwonek) w naszym kraju, wywiad wojskowy. Pan poseł Krzysztof Gawkowski, klub Lewica. Czas minął. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Bardzo proszę, panie pośle.

Wysoka Izbo! Początek trzeciej dekady XXI w. to, z jednej strony, galopujące procesy globalizacji, z drugiej doświadczenia cywilizacyjne związane z pandemią. W czasie pandemii COVID-19 przyspieszył proces cyfryzacji i dlatego zintegrowane działania dotyczące zapewnienia cyberbezpieczeństwa powinny stać się kluczowym elementem zapewnienia sprawnie funkcjonującego państwa. Obecnie mamy różnego rodzaju zakłócenia, które wpływają na cyberprzestrzeń. Skutki ich często są katastrofalne, ograniczona jest sprawność w funkcjonowaniu administracji publicznej. Brak odpowiedniej cyberochrony może dotykać zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Rolą państwa jest zatem stworzyć takie warunki do przeciwdziałania cyberprzestępstwom, które zapewnią odpowiedni jego poziom i będą odpowiadały na wyzwania współczesności. Bezpieczna cyberprzestrzeń to gwarancja możliwości korzystania z rozwoju technologicznego, szybkiego reagowania i walki z incydentami. Zakłócenie prawidłowości działania systemów informacyjno-sterujących państwa może mieć znaczenie krytyczne i powinniśmy umieć jemu przeciwdziałać. Zasadne zatem wydaje się powołanie służby, która będzie stała na straży cyberbezpieczeństwa i stanowiła nowy odwód w walce z cyfrowymi przestępcami. Nowa jednostka powinna być jednak dobrze zorganizowana i wykonywać zadania bardzo profesjonalnie. W proponowanym projekcie zmiany ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości widać wiele niedoskonałości, które w przyszłości mogą utrudniać sprawne funkcjonowanie służby. Rząd proponuje powołanie w ramach struktur Policji specjalnego nowego rodzaju służby, która będzie zajmowała się cyberbezpieczeństwem, a przecież część takich zadań już funkcjonuje. Zasadne jest zatem pytanie, czy taka służba nie powinna mieć charakteru indywidualnej instytucji. Lewica złożyła już taki projekt ustawy, który zakłada powołanie Agencji Cyberbezpieczeństwa i stworzenie instytucji realizującej zadania prewencyjne i edukacyjne. Stanowiłaby kluczową instytucję cywilnej ochrony interesów RP. W projekcie rządowym większą uwagę poświęca się reakcji na incydenty, a w projekcie Lewicy - działaniom prewencyjnym i szkoleniowym. W uzasadnieniu projektu rządowego autorzy słusznie wskazali, że Policja nie jest w pełni przygotowana do walki z nowoczesnymi formami przestępczości, w tym szczególnie z cyberprzestępczością. Wynika to m.in. z charakteru czynności wykonywanych przez służbę kryminalną, w ramach której funkcjonują komórki organizacyjne zwalczające cyberprzestępczość. Jak piszą w uzasadnieniu autorzy, w większości przypadków działania policjantów zwalczających cyberprzestępczość rozpoczynają się w momencie uzyskania informacji, a to błąd. Autorzy dalej podkreślają, że obecna struktura Policji, liczba etatów oraz posiadane siły i środki nie pozwalają na skuteczną walkę z tą barierą i że ciężko będzie działać w zakresie cyberbezpieczeństwa w rozszerzonym zakresie. Lewica szczególnie mocno zwracała uwagę na zaniedbania rządu w zakresie walki z cyberprzestępczością. 6 lat zaniechań to najmniejszy z zarzutów, jaki można postawić władzy. Warto również przypomnieć o wykorzystywaniu cyberprzestrzeni do walki politycznej, w której ważną rolę odgrywały służby państwowe. Przypominam tu m.in. sprawę senatora Krzysztofa Brejzy oraz wiele innych incydentów wskazujących na upolitycznienie służb mających za zadanie przeciwdziałać zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Mimo wielu wątpliwości uważamy jednak, że wzmocnienie ochrony państwa w zakresie cyberbezpieczeństwa jest ważne i potrzebne. Chcemy pracować nad tą ustawą, ale chcemy też pilnować, aby nowe jednostki nie stawały się miejscem walki z obywatelami w cyberprzestrzeni. Będziemy zgłaszali poprawki dotyczące m.in. nadzoru nad służbą i oznaczenia konkretnych zadań, które będą wykluczały polityczne wpływy partii rządzącej. Nowa służba nie może być batem na niepokornych obywateli wyrażających swoje niezadowolenie w Internecie, a bezpieczna cyberprzestrzeń to polska racja stanu. O takie prawo będzie upominała się Lewica. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.

Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści przedstawiam stanowisko dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Powołanie w miejsce istniejących biur Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, jego usamodzielnienie i wzmocnienie pod względem strukturalnym i finansowym uważamy za dobry krok. Dobrze, że to wreszcie nastąpiło. Oczywiście uważamy, że mogło to nastąpić prędzej, ale dobry jest kierunek, w którym należy podążać.

Tego, takiej strategii i takiego systemu, nam brakuje.

To wymaga bardzo ścisłego i precyzyjnego określenia, ponieważ należy chronić prawa człowieka, prawa obywatela, a zatem każda ingerencja służb, nawet w słusznym interesie, musi być dobrze opisana i nadzorowana.

To powinno być też nieuchronne i powinno iść, jak uważamy, dwutorowo. Projekt ustawy powołujący Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości powinien być jednak procedowany kompleksowo wraz z projektem ustawy o szczególnych zasadach wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Projekt ten zakłada stworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa oraz określa wynagrodzenia osób realizujących zadania z tego zakresu. Oddzielne uchwalanie tych projektów.

Może to spowodować odpływ najlepszych kadr z Policji do innych jednostek sektora publicznego zajmujących się cyberbezpieczeństwem.

Zakłada się też, że siedzibą nowej instytucji będzie Warszawa.

Uważam też, że należy dokładnie sprecyzować i określić - tu już nie chcę wnikać w szczegóły - kryteria przyjęcia do służby.

Wysoka Izbo! Będziemy pracować nad tym projektem. Prosimy oczywiście o skierowanie go do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Dziękuję bardzo, panie pośle. Ciągle, nieustająco pani - kobieta - marszałek. Pan poseł Dobromir Sośnierz w imieniu Konfederacji. Zwalczanie cyberprzestępczości to jest oczywiście ważna sprawa, ale czy na pewno potrzebujemy do tego uroczystego wyodrębnienia kolejnej, nowej służby, takiego papierowego przeniesienia etatów czy nowych odznak na mundury, to już nie jestem przekonany.

Niestety skuteczność walki z cyberprzestępczością nie zależy od stosunków służbowych wewnątrz Policji czy od kroju odznaki na mundurze, więc obawiam się, że to niestety działanie w dużej mierze pozorne. Co jednak ciekawe, w uzasadnieniu ubolewa się, że w większości przypadków - to jest cytat - działania policjantów zwalczających cyberprzestępczość rozpoczynają się w momencie uzyskania informacji o zaistniałym incydencie, tym samym sprawcy czynów zabronionych są o krok przed organami ścigania. No cóż, czy ustawodawca zmierza do tego, żeby policjanci rozpoczynali działania, zanim się dowiedzą, czy też żeby dowiadywali się o incydentach, zanim się one wydarzą? Oba te pomysły brzmią groźnie. Mnie się niestety wydaje, że musimy się pogodzić z tym, że Policja reaguje wtedy, kiedy się coś wydarzy, kiedy przestępstwo zostanie dokonane, inaczej zamieszkalibyśmy chyba w obozie wielkiego brata, który czytałby nam w myślach. Raczej wolelibyśmy tego uniknąć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie pośle.

Panie Ministrze! Zacznę od tego, co jest jak gdyby poza kwestią i co nie ulega wątpliwości. Otóż nie ulega wątpliwości, że w nowoczesnym cyfrowym świecie rośnie i będzie rosła liczba przypadków dotyczących zagrożeń, które w tym nowoczesnym cyfrowym świecie się pojawiają. Warto zacytować wypowiedź jednego z moich przedmówców, który powiedział z tej mównicy, że bezpieczna cyberprzestrzeń to jest polska racja stanu. W pełni podzielam tę tezę, w pełni popieram to hasło, dlatego że postępująca nowoczesność, postępujący w szalony sposób rozwój technologii generuje i na pewno będzie generował zdarzenia, które są z pogranicza świata legalnego i nielegalnego, w tym zdarzenia, które są po prostu przestępstwami. Wzrost liczby tych incydentów, wzrost ich wagi - to również jest poza kwestią, z tym trzeba walczyć. Jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że w państwie polskim dysponujemy wybitnymi specjalistami od raportowania takich właśnie incydentów komputerowych, incydentów teleinformatycznych. Ci specjaliści dziś są skupieni raczej poza strukturami Policji, ale są, funkcjonują. Nie dalej jak wczoraj na posiedzeniu komisji innowacyjności i cyfryzacji debatowaliśmy nad aktem prawnym, który przyznaje im specjalne wynagrodzenia. Ten akt jest również w naszej ocenie ze wszech miar godzien poparcia. Nie przekonuje mnie myślenie, które pan minister zawarł w uzasadnieniu do tej ustawy. Piszą państwo o powołaniu nowej jednostki, o wyposażeniu tej jednostki w sprzęt, o budowie siedziby dla tej nowej jednostki. To nie jest dobre myślenie. Incydenty komputerowe to nie są incydenty, w których wyjaśnieniu, prześwietleniu, w zdobyciu dowodów pomoże nowa siedziba czy sprzęt. To są incydenty wymagające specjalistycznej, unikalnej wręcz wiedzy i obawiam się, że zakreślenie liczby pracowników tej nowej służby na poziomie 1800 etatów nie będzie równorzędne z pozyskaniem z rynku 1800 wykształconych specjalistów, dla których świat cyfrowy nie ma tajemnic.

Budzi to mój przestrach nie dlatego, że uważam, że takich przestępstw nie należy dotykać, ale uważam, że system raportowania tego typu przypadków zastosowania kontroli operacyjnej w naszym kraju jest daleko niedoskonały, a sama kontrola wkracza oczywiście bardzo głęboko w prywatność (Dzwonek) Polek i Polaków. Będziemy pracować nad tym projektem w komisji. Dziękuję bardzo. Zamykam listę osób chcących zadać pytanie. Wyznaczam czas - 1 minuta. Pytanie pierwsze zada pan poseł Jan Szopiński, klub Lewica. Wysoka Izbo! Ustawa wymienia cały szereg kluczowych stanowisk, na których obsadzani mają być oficerowie Policji. Są tutaj wszyscy komendanci wszystkich możliwych formacji, ludzie, którzy powinni być wzorem do naśladowania, lub, jak to się określa w nomenklaturze PiS, ludzie kryształowi. Ustawa ta mówi nam, że ludzie ci nie muszą być poddawani żadnej weryfikacji. Ustawa mówi wprost, że mogą być poddani, ale skoro mogą, to nie jest to obowiązkowe. Zatem chciałbym zadać być może bardzo niepopularne pytanie, ale jednak pytanie: Czy nie jest tak, że zgodnie z tą ustawą w razie potrzeby można mianować równie dobrze wszystkich szwagrów lub osoby potrzebne władzy, które mogą być kiedyś potrzebne do zwalczania opozycji? Poseł Rafał Adamczyk, klub Lewica. Bardzo proszę, panie pośle. Wysoka Izbo! W uzasadnieniu ustawy czytamy: W chwili obecnej polska Policja, jak również organy ścigania innych państw nie są w pełni przygotowane na walkę z nowoczesnymi formami przestępczości, w tym szczególnie z cyberprzestępczością. Panie ministrze: Czy uważa pan, że 1800 etatów, które mają być, mają powstać, to jest liczba wystarczająca do walki z cyberprzestępczością? Czy nie należałoby zwiększyć i bardziej przyśpieszyć aktywowania tych etatów w kolejnych latach? Dziękuję bardzo. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Panie Ministrze! Chciałem zapytać o art. 9, który w istocie może posłużyć do de facto czystki w szeregach funkcjonariuszy, którzy dzisiaj zajmują się przestępstwami związanymi ze światem cybernetycznym. Chciałem zapytać o to, z jakich powodów tak, a nie inaczej ministerstwo i rząd zadecydowali, że w zasadzie po 5 miesiącach będzie można wszystkich funkcjonariuszy wydalić ze służby. Po drugie, czy była prowadzona analiza kompetencji funkcjonariuszy, a jeżeli tak, to w jaki sposób, jak ona wygląda, jakie kompetencje dzisiaj posiadają ci funkcjonariusze?

Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan poseł Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Nie ma. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Problem cyberataków narasta i będzie narastał, jako że coraz większa część naszego życia przenosi się do sieci.

Jak się szacuje, wynosi mniej niż 10%. Ustawa słusznie zapewnia Policji zwiększone fundusze, a więc i możliwości przyciągania ekspertów z rynku prywatnego, jeżeli chodzi o komputery. Mam pytanie. Część banków nie zgłasza nawet ataków, bojąc się utraty dobrego imienia.

Pani poseł Małgorzata Pępek, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Projekt zakłada zatrudnienie 1800 pracowników.

Skąd zamierza się pozyskać taką liczbę wykwalifikowanej kadry, głównie informatyków gotowych do pracy, skoro na wolnym rynku brakuje takich specjalistów? W projekcie proponuje się dodatek służbowy w wysokości od 70% do 130% przeciętnego uposażenia, co nie stanowi nawet połowy, jaką oferuje się dla specjalistów z wysokimi kwalifikacjami. Czy nie skończy się to tak, że będą biura, nowoczesny sprzęt, tylko nie będzie miał kto pracować albo będzie się zatrudniać słabych specjalistów, wypełniając braki? Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Pełnomocnikiem rządu do spraw cyberbezpieczeństwa jest pan minister Cieszyński. Taka kwota padała dzisiaj w nocy, jak mieliśmy dyskusję. Nie powierzyłabym mu nawet jednego grosza do wydania z publicznych pieniędzy. Nie wierzę panu, nie wierzę rządowi, że rzeczywiście to będzie miało na celu zwalczanie cyberprzestępczości. Jak państwo nas o tym przekonają? Może lepiej te pieniądze wydać na leczenie dzieci chorych na SMA, bo to jest bardzo drogie. Uratowalibyśmy życie kilkanaścioro dzieciom. Pan poseł Adam Szłapka, Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze! Cyberprzestępczość to jest oczywiście wyzwanie naszych czasów i słusznie, że rząd zaczął się tym tematem zajmować, tym bardziej że toczy rząd największa afera dotycząca wycieku maili. W związku z tym pytania. Czy ta nowa służba z urzędu zajęłaby się przede wszystkim ściąganiem tych osób, które dysponują tymi mailami, nielegalnie je udostępniają, czy ministrem Dworczykiem, który korzystał z prywatnych środków komunikacji do przesyłania informacji państwowych, w tym informacji niejawnych, czy też ujawnieniem przestępstw, które ukazały się po ujawnieniu tych maili? O to chciałbym zapytać pana ministra - to po pierwsze. A po drugie, mamy w gruncie rzeczy do czynienia z powołaniem w zasadzie nowej służby specjalnej. Pytanie: Jak będzie wyglądała koordynacja tego? Czy to będzie. No na razie tak. Pan poseł Krzysztof Gawkowski, klub Lewica. Pani Marszałek! Panie Ministrze!

Dzięki temu moglibyśmy lepiej koordynować ją z innymi służbami. Zresztą taką propozycję składaliśmy. Prosiłbym, panie ministrze, o odpowiedź na piśmie i rozważenie tego, dlatego że wydaje się, że dodatkowe miejsce w strukturze Policji dla cyberbezpieczeństwa może ograniczać możliwości tej służby. A więc bardzo bym prosił o to, żebyśmy mogli do takiego tematu podejść szerzej, szczególnie że dzisiaj jest pierwsze czytanie i będziemy jeszcze tygodniami nad tym pracowali. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan poseł Tomasz Szymański, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Jak już wiemy, szanowni państwo, nowe Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości ma powstać z wyodrębnionych biur do walki z cyberprzestępczością zlokalizowanych w Komendzie Głównej Policji, a także w wojewódzkich komendach.

To jest zupełnie inna materia. Cyberprzestępczość cechuje się zupełnie innymi, niedookreślonymi dzisiaj walorami i to powinno być pierwszą rzeczą, którą to nowe biuro powinno się zająć. Moje obawy wzbudza, szanowni państwo, jednak fakt, skąd zamierzacie zrekrutować w ciągu roku 500 specjalistów do tego nowego biura.

Pani poseł Krystyna Skowrońska, Koalicja Obywatelska. Panie i Panowie Posłowie! Dzisiaj będziemy głosować nad ustawą o utworzeniu Funduszu Cyberbezpieczeństwa. Pan minister odpowiedzialny za resort cyfryzacji wskazał, że wynagrodzenie pracownika będzie wynosić ok. 40 tys. zł. Wątpliwości budzi również możliwość zrekrutowania kolejnych pracowników do tego centralnego biura.

Pani poseł, dziękuję bardzo. Nie, przepraszam. Bardzo proszę, panie pośle. Wysoka Izbo! Kwestia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni będzie nabierała znaczenia. Z roku na rok tych przestępstw, które są dokonywane właśnie w wirtualnym świecie, będzie coraz więcej, dlatego że coraz więcej korzystamy z usług, które oferuje Internet. Natomiast ja chciałbym przy tej okazji wyrazić ogromne uznanie dla wszystkich policjantów pracujących w różnych obszarach, nie tylko w naszych miejscowościach, również na granicy. I bardzo bym prosił o wyrażanie szacunku dla policjantów, aby nie upolityczniać tej służby, aby mieć szacunek dla funkcjonariuszów doświadczonych, z wiedzą, z zaangażowaniem, a nie oceniać ich tylko pod kątem dyspozycyjności.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Wysoka Izbo!

Natomiast ja chciałam zadać konkretne, merytoryczne pytanie. Czy nie uważacie, że z Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie należałoby wyłączyć i wzmocnić tzw. CERT-u? Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Pani Marszałek! PiS mówi o cyberbezpieczeństwie, a tak naprawdę ostatnie miesiące, panie ministrze, to jest wasza kompromitacja. Cała Polska czyta maile Dworczyka, więc może jest to w tej chwili okazja, szanowni państwo, żebyście w końcu stanęli przed Wysoką Izbą i wyjaśnili tę sytuację. Jak to jest możliwe, że z maili z prywatnej skrzynki wszyscy mogą dowiadywać się o przetargach, o zakupie skomplikowanego sprzętu wojskowego? To jest rzecz absolutnie skandaliczna i przecież przez ostatnie miesiące pokazaliście to, że cyberbezpieczeństwo nie istnieje, a osoby za to odpowiedzialne czy też najważniejsi członkowie Rady Ministrów tak naprawdę skompromitowali się, używając prywatnych skrzynek.

Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Jedynie wnoszę o przemyślenie takiego rozwiązania, aby Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, która ma najlepszych specjalistów w obszarze polskiej administracji rządowej, miała rzeczywiście możliwość takiej biznesowej współpracy z Policją. Zresztą spółka jest podległa panu ministrowi. Ważne jest to, żeby te wszystkie zasoby, które dotyczą cyberbezpieczeństwa w obszarze państwa, zintegrować. Padają słuszne pytania o kadry. Być może dobrym pomysłem jest to, aby rozpocząć od razu po powołaniu tego biura współpracę z kilkoma wyższymi uczelniami, np. z Politechniką Opolską, w zakresie dostarczania kadr do tej bardzo ważnej służby. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję uprzejmie. Pan poseł Michał Krawczyk, Koalicja Obywatelska. Czy kiedy powstanie ta wasza nowa fantastyczna służba do zwalczania cyberprzestępczości, to czy zajmie się ona ministrem Michałem Dworczykiem? Czy zajmie się premierem Mateuszem Morawieckim i pozostałymi członkami polskiego rządu, którzy wykorzystywali swoje prywatne skrzynki do wysyłania informacji, które są wrażliwe z punktu widzenia państwa polskiego? Czy to przypadkiem też nie jest cyberprzestępstwo? I czy nowa służba będzie zajmować się wszystkimi cyberprzestępstwami czy tylko takimi, które są dla was wygodne? Panie Ministrze! Co z tymi pracownikami biura Policji do spraw walki z cyberprzestępczością, którzy nie przejdą weryfikacji pana ministra, którzy nie będą, być może, dyspozycyjni wobec obecnej władzy, którzy nie będą chcieli wykonywać upolitycznionych rozkazów? Co z tymi ludźmi, którzy są związani rozkazami, pracując w Policji? Gdzie ich przesuniecie? Pod koniec panowania ostatnich carów jeden człowiek - Lenin, z którego dużo czerpiecie, powiedział, że państwo, w którym jest więcej policjantów niż nauczycieli, to jest państwo autorytarne i policyjne. Jeszcze u nas tak nie jest, ale staracie się o to, staracie. Fundujecie nam teraz następną służbę, 2 tys. świetnie wykwalifikowanych i dobrze opłacanych ludzi. Po co, skoro w każdej jednostce wojewódzkiej Policji jest już taka komórka do spraw cyberbezpieczeństwa? Ano po to, żeby inwigilować całe społeczeństwo. Paradoksalnie jako opozycja nie powinniśmy się tym martwić, bo w tak półautorytarnym kraju, jakim jest Polska, to najpierw będziecie sprawdzali swoich.

Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Uprzejmie proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji ministra Macieja Wąsika o udzielenie odpowiedzi na postawione pytania. Bardzo proszę, panie ministrze. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za te wszystkie wystąpienia, zarówno klubowe, jak i pytania, które padły z tej mównicy. Chciałem odpowiedzieć w taki sposób, podkreślić jedną rzecz: to nie będzie nowa służba.

To jest Policja, to jest zmiana ustawy o Policji. To ma być służba, która jest utworzona na wzór Centralnego Biura Śledczego, szanowni państwo. Skorzystam z tej okazji, że na tej sali jest twórca Centralnego Biura Śledczego, poseł Marek Biernacki, ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji, który stworzył służbę, która rozprawiła się z polską przestępczością zorganizowaną.

To nie będzie nowa służba, to będą policjanci. Żeby policjanci mogli pracować w tej służbie, muszą być dobrze wynagradzani, bo rynek ssie fachowców. Szanowni państwo, stąd dodatek.

Czyli oprócz tych dodatków, które przewiduje ustawa o CBZC, będzie można czerpać z tego funduszu, o którym wczoraj mówił minister Janusz Cieszyński.

Padło tutaj pytanie, dlaczego chcemy tworzyć ten wyspecjalizowany pion. Dlatego że policjanci w tych biurach, które zwalczają cyberprzestępczość, które są na poziomie komend wojewódzkich, przede wszystkim zarabiają tyle, ile ich koledzy wykonujący inne zadania. Jest odpływ fachowców. Musimy im dobrze zapłacić.

To jest zdecydowanie za mało i oni są słabo opłacani. Chcemy im dać lepsze możliwości pracy, lepszy sprzęt, lepsze siedziby, lepsze warunki, lepszą strukturę. Chciałem podkreślić, że ci policjanci, którzy nie przejdą weryfikacji, zostaną w strukturach Policji i będą wykonywali inne zadania służbowe. Nikt nie zostanie zwolniony z Policji, dlatego że nie dostał się z wydziału zwalczania cyberprzestępczości do CBZC. Potrzebujemy cały czas policjantów, mamy deficyty w tym zakresie, liczba wakatów maleje, ale jeszcze trochę ich zostało. Szanowni Państwo! Pan poseł Gawkowski pytał, dlaczego nie stworzymy nowej służby. Dlatego że to ma być. Ustawa o cyberbezpieczeństwie dzieli jak gdyby cały ten porządek cyberbezpieczeństwa na trzy części: wojsko - zajmuje się tym MON, sfera gov, rządowa - którą zajmuje się CERT i generalnie ABW, i NASK - który zajmuje się pozostałymi użytkownikami Internetu, których jest najwięcej. Ale NASK nie ściga. NASK zabezpiecza, NASK może edukować, ale nie ściga. Dlatego uważamy, że potrzebna jest służba, która będzie chroniła nie instytucje rządowe, nie Sejm, ale właśnie szarych obywateli. Dlatego jest to Policja.

Podjęliśmy taką decyzję, patrząc także na doświadczenia Centralnego Biura Śledczego.

Chciałbym natomiast odnieść się do jednego wystąpienia w sposób krytyczny. Panie pośle Frysztak, nie można w wystąpieniu klubowym proponować, żeby ściganiem cyberprzestępczości na poziomie obywateli zajmował się wywiad wojskowy. Jak pan widzi ściganie przestępczości przez wywiad? To jest po prostu śmieszne. Chciałbym podkreślić, że to nie jest służba przeciwko komuś. To jest służba dla obywateli, dlatego chcemy, żeby to była Policja. Widzimy - jest o tym mowa w uzasadnianiu ustawy - jak bardzo rośnie cyberprzestępczość na poziomie szarych obywateli.

Musimy mieć służbę, która im pomoże. Bardzo proszę wszystkich państwa posłów, którzy mają wątpliwości, o zgłaszanie ich w komisjach. Jesteśmy otwarci, będziemy na ten temat rozmawiać. Jesteśmy przekonani, że jesteśmy w stanie was przekonać, ewentualnie przyjąć wasze uwagi i poprawki do tego projektu, żeby był on jak najlepszy. Dziękuję, panie ministrze. Pół minuty, dobrze? Panie Ministrze! To, co pan powiedział, jest zaprzeczeniem tego, co powiedziałem ja.

Trzeba jasno powiedzieć, że to w żaden sposób nie będzie poprawiało koordynacji.

Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Do głosowania nad tym wnioskiem przystąpimy w bloku głosowań. Dziękuję.

Wznawiam obrady. Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych, druk nr 1771. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego wniosku. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o uchwałach Senatu w sprawie ustaw: - o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, - o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, - o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, - o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Sprawozdania to odpowiednio druki nr 1770, 1738, 1750 i 1751. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o uchwałach Senatu w sprawie ustaw: - o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, - o zmianie ustawy o ochronie gruntów leśnych i rolnych, - o rodzinnym kapitale opiekuńczym, - o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, - o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, - o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Sprawozdania to odpowiednio druki nr 1757, 1773, 1746, 1749, 1752 i 1735. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań. Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Proszę bardzo, pan poseł Borys Budka, Koalicja Obywatelska, wniosek formalny. Wysoki Sejmie! Wnoszę o przerwę 2-godzinną w celu przygotowania przez ministra zdrowia i premiera Morawieckiego kompleksowej informacji na temat strategii rządu w walce z COVID-em. Polacy czują się zagrożeni, Polacy czują już nie tylko drożyznę, ale także olbrzymi lęk przed tym, że ta fala będzie coraz większa. Czym wy się zajmujecie? Po raz kolejny tylko roszadami wewnętrznymi, tym, jak zapewnić sobie większość w parlamencie, a Polaków zostawiacie samym sobie. 25 tys. zachorowań dzisiaj. Blisko 500 zgonów. To jest efekt braku polityki waszego rządu. Nie robicie nic.

Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1753. W dodatkowym sprawozdaniu komisje przedstawiają poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Komisje wnoszą o ich odrzucenie. Ich przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 8. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 3., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 8., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Działa? Działa.

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa w brzmieniu z druku nr 1753, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 15. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1756-A. Proszę pana posła Zdzisława Sipierę o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoki Sejmie! Dodatkowe sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw.

Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1756. Komisja przedstawia jednocześnie wnioski mniejszości oraz poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 1., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Działa? Działa, tak? Dobrze.

Sejm poprawkę odrzucił. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek mniejszości odrzucił. O co chodzi, przepraszam? Proszę państwa, ale to jest coś nieprawdopodobnego. Palcem jeszcze państwo pokażcie. Tak, ten brzydko się zachowuje, tamten krzyczy. Ludzie kochani. Dorośli ludzie. Naprawdę, to jest coś niebywałego.

Te zachowania, zwracanie uwagi naprawdę nie przystoją posłom na sali sejmowej. Przystępujemy do głosowania.

Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 2., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 3., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 4., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 7., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Przyjęcie tej propozycji spowoduje bezprzedmiotowość poprawek 8. i 11. Głosujemy. Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki odrzucił. Przyjęcie tej poprawki spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 10. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 12., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 13., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 14., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 6. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 7. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw w brzmieniu z druku nr 1756, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw. Powracamy do rozpatrzenia punktu 3. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022.

Wysoka Izbo! Pragnę przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022, druk nr 1708-A. Do projektu zgłoszono 13 poprawek. Poprawki od 1. do 4. oraz 11. uzyskały negatywną opinię komisji, pozostałe poprawki zostały przyjęte. Rekomenduję Wysokiej Izbie przyjęcie całego projektu ustawy wraz z poprawkami. Komisja przedstawia również poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 7. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. W 9. poprawce wnioskodawcy proponują, aby po art. 53 dodać nowy artykuł dotyczący możliwości zwiększenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 9. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

W 10. poprawce wnioskodawcy proponują, aby po art. 53 dodać nowy artykuł dotyczący przekazania w 2022 r. dotacji Instytutowi Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 10. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 13. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 w brzmieniu z druku nr 1708, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022. Powracamy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1748-A. Proszę pana posła Dariusza Olszewskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam wielką radość, a zarazem zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej dodatkowe sprawozdanie z druku nr 1748-A o rządowym projekcie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 r., druki nr 1727 i 1748. Szanowni Państwo! Podczas drugiego czytania zgłoszono 13 poprawek do wspomnianego przeze mnie projektu ustawy.

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wnoszą o przyjęcie w całości rządowego projektu ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 r. Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1748. Komisje przedstawiają również poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisje wnoszą o ich przyjęcie. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 9. i 10., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawki przyjął. 11. poprawka stała się bezprzedmiotowa. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 12. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 13. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku w brzmieniu z druku nr 1748, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 6. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1741-A. Proszę panią poseł Józefę Szczurek-Żelazko o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Komisja Zdrowia w dniu 17 listopada na posiedzeniu rozpatrzyła poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Zgłoszono 15 poprawek.

Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1741. Komisja przedstawia również wnioski mniejszości, a także w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Z poprawką tą łączy się 2. poprawka oraz tożsamy 2. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. poprawki i 5. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

za przyjęciem 7. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Z poprawką tą łączy się 9. poprawka. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 8. i 9., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Z poprawką tą łączą się 13. poprawka i tożsamy 8. wniosek mniejszości oraz 14. poprawka i tożsamy 9. wniosek mniejszości. Przyjęcie tych propozycji spowoduje bezprzedmiotowość poprawek 11. i 12. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 11. i 12., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawki przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 15. poprawki oraz 10. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1741, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Powracamy do rozpatrzenia punktu 7. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1737-A. Proszę pana posła Jerzego Maternę o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej mam zaszczyt przedstawić dodatkowe sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1731 i 1737. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na dzisiejszym posiedzeniu rozpatrzyła poprawki i rekomenduje przyjęcie trzech poprawek oraz przyjęcie w całości projektu ustawy. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1737. Komisja przedstawia również w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1737, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Powracamy do rozpatrzenia punktu 8. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1740-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Zdzisława Sipierę o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Dodatkowe sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. W drugim czytaniu wpłynęły cztery poprawki.

Komisja przedstawia w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Poprawki 2. i 3. zostały zgłoszone do art. 3 projektu ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1740, wraz z przyjętą poprawką, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 11. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1747-A. Składam dodatkowe sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. Podczas drugiego czytania w dniu wczorajszym zgłoszono pięć poprawek.

Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1747. Komisja przedstawia w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawki przyjął. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1747, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. Powracamy do rozpatrzenia punktu 13. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1739-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę panią poseł Annę Paluch o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! 16 listopada odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody.

Komisja w dniu dzisiejszym, czyli 17 listopada, przeanalizowała szczegółowo te poprawki i rekomenduje Wysokiej Izbie odrzucenie wszystkich pięciu poprawek.

Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1739. Komisja przedstawia również w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1739, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody. Powracamy do rozpatrzenia punktu 19. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskich projektach uchwał o solidarności w sprawie ochrony polskich granic oraz w sprawie politycznego oraz humanitarnego kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Przechodzimy do głosowania. Komisja wnosi o przyjęcie projektu uchwały z druku nr 1774. Zgłoszona poprawka została paniom i panom posłom doręczona do druku nr 1774. W poprawce wnioskodawcy proponują w akapicie czwartym skreślić zdanie trzecie. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania nad całością projektu uchwały. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu uchwały w brzmieniu z druku nr 1774, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Wniosek formalny, pan poseł Borys Bardzo dziękuję, pani marszałek. Bardzo proszę o zdjęcie głosowania nad poprawką, która w tej chwili jest przed nami. Doszło do rzeczy niedopuszczalnej. Ustawa dotyczy zmiany ustawy o Narodowym Banku Polskim, była powszechna zgoda dotycząca upoważnienia ministra sprawiedliwości do wydania odpowiedniego rozporządzenia. I w drugim czytaniu, tutaj na sali, Ministerstwo Sprawiedliwości zgłasza poprawkę wychodzącą absolutnie poza zakres ustawy, bo ministrowi sprawiedliwości już nie wystarcza Fundusz Sprawiedliwości, tylko dokłada jeszcze do tzw. funduszu więziennictwa ponad 10% z tego, co teraz jest. Ustawa, która nazywała się: ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim, i taką przedłożyliście.

Znowu was minister sprawiedliwości po prostu oszukuje, panie prezesie. Ma Fundusz Sprawiedliwości, a teraz jeszcze będzie.

Proszę bardzo o odpowiedź pana. To za waszych czasów praca dla więźniów. A my tą poprawką doprowadzamy do tego, że. praca dla więźniów się będzie rozwijała i jeszcze więźniowie będą mieli dzięki Polskiemu Ładowi podwyżkę. Także więc proszę Wysoką Izbę o poparcie.

Panie pośle, zwracam się do pana przewodniczącego Budki, nie mogę w ten sposób zdjąć tego głosowania. Powracamy do rozpatrzenia punktu 21. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim. Komisja wnosi o przyjęcie projektu ustawy z druku nr 1685. Zgłoszone poprawki zostały paniom i panom posłom doręczone do druku nr 1685. Przyjęcie tych poprawek spowoduje zmianę tytułu ustawy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki przyjął. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy. Powracamy do rozpatrzenia punktu 22. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu, który poddam pod głosowanie. Odrzucenie tego wniosku oznaczać będzie, że Sejm, zgodnie z propozycją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu, skierował ten projekt ustawy do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w druku nr 1742, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił, a tym samym skierował ten projekt ustawy do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 33. porządku dziennego: Informacja rządu w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i podejmowanych działań - głosowanie. Wobec propozycji przyjęcia przedstawionej informacji do wiadomości zgłoszono sprzeciw. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem do wiadomości informacji rządu w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i podejmowanych działań, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm informację przyjął do wiadomości. Przypominam, że Koło Parlamentarne Polska 2050 złożyło wniosek o uzupełnienie porządku dziennego o punkt obejmujący informację prezesa Rady Ministrów o powodach wstrzymania przez Komisję Europejską prac merytorycznych nad oceną polskiego Krajowego Planu Odbudowy oraz o zastrzeżeniach merytorycznych co do zawartości polskiego Krajowego Planu Odbudowy. W związku ze zbliżaniem się terminu, o którym mowa w art. 173 ust. 5 regulaminu Sejmu, poddam pod głosowanie wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. Przypominam, że zgodnie z art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu głosowanie to nie jest poprzedzone debatą ani zadawaniem pytań. Przystępujemy do głosowania w sprawie wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt obejmujący informację prezesa Rady Ministrów dotyczącą Krajowego Planu Odbudowy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek o uzupełnienie porządku dziennego odrzucił. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 34. porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Józefa Mackiewicza (druk nr 1734) Proszę wicemarszałek Sejmu panią Małgorzatę Kidawa-Błońską o przedstawienie uzasadnienia projektu uchwały. W październiku tego roku Sejm zgodnie ustanowił rok 2022 Rokiem Józefa Mackiewicza. Dyskusja była zgodna i tutaj nie było wątpliwości, jednak w projekcie tej uchwały pojawił się błąd i projekt prezydialny ten błąd koryguje. Dziękuję bardzo. Nikt się nie zgłasza. Proponuję, aby Sejm niezwłocznie przystąpił do drugiego czytania projektu uchwały. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w drugim czytaniu projektu uchwały? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały zawartego w druku nr 1734, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Józefa Mackiewicza. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 30. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1726 i 1752) Proszę panią poseł Katarzynę Czocharę o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić dodatkowe sprawozdanie połączonych Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1726. Marszałek Sejmu zgodnie z regulaminem Sejmu skierowała w dniu 8 listopada 2021 r. uchwałę Senatu w powyższej sprawie do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Zdrowia w celu rozpatrzenia.

Przypominam, że Sejm odrzuca poprawki Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Głosować będziemy nad wnioskami o odrzucenie poprawek Senatu.

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął.

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nikt nie był za, przeciw - 431, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1 - za, przeciw - 431, nikt się nie wstrzymał. W 20. poprawce do art. 16g ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Senat proponuje zmianę ust. 4. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął.

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

2 - za, przeciw - 431, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 23. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druki nr 1719 i 1757) Proszę pana posła Jerzego Małeckiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Panowie Premierzy! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie połączonych Komisji: Finansów Publicznych oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, druk nr 1719. Komisje: Finansów Publicznych oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi po rozpatrzeniu powyższej uchwały na posiedzeniu w dniu wczorajszym, tj. 16 listopada, rekomendują obie poprawki odrzucić.

Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego.

Głosujemy.

Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 24. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druki nr 1720 i 1770) Proszę pana posła Jana Dudę o przedstawienie sprawozdania komisji. Panowie Premierzy! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić Wysokiej Izbie sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Senat po rozpatrzeniu przyjętej przez Sejm ustawy zgłosił osiem poprawek. Połączone komisje po zapoznaniu się z poprawkami Senatu wszystkie poprawki Senatu opiniują pozytywnie i wnoszą o ich przyjęcie przez Wysoką Izbę. Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Łącznie z tą poprawką będziemy głosować nad poprawkami 6. i 7. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

1 - za, przeciw - 430, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Nikt nie był za, przeciw - 431, nikt się nie wstrzymał. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 3. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 4. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 5. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 8. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 25. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druki nr 1721 i 1773) Proszę pana posła Leszka Galembę o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, druk nr 1721. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po rozpatrzeniu powyższej uchwały na dzisiejszym posiedzeniu pozytywnie opiniuje cztery poprawki wniesione przez Senat. Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego.

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Nikt nie był za, przeciw - 430, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 4. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Nikt nie był za, przeciw - 432, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 26. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1723 i 1738) Proszę panią poseł Annę Paluch o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 54 ust. 1 regulaminu Sejmu, skierowała w dniu 3 listopada tego roku uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z druku nr 1723 do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu rozpatrzenia. Komisja tę uchwałę, zawierającą jedną poprawkę do wzmiankowanej ustawy, rozpatrzyła 15 listopada tego roku i rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie poprawki Senatu.

Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 27. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym (druki nr 1722 i 1746) Proszę panią poseł Urszulę Rusecką o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Składam sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Pani marszałek Sejmu skierowała w dniu 3 listopada 2021 r. uchwałę Senatu w powyższej sprawie do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia 13 poprawek senackich. Komisja w dniu 15 listopada rozpatrzyła te poprawki i wnosi do Wysokiej Izby o to, aby sześć poprawek przyjąć, a siedem poprawek odrzucić. Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

1 - za, przeciw - 431, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 4. i 9., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawki bezwzględną większością głosów. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 5. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 10. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 11. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Komisja wnosi o ich odrzucenie. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 12. i 13., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 28. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (druki nr 1725 i 1750) Proszę pana posła Aleksandra Mrówczyńskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, druk nr 1725.

Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 1. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 4. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 5. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 6. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 7. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 8. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 9. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 10. i 18., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 11. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 12. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 13. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

W 14. poprawce do art. 55 Senat proponuje m.in. skreślić ust. 4. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 14. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 15. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 16. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 17. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 31. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1717 i 1751) Proszę pana posła Patryka Wichra o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Komisji Zdrowia przedstawić sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1717. Szanowna pani marszałek stosowną decyzją skierowała do prac w Komisji Zdrowia niniejszą uchwałę. Komisja w dniu 16 listopada rozpatrywała jej treść.

Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 3. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 4. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 5. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 6. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 7. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 32. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druki nr 1718 i 1735) Proszę pana posła Aleksandra Mrówczyńskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Szanowna Pani Marszałek! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, druk nr 1718.

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosowało 430 posłów. Nikt nie był za, przeciw - 430, nikt się nie wstrzymał. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druki nr 1724 i 1749) Proszę pana posła Kazimierza Moskala o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Składam sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, druk nr 1724. Marszałek Sejmu skierowała w dniu 3 listopada 2021 r. uchwałę Senatu w powyższej sprawie do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w celu rozpatrzenia. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży po rozpatrzeniu powyższej uchwały na posiedzeniu 15 listopada 2021 r. wnosi, żeby Wysoki Sejm uchwałę Senatu odrzucił. Przypominam, że Sejm odrzuca uchwałę Senatu odrzucającą ustawę bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Głosować będziemy nad wnioskiem o odrzucenie uchwały Senatu.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem uchwały Senatu odrzucającej ustawę z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 35. porządku dziennego: Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 1771) Prezydium Sejmu na podstawie art. 20 ust. 1 regulaminu Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionych propozycji? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku w brzmieniu z druku nr 1771, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm podjął uchwałę w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny 42. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze wygłosić oświadczenie? Nikt się nie zgłasza. Listę posłów zgłoszonych do oświadczeń uważam zatem za zamkniętą.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu polskich melomanów i wszystkich mieszkańców Bydgoszczy zwracam się do pana wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, mecenasa sztuki i kultury z serdeczną prośbą o wsparcie budowy kampusu Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy dodatkową kwotą 140 mln zł, niezbędną do rozpoczęcia i zakończenia tej inwestycji, tak bardzo potrzebnej, jeżeli chodzi o polskie opery i filharmonie, a także w odniesieniu do promocji polskiej muzyki w Europie i na wszystkich kontynentach. Budowa kampusu akademickiego jest warunkiem koniecznym dla dalszej profesjonalnej działalności i rozwoju Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, a także dla twórczego wykorzystania potencjału kadry dydaktycznej, w której są tacy mistrzowie jak przewodnicząca jury 18. międzynarodowego konkursu chopinowskiego pani prof. Katarzyna Popowa-Zydroń, członkini jury konkursu pani prof. Ewa Pobłocka czy zwycięzca 15. konkursu chopinowskiego z roku 2005 pan prof. Rafał Blechacz. W tegorocznym konkursie chopinowskim w grupie 45 najlepszych młodych pianistów świata aż 7, czyli 15%, było studentami bydgoskiej akademii i podopiecznymi profesorów pracujących w Bydgoszczy. Na uczelni kształcą się studenci muzyczni ze wszystkich miast Polski, a także studenci z Chin i Korei Południowej. W listopadzie br. jubileusz 40-lecia działalności obchodził Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej, którego absolwenci śpiewają obecnie na scenach operowych i estradowych całego świata. Dzięki grającym i śpiewającym absolwentom i profesorom akademii sukcesy artystyczne święcą także instytucje, które współprowadzone są przez pana ministra kultury, czyli Opera Nova i Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy, a także orkiestry i chóry z innych miast Pomorza i Kujaw. W budżecie państwa na budowę kampusu akademii muzycznej zarezerwowano 290 mln zł, ale po otwarciu ofert przetargowych okazało się, że do zrealizowania budowy jest potrzebna kwota aż o 140 mln wyższa. W tej sytuacji jedynie pan premier jako minister kultury i dziedzictwa narodowego może spowodować zwiększenie budżetu na budowę kampusu akademii muzycznej.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Grzegorz Lorek, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Bo ni z tego, ni z owego mamy Polskę na pierwszego” - ten zgrabny wierszyk, którego autorstwo jest przypisywane samemu Józefowi Piłsudskiemu, bardzo trafnie oddaje atmosferę tamtego listopadowego dnia sprzed ponad 100 lat. Lekkie słowa, ale nikt lepiej nie wiedział niż ówczesny naczelnik państwa polskiego, ile odzyskanie owej Polski kosztowało jego samego i kilka wcześniejszych pokoleń Polaków. Nie wchodząc jednak w meandry ówczesnej polityki międzynarodowej i prawdziwe mistrzostwo gry dyplomatycznej takich polskich mężów stanu jak wspomniany Józef Piłsudski czy Roman Dmowski, warto wspomnieć, jak koniec tego konfliktu, zwanego wielką wojną, wyglądał w moim rodzinnym mieście. Piotrków Trybunalski był jednym z ważniejszych ośrodków niepodległościowych na ziemiach polskich. Znajdujące się wówczas pod austro-węgierską okupacją miasto stało się ważne, dlatego że władze okupacyjne zezwoliły na oficjalną działalność polskich organizacji patriotycznych. Tutaj działały punkty werbunkowe Legionów Polskich tworzące zalążki późniejszych Polskich Sił Zbrojnych, tutaj też działało harcerstwo, które rekrutowało wśród swoich szeregów wielu żołnierzy. Miasto było też potężnym ośrodkiem wydawniczym, w którym drukowano tysiące publikacji patriotycznych, ale także literaturę naukową, choćby z zakresu historii Polski. Na ulicach Piotrkowa Trybunalskiego można było spotkać Władysława Sikorskiego, Juliusza Kadena-Bandrowskiego, Józefa Becka i wielu innych. Obok oficjalnej działalności zdawano sobie sprawę, że kiedyś trzeba będzie stanąć do walki. Aktywnie działała konspiracja Polskiej Organizacji Wojskowej, Sokoła i wielu innych. Uznano, że należy przejąć inicjatywę, gdyż okupującym ziemie polskie państwom centralnym, mówiąc kolokwialnie, nie wiodło się najlepiej. W Niemczech i na terenach monarchii c.k. wybuchały niepokoje, które przeradzały się w rewolucję. Okupanci byli słabi. Atmosfera była sprzyjająca, tym bardziej że do Piotrkowa docierały plotki o masowych rozbrojeniach Austriaków w Krakowie. W Piotrkowie Trybunalskim pierwszy oddział, który złożył przysięgę na wierność Polsce, utworzył mjr Brezany, będący najprawdopodobniej jednym z oficerów organów werbunkowych. W mieście stacjonowały dość poważne siły okupacyjne. Mimo to zdecydowano się rozpocząć akcję. Otoczono koszary wojskowe i po pertraktacjach udało się wynegocjować złożenie broni. Nakazano Austriakom opuszczenie miasta w ciągu 4 dni. Major Brezany 5 listopada wydał zarządzenie o obowiązku zachowania spokoju w czasie wycofywania się wojsk austriackich. Nie ma wielkiej historii bez małych wydarzeń. Przejęcie władzy w moim mieście odbywało się bez spektakularnych walk, ale może to i dobrze.

Bardzo proszę, pani poseł Monika Falej, Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przez ostatnie tygodnie byliśmy świadkami, jak posłowie PiS, ministrowie, a nawet sam pan premier jeździli po kraju i rozdawali pieniądze, a raczej kartoniki z cyferkami, bo na razie tyle warte są czeki Morawieckiego przekazywane w ramach inwestycji strategicznych Polskiego Ładu. Pieniądze, które miały trafić do Polski z Unii Europejskiej, nie trafiły i być może w ogóle do Polski nie trafią. Cierpimy my wszyscy.

Samorządy ciężko pracowały na te pieniądze i wciąż na nie czekają. Wzywam pana, by zaczął pan respektować europejskie prawo, by nie szedł pan na wojnę ze wspólnotą samorządową, którą sami tworzymy. Czas się opamiętać. Bardzo proszę, pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050.

Bardzo dziękuję. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Pragnę wyrazić stanowczy sprzeciw wobec planowanej likwidacji Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej jako samodzielnego podmiotu.

Oczywistym skutkiem tej decyzji będzie to, że bielsko-bialska izba pozbawiona zostanie niezależności w podejmowaniu decyzji. Tymczasem to właśnie ta izba działająca od wielu, wielu lat, od kilkudziesięciu lat, najlepiej zna potrzeby lokalnej przedsiębiorczości i najlepiej reprezentuje interesy lokalnej przedsiębiorczości zarówno w otoczeniu zewnętrznym, jak i na Podbeskidziu. Reprezentuje ona przedsiębiorców w kontaktach z miejscowym samorządem. Ważnym aspektem jest również fakt, że izba jest w bardzo dobrej kondycji finansowej i posiada znaczący majątek. I ten majątek, który został wypracowany przez izbę, przez bielskich przedsiębiorców, będzie przekazany do centrali w Katowicach. Takie działanie jest absolutnie niedopuszczalne i szkodliwe zarówno dla lokalnej przedsiębiorczości, jak i dla przedsiębiorczości w ogóle. Szanowni Państwo! W trosce o zachowanie aktualnego statusu Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej jako ważnego podmiotu dla południowego subregionu województwa śląskiego i tej części historycznej Małopolski zwracam się dzisiaj do pana ministra o niedopuszczenie do likwidacji samodzielności izby w Bielsku Białej. Składam również na ręce pana ministra właściwego do spraw gospodarki interpelację w tej sprawie, licząc na to, że te złe zmiany, złe decyzje zostaną zatrzymane i rząd nie przyczyni się do tego, że ten ważny organ przedsiębiorców, ta ważna reprezentacja przedsiębiorców zostanie zlikwidowana, ponieważ dobrze służy ona naszym przedsiębiorcom i naszemu regionowi. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W dniu 4 października miało miejsce bardzo ważne wydarzenie dla Wojska Polskiego, uczelni wojskowych, ale i społeczności miasta Dęblina. Stacjonująca w Dęblinie Lotnicza Akademia Wojskowa otrzymała nowy sztandar. Uroczystość odbyła się na placu przed pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt. W trakcie uroczystego apelu miała miejsce ceremonia odczytania aktu ufundowania sztandaru przez przedstawicielkę społecznego komitetu fundatorów, burmistrz Dęblina panią Beatę Siedlecką. Pełniła ona również jakże zaszczytną funkcję matki chrzestnej. Sztandar został przekazany na ręce rektora-komendanta gen. pilota Krzysztofa Cura. Jak powiedział komendant-rektor: „Dęblińska Szkoła Orląt jest uczelnią kształcącą kandydatów na żołnierzy zawodowych w Siłach Zbrojnych oraz studentów studiów cywilnych w trudnej, ale i satysfakcjonującej dziedzinie - lotnictwie. Aktualnie uczelnia prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne, studia podyplomowe, kursy doskonalenia zawodowego oraz kursy kwalifikacyjne na kolejny stopień wojskowy. W związku z modernizacją wojska przed uczelnią postawione zostały nowe cele i wyzwania. Zachęcam do zapoznania się z bogatą ofertą Lotniczej Akademii Wojskowej. Niełatwo znaleźć uczelnię o podobnych możliwościach - nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Szkoła Orląt to miejsce, które pozwala realizować marzenia pośród ludzi wywodzących się ze środowiska wojskowego, jak i cywilnego, których łączą wspólne zainteresowania i pasja do lotnictwa od wielu lat” W związku z powyższym trochę historii. W wyniku zaplanowanej wieloletniej rozbudowy Szkoła Orląt stała się jedną z najnowocześniejszych szkół lotniczych na świecie. Na liście wybitnych absolwentów figuruje m.in. Zdzisław Krasnodębski, urodzony w Woli Osowińskiej w gminie Borki w powiecie radzyńskim, wnuk powstańca styczniowego i zesłańca na Sybir, ale także pierwszy dowódca 303. Dywizjonu Myśliwskiego. Wychowankami byli również piloci Walerian Jesionowski, dowódca 308. Dywizjonu Myśliwskiego, Stefan Łaszkiewicz, pierwszy dowódca tegoż dywizjonu, czy w końcu Stanisław Skalski, as myśliwski z okresu drugiej wojny światowej o największej liczbie zestrzeleń wśród polskich pilotów. Jeśli chcemy poznać trochę bliżej historię polskiego lotnictwa, to gorąco zachęcam, szczególnie młodzież, do odwiedzenia Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie właśnie. Najważniejszym eksponatem jest niewątpliwie relikwia - sztandar Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie z okresu drugiej wojny światowej. Zobaczymy też zrekonstruowany domek pilota z czasu bitwy o Anglię, umundurowanie i pamiątki nawiązujące do słynnego dywizjonu 303. Wystawa plenerowa to ponad 80 statków powietrznych. W tych listopadowych dniach pamiętajmy o bohaterskich polskich lotnikach, z których wielu oddało swoje życie w obronie ojczyzny, zgodnie z maksymą, także Lotniczej Akademii Wojskowej, „Pro patria semper” - „Zawsze dla ojczyzny” Mam i ja swoje związki z lotnictwem. Od początku tej kadencji zasiadam na miejscu nr 303. Wobec tego czuję się zobowiązany do poświęcenia większej uwagi „stolicy polskich skrzydeł” - miastu Dęblin. Bardzo proszę, pan poseł Jacek Kurzępa, Prawo i Sprawiedliwość.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Drodzy Lubuszanie! Kontynuuję wraz z wami wędrówkę poparcia dla polskich żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej, wszystkich innych formacji, które bronią teraz granicy. Pozwólcie, że pierwszy akapit zaadresuję do pani por. Anny Michalskiej, rzecznik prasowej Straży Granicznej. Jest pani dzielną i twardą kobietą oraz profesjonalną funkcjonariuszką. Trzymam za panią kciuki. Aniu, wytrwaj, gdyż jesteś wybitna. Po raz kolejny my, Lubuszanie, spotkamy się jutro w ramach akcji „Murem za polskim mundurem” tym razem w Międzyrzeczu w pobliżu muzeum międzyrzeckiego w okolicy pomnika gen. brygady Józefa Dowbor-Muśnickiego, wielkiego dowódcy powstania wielkopolskiego. Zapraszam Lubuszan na godz. 14, by właśnie tam wspólnie w spontanicznym odruchu serc przesłać wyrazy wdzięczności dla wszystkich broniących obecnie naszych granic. Adresujemy swoje myśli do żołnierzy 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, oddając także hołd Krystianowi, ufając, że uda się uniknąć wszelkich podobnych tragedii. Drodzy mieszkańcy Międzyrzecza, przybywajcie. Weźcie ze sobą biało-czerwone flagi, bądźcie gotowi wraz ze wspólnotą tych, którzy się tam zgromadzą, żeby odśpiewać a cappella hymn państwowy, a później „Rotę”

Wracając do tych dwóch miejsc, dziękuję samorządowcom, którzy bez względu na polityczne rodowody towarzyszyli nam w tych wiecach, oraz dziękuję za ich logistyczną pomoc przy ich organizowaniu. Dziękuję burmistrzowi Żagania, Andrzejowi Katarzyńcowi, wójtom gminy wiejskiej Żagań - Leszkowi Ochrymczukowi, gminy Wymiarki - Lechowi Miszewskiemu, radnym powiatowym i miejskim powiatu żagańskiego, żarskiego, mieszkańcom tych miejscowości, zespołom śpiewaczym „Mała Tęcza” i „Złoty Kłos” za to, że byliście, uświetniliście i wsparliście. Dziękuję burmistrzowi Krosna Odrzańskiego, Markowi Cebuli, staroście krośnieńskiemu, Grzegorzowi Garczyńskiemu, radnym z tego terenu, Wojciechowi Brudzińskiemu, mieszkańcom Krosna Odrzańskiego i okolic. Dziękuję pani staroście międzyrzeckiej, Agnieszce Olender, dyrektorowi muzeum międzyrzeckiego, Andrzejowi Kirmielowi, społecznikom związanym z lokalną grupą rybacką Obra - Warta, leśnikom, mieszkańcom w ogóle, tym, którzy zechcą jutro, a wcześniej w wymienionych miastach: Żagań, Krosno, wspólnie oddać swój czas i swoje serce tym, którzy dzisiaj bronią naszej ojczyzny. Dziękuję również tym, którzy na rozlicznych portalach internetowych, wirtualnych komunikatorach pomnożą nasz gest solidarności i wsparcia skierowany do żołnierzy 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej i wszystkich innych jednostek, i formacji, i służb, które teraz bronią granicy. Niech wracają cali i zdrowi. Niech strzeże ich opatrzność, a nas niech strzegą oni. Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Waldemar Andzel, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować organizatorom, a przede wszystkim uczestnikom tegorocznego Marszu Niepodległości. Nadanie temu wydarzeniu charakteru państwowego było bardzo dobrym posunięciem, za co również dziękuję. Intencją wszystkich uczestników była nie tylko pamięć o walce Polski o niepodległość, ale przede wszystkim była nią troska i szacunek dla polskiego munduru. Intencja ta pozwoliła oddać hołd funkcjonariuszom Straży Granicznej, policjantom, żołnierzom zawodowym i Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy dbają o bezpieczeństwo Polski i Unii Europejskiej na wschodniej granicy. Jesteście naszymi bohaterami. Wsparcie dla polskiego munduru jest ważne, szczególnie dzisiaj, kiedy bezpieczeństwo polskiej granicy jest brutalnie naruszane. Polskie służby zostały zmuszone do użycia armatek wodnych, a jeden z policjantów został poważnie ranny. Międzynarodowa opinia nie ma wątpliwości, że jest to kryzys polityczny mający na celu destabilizację Unii Europejskiej. Reżim Łukaszenki organizuje międzynarodowy handel ludźmi. Zrozumieli to już wszyscy w Europie poza totalną opozycją polskiego rządu. Na szczęście póki rządzi Prawo i Sprawiedliwość nie ma mowy o jakimkolwiek szlaku migracyjnym wiodącym przez Polskę do Europy Zachodniej. Będziemy wzmacniać granicę, budować mur i stale reagować. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Tomasz Głogowski, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie!

Na powtarzane kilkukrotnie pytanie, dlaczego tak rząd boi się dopuszczenia dziennikarzy do strefy stanu wyjątkowego, odpowiedział, że Ameryka przegrała wojnę w Wietnamie, dlatego że byli w Wietnamie na miejscu dziennikarze. Przekazywali to, co się działo, to, co nie spodobało się wyborcom amerykańskim, obywatelom amerykańskim. A więc domyślam się, że premier uważa, że dziennikarze pokazywaliby sytuacje, które by się wyborcom nie podobały.

Przyznam, że kiedy to przeczytałem, uznałem, że już przesadzono, że ktoś, kto nie lubi rządu, przesadził z tak nieprawdziwą informacją.

Dzisiaj, przed chwilą Sejm uchwalił kolejną ustawę, która odbiera wolności obywatelom, ustawę nazwaną trochę mylnie: o obronie granicy. Ona niczego nie zmienia dla uchodźców, dla tych, którzy chcą się wedrzeć na granicę. Służby państwowe powinny bronić granicy bez względu na to, czy jest stan wojenny lub wyjątkowy. Ustawa zabiera tylko wolności obywatelom. Zabiera obywatelom polskim podstawowe wolności, takie jak prawo do swobodnego poruszania się po terenie ojczyzny, wolność prowadzenia działalności gospodarczej, prawo do dostępu do informacji.

Jeżeli Niemcy szacują liczbę emigrantów, o których wiedzą, którzy się zgłosili do obozów, na 8, 9, 10 tys. - tych, którzy przeszli przez Białoruś, a z Białorusi przez Polskę do Niemiec. Pan minister Kamiński mówił parę dni temu, że oni prawdopodobnie w olbrzymiej większości znaleźli się w Polsce przez Litwę.

W tej chwili opinia światowa ma tylko przekaz ze strony dziennikarzy wpuszczonych przez Łukaszenkę do tych miejsc, do których zgodził się ich wpuścić. Nie ma możliwości zweryfikowania tego przez dziennikarzy z drugiej strony.

Gdyby mieli w tej telewizji codziennie przekazywać, że ta granica nie jest otwarta, jak przekonują ich opłacani przez Łukaszenkę i Putina przemytnicy, to pewnie wielu z nich nie zdecydowałoby się na podróż.

Wysoka Izbo! Od chwili, w której zostałem posłem na Sejm RP, z dumą i rzetelnością realizuję swoje obowiązki, gdyż wiem, że jako reprezentant moich wyborców muszę uczciwie, z pełnym zaangażowaniem prowadzić działania, które rozwiązują ich problemy i zaspokajają potrzeby. Mam już swoje lata. Znam życie z najbardziej trudnych i ciężkich jego stron. Jestem na emeryturze, po 45 latach pracy w branży górniczej. Mówię to dlatego, że jeżeli ktoś myśli, że to, co robię jako poseł, wykonuję dla kariery lub innych osobistych czy rodzinnych celów, to jest w wielkim błędzie. Przez całe życie kierowałem się uczciwością i solidnością inżynierską.

W związku z tym nie mogę milczeć. Twórcy wymienionego przeze mnie reportażu w jednej półgodzinnej audycji zmieszali ze sobą szkodliwe społecznie, niezgodne z prawem działania dawnych władz samorządowych gminy Bogatynia, sprawę osuwiska, które miało miejsce w kopalni w 2016 r., oraz kwestię negocjacji z Czechami w kontekście wyroku TSUE. W czasie udzielania wywiadu do reportażu zostałem zaskoczony jego formułą i atakiem na mnie.

Przykro mi, że redaktorzy TVN nakłaniani są do ukazywania spraw w tak nieprofesjonalny i nieobiektywny sposób. Dlaczego nie wznieśli się na wyżyny obiektywnej, sprawiedliwej oceny zaistniałych zdarzeń? Dlaczego wybrano pseudoeksperta do wypowiadania się w sprawach związanych z osuwiskiem w kopalni Turów? Dlaczego nie zadali sobie trudu, aby zapoznać się z opinią Wyższego Urzędu Górniczego, protokołem końcowym komisji w spółce PGE GiEK oraz ekspertyzami niezależnych specjalistów oceniających przyczyny i skutki osuwiska w kopalni Turów? Dlaczego nie zadali sobie trudu, aby porównać to zdarzenie z podobnymi przypadkami zaistniałymi w innych znanych kopalniach odkrywkowych? Dlaczego nie zadali sobie trudu, aby stwierdzić, że mój syn ma 27-letnie doświadczenie w pracy górniczej, posiada zatwierdzenie Okręgowego Urzędu Górniczego do pełnienia funkcji kierownika ruchu zakładu górniczego oraz ma niezbędne wykształcenie? Członkiem Rady Nadzorczej spółki PGE GiEK został nie przez nepotyzm, ale w wyniku wyboru przez kilkunastotysięczną załogę tego koncernu. Jego nieszczęściem, oczywiście w cudzysłowie, jest to, że ma ojca, który jest obecnie posłem na Sejm RP. Jestem przekonany, że nie jest to ostatni reportaż stacji TVN atakujący ludzi, którzy bronią niezależności energetycznej Polski. Celem jest także wywołanie społecznego przyzwolenia na likwidację polskiego przemysłu węgla kamiennego i brunatnego. Trwają negocjacje z Czechami w sprawie Turowa. Zniekształcenie rzeczywistości w tym reportażu na pewno nam nie pomoże. Zwracam uwagę wszystkich posłów na tej sali na jedną rzecz: dzisiaj celem jestem ja, jutro może być każdy z was bez względu na przynależność partyjną. Pragnę oświadczyć, że jako poseł na Sejm RP nie zgadzam się z takim traktowaniem tej sprawy i dalej będę podejmował działania, aby zmiany w funkcjonowaniu górnictwa, energetyce polskiej zapewniały naszemu krajowi bezpieczeństwo i niezależność energetyczną. Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Aleksander Mrówczyński, Prawo i Sprawiedliwość.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Słowa te powinny być drogowskazem każdego Polaka. Naszym obowiązkiem jest pamięć o poprzednich pokoleniach, o czasach minionych, wspaniałych i dramatycznych dla naszej ojczyzny. Ze wspaniałych momentów historii Polski musimy być dumni, z trudnych i ciężkich - wyciągać wnioski. Słowa amerykańskiego poety i filozofa George’a Santayany: kto nie pamięta historii, skazany jest na jej ponowne przeżycie, doskonale komponują się ze słowami marszałka Piłsudskiego - pamięć o przeszłości jest kluczowa dla każdego człowieka, narodu.

Wspominamy powstańców insurekcji kościuszkowskiej, powstań: listopadowego, styczniowego, wielkopolskiego, śląskiego. Ofiara ich krwi przyczyniła się do odzyskania niepodległości. Wspominamy ofiary, wcielonych do zaborczych armii podczas wielkiej wojny, chylimy czoła przed obrońcami II RP w czasie sowieckiego ataku w 1920 r.

Blisko naszej pamięci są harcerze Szarych Szeregów, partyzanci Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, wspaniali młodzi ludzie, którzy oddali życie w powstaniu warszawskim. Pamiętamy o tragicznych losach żołnierzy 2. korpusu gen. Władysława Andersa, dla których nie było powrotu do Polski po II wojnie światowej. Wzorem dla wszystkich powinni być żołnierze niezłomni, wyklęci przez komunistyczny terror przyniesiony na bagnetach Armii Czerwonej.

W naszej pamięci są ofiary robotniczych strajków w Poznaniu, na Wybrzeżu, w Radomiu i w kopalni Wujek.

Te setki tysięcy zesłańców, katorżników, więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i sowieckich łagrów, więźniów politycznych PRL-u, internowanych, szykanowanych w czasie tzw. demokracji ludowej, wszystkich ich łączyło jedno - miłość do naszej ojczyzny, do Polski. Polska jest matką szczególną, niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej - te słowa naszego ukochanego św. Jana Pawła II idealnie oddają pobudki, jakimi kierowały się poprzednie pokolenia naszych rodaków. Miłość do ojczyzny, miłość szczególna, warta każdej ofiary, nawet ofiary życia. Nic nie jest wieczne ani dane raz na zawsze - niech te słowa każdy z nas pamięta, aby zachować świadomość o tym, że każdego dnia musimy budować, wzmacniać, dbać o naszą wspólną Rzeczpospolitą Polską. Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Tomasz Olichwer, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym uświadomić państwu, jak wygląda zapewnienie bezpieczeństwa i dbanie o zdrowie obywateli, którzy zaszczepili się przeciw COVID-19. Obecnie przy podejrzeniu ponownego zachorowania odmawia się takim osobom wykonania u nich testów. Tak zwani poprawni obywatele zaszczepili się, w związku z tym nie tylko zmniejszyli ryzyko większych powikłań podczas choroby, ale również zmniejszają koszty związane z leczeniem ponoszone przez państwo. A co za to mają? Są żołnierzami do pracy, którym nie wykonuje się testów, bo szkoda na ten cel środków finansowych, bo zawyżają statystyki osób zarażonych, bo prawdziwe wyniki pokażą nieudolność naszego kraju w walce z COVID-19? Nasuwa się również pytanie, czy dokładne sprawdzenie stanu zdrowia przez wykonanie testu na COVID-19 osobie zaszczepionej to przywilej, czy też raczej zaniedbanie. Czy ktoś z rządu panuje nad tą sytuacją? Przypominam, że osoby zaszczepione dalej mogą chorować i zarażać innych. To, co się obecnie dzieje, nie ma nic wspólnego z opanowaniem sytuacji, a wręcz jest fałszowaniem jej. Dlatego nie mogę przejść obok tego obojętnie. W związku z tym apeluję również z tego miejsca o rozwagę i zapewnienie Polakom przemyślanego bezpieczeństwa podczas pandemii. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! 14 listopada to Światowy Dzień Seniora, okazja do życzeń i podziękowań za aktywność seniorów, ale również do rozmów o ich roli i ich obecności w różnych sferach naszego życia społecznego. Starzenie się jest naturalnym procesem i każdy z nas prędzej czy później doświadczy tego etapu życia. Dlatego niezwykle ważne jest, by wszelkie działania, inicjatywy o zasięgu lokalnym czy ogólnopolskim zwracały uwagę społeczeństwa na problemy, z jakimi zmagają się seniorzy. To nie tylko problemy zdrowotne czy ekonomiczne, lecz przede wszystkim samotność i odizolowanie, które ze względu na panującą pandemię drastycznie się zwiększyły. Pamiętajmy, że pomimo wieku osoby starsze nadal stanowią pod różnymi względami bardzo aktywną część społeczeństwa, dzięki której prężnie rozwija się działalność organizacji pozarządowych, np. upowszechniających wiedzę, religijnych czy promujących konkretne zainteresowania. Seniorzy bardzo chętnie biorą udział w wolontariacie, współpracują z samorządem lokalnym. Należy zauważyć, iż tzw. aktywność nieformalna na rzecz rodziny przynosi długofalowe i zakrojone na szeroką skalę korzyści. Wypełniając rolę dziadków, często zapewniają opiekę wnukom i przekazują wiedzę niezbędną do odkrywania świata. Jest to niezwykle istotny fakt, gdyż pokazuje, jak ważna dla funkcjonowania seniorów jest właśnie integracja pokoleniowa. Angażując osoby starsze w różnego rodzaju akcje i projekty, pokazujemy im, że są nadal dla nas ważne, a ich działania często są niezbędne. Każdy z nas ma w swoim najbliższym otoczeniu osoby w podeszłym wieku, które wymagają specjalnej opieki i szczególnego zainteresowania zarówno ze strony rodziny, jak i społeczeństwa. Jesteśmy im to winni jako wyraz naszej wdzięczności zarówno za dar życia, wychowanie, kształtowanie systemu wartości, jak i przekazanie wiary, poszanowania dla zasad, kultury i tradycji. Niech ten dzień poświęcony seniorom na całym świecie pobudzi także nas, parlamentarzystów, oraz całe społeczeństwo do zastanowienia się nad tym, jakie rozwiązania systemowe możemy jeszcze wprowadzić, by ułatwić osobom starszym funkcjonowanie w dzisiejszej rzeczywistości. Bardzo proszę, pani poseł Elżbieta Duda, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Kilka dni temu obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Przy tej okazji chciałabym poruszyć problem edukacji patriotycznej.

Informacja o wpływie interpelacji, zapytań oraz odpowiedzi na nie dostępna jest w Systemie Informacyjnym Sejmu. Na tym kończymy 42. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Protokół posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w Sekretariacie Posiedzeń Sejmu.